rynek pracy w tej chwili, pomimo bardzo ciemnych prognoz, które były po drugim kwartale tego roku, prawdopodobnie zamkniemy wskaźnikiem bezrobocia 6,1% w roku 2020. Dalej, proszę państwa, jeżeli chodzi o wyniki przedsiębiorstw, są one oczywiście gorsze, jest niższa rentowność. Są oczywiście sektory, gdzie rentowność nawet wzrosła i jest wyraźnie powyżej stopy zwrotu z innych inwestycji, które oferuje rynek, natomiast co warto podkreślić, poprawiły się wskaźniki płynności w gospodarce. I to jest optymistyczna wiadomość, bo firmy zazwyczaj upadają nie dlatego, że mają straty, ale dlatego, że tracą płynność. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, obserwujemy, że nie ma załamania, jeżeli chodzi o wycofywanie się z działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej pokazuje w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 16%, jednak liczba wniosków o wznowienie działalności wzrasta. Można powiedzieć, że w bieżącym roku złożono o 17% wniosków mniej w porównaniu z okresem ubiegłorocznym, ale spadła też liczba firm kończących działalność. Tych danych jest oczywiście, drodzy państwo, znacznie więcej, natomiast syntetyczny obraz, jeżeli chodzi o prognozy gospodarcze na przyszły rok, w mojej ocenie - to jest mniej może istotne, ale również w ocenie ośrodków analitycznych polskich i zagranicznych - jest pozytywny. Jeżeli nie dojdzie do innych niespodziewanych zdarzeń, czeka nas wzrost pozwalający uzyskać poziom roku 2019. Przepraszam, że tak syntetycznie. Dziękuję, panie ministrze. Chciałem panu powiedzieć, że poszło panu całkiem dobrze jak na pierwszy raz, więc może pan dzisiaj spać spokojnie. Proszę państwa, mam taki dylemat, którym się z państwem podzielę. Dobrze, ale zanim pani pokrzyczy, pani poseł, to niech pani posłucha. Jest 41 osób zgłoszonych do dyskusji.

Jak wiecie, ja nie przerywam, ale będziecie mieli przynamniej taki liczniczek, który będzie wam pokazywał, że trzeba iść do brzegu. Dobrze? Proszę bardzo, pani poseł. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani poseł z Platformy zamierzała prawdopodobnie w swoim wystąpieniu zdyskredytować działania rządu, ale dowiodła raczej, że były one szybkie i wymierne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji światowej pandemii najszybciej, jak było to możliwe, przygotował instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców, dla pracodawców i pracowników. Skuteczność działań rządu potwierdzają twarde dane. Do polskich firm trafiło do tej pory ponad 165 mld zł. Udało się uchronić również 6 mln miejsc pracy.

Przygotowane tarcze antykryzysowe i ich kolejne nowelizacje pozwoliły na udzielenie wsparcia wielu branżom. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał kolejny instrument tarczy w sprawie pomocy branżowej dla firm - tarczę 6.0. To wsparcie dla 40 branż i pomoc dla 270 tys. podmiotów. Przed nami kolejna tarcza opiewająca na 35 mld zł.

Panie Ministrze! Jak można ocenić skalę pomocy z tarcz antykryzysowych na tle innych krajów Unii Europejskiej w perspektywie [[Dzwonek]] możliwości finansowych Polski? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Targi książki, targi pracy, targi turystyczne, targi konserwatorów zabytków, targi zbrojeniowe - to polska marka. Zdobyliśmy rynek, byliśmy liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, promowaliśmy Polskę, polskich przedsiębiorców. Z dnia na dzień te firmy znalazły się w stanie agonii. Prawdopodobnie będą mogły normalnie funkcjonować dopiero na jesieni przyszłego roku - wiemy, jak długo trwa proces przygotowywania targów, a poza tym firmy, które mają wziąć udział w targach, także muszą zacząć normalnie funkcjonować. Do tego dochodzą branże powiązane, czyli hotele, cateringi, promocja, wydawcy. Tak naprawdę do września straty w tej branży wyniosły już 1 mld zł.

Rozmawiałam z przedstawicielami branży targowej. Nie wiem, czy państwo z rządu z nimi rozmawiają, ale jeżeli nie pomożemy tej branży, to będzie nie tylko upadek targów w Polsce, lecz także szansa na przejęcie ich przez firmy zagraniczne, [[Dzwonek]] które na to czekają. Już dawno minęło 21 dni. Nie dostałam odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Katarzyna Kretkowska, Klub Parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo!

W informacji bieżącej, w zagajeniu, był przywołany przypadek przedsiębiorcy z Wielkopolski, z Wrześni koło Poznania, który popełnił samobójstwo.

O taką pomoc klub Lewicy dopomina się od samego początku pandemii. Chodzi o proste narzędzia, które zostały uruchomione w Europie, a nie zostały uruchomione w Polsce.

Polscy przedsiębiorcy nie dostali podstawowej pomocy, tzn. pokrycia bądź zawieszenia kosztów stałych. Dlaczego przedsiębiorstwa wynajmujące powierzchnie (Dzwonek) w centrach handlowych dostały ustawowe zawieszenie płatności czynszu, a żadne inne przedsiębiorstwa takiego ustawowego zawieszenia płatności czynszu nie otrzymały?

Dziękuję.

Pani poseł Borowiak ze sprostowaniem. Proszę bardzo. Wysoki Sejmie! Szkoda, że pani poseł z Lewicy swoim głosem spowodowała to, że musimy zabrać w tym momencie czas przeznaczony dla kolejnych osób, które chciały panu ministrowi postawić pytanie. Pani poseł, nie mogę się nie odnieść do pani słów.

Pani poseł, jeżeli dla pani poseł z Lewicy ponad 165 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców, jeżeli dla pani poseł z Lewicy uratowanie 6 mln miejsc pracy to jest nic, to naprawdę serdecznie gratuluję.

Pani poseł, naprawdę, proszę zejść na ziemię i myśleć realnie. Dziękuję pani serdecznie. Myślę, że to jest tak, że jedna pani poseł ma taki pogląd w tej sprawie, a druga inny. Po to jest Sejm, żeby się tymi poglądami wymieniać. Pan poseł Dariusz Kurzawa, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Codziennie spotykam się z przedstawicielami branż eventowych, gastronomicznych czy turystycznych. Turystyka, chciałbym przypomnieć, to nie tylko Tatry, morze, ale także Kujawy z pięknym Gopłem, zabytki i atrakcje Strzelna, Inowrocławia, Bydgoszczy, Żnina, Kruszwicy, Tucholi. Średnie dochody branży turystycznej i gastronomicznej to obecnie zaledwie 10% wpływów sprzed pandemii. Mimo częściowego otwarcia galerii widać w nich, jak wiele sklepów jest likwidowanych.

Potrzebne są przede wszystkim - i apeluję tutaj o to - bezzwrotne środki pomocowe właśnie dla taksówkarzy, restauratorów, hotelarzy, branży eventowej, i to nie drobne 5 tys. zł, ale chodzi tu też o zaangażowanie środków unijnych, a także zwolnienie z podatków, ponieważ bez tej pomocy po prostu te branże nie przetrwają, a wygląda na to, że pandemia zostanie z nami jeszcze dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Urszulę Rusecką z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Miałam nadzieję na naprawdę merytoryczną dyskusję, ponieważ temat jest ważny i trudny. W związku z powyższym przysłuchałam się wypowiedzi pani sprawozdawcy, jak również pani marszałek, i dochodzę do wniosku, że państwo w ogóle nie znacie tej pomocy, która jest przez rząd Polski. To jest, przepraszam bardzo, w tarczy 6.0.

Skoro do rzeczy, to powiem tak: jeżeli chodzi o zarządzanie w sprawach kryzysu, rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę zdał egzamin.

Chciałem powiedzieć, że brałem udział w tych burdach wielokrotnie i. I mam uprzejmą prośbę, gdyż tak sobie Sejm wyobrażam, żebyśmy się wzajemnie nie obrażali. Ja uczestniczyłem w marszach kobiet walczących o swoje prawa, a nie w burdach ulicznych. Wysoka Izbo!

Wczoraj, proszę państwa, rozmawiałam z panią Izą z Wisły, która od 15 lat z powodzeniem prowadzi biznes apartamentowy. To prawda, może pani sprawdzić, podam pani wszystkie dane, proszę pani. Proszę państwa, wy nie tylko nie pomagacie, ale ten chaos, jaki panuje w tej pomocy... raz wedle PKD, gdzie 30, 40 branż wspieracie. Nie dostał żadnego wsparcia, a trzy razy miał kontrolę policji. Takie jest wsparcie dla branży turystycznej. Naprawdę ci ludzie błagają o pomoc.

Nie planuje się biznesu z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Chyba panie w życiu nie zarobiły złotówki na swoje konto, dlatego o tym pojęcia nie macie. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! liczbami, bo z tego, mówiąc krótko, polski przedsiębiorca nic nie ma. Prawda jest taka, że to jest wasz obowiązek, żeby dbać o polską gospodarkę, bo dzisiaj po prostu rządzicie. W związku z tym łaski nie robicie, że wprowadzacie różne mechanizmy, a ja zakładam, że dyskutujemy tutaj o tym, jak poprawić te mechanizmy, żeby one dotarły rzeczywiście do większej liczby przedsiębiorców. Zwracam uwagę, że gospodarka funkcjonuje tak, że to są naczynia połączone. Czyli, mówiąc krótko, jeżeli ktoś nie korzysta z restauracji czy one są zamknięte, czy nie korzysta z hotelu, to w związku z tym iluś usługobiorców tego hotelu również nie ma żadnych przychodów, a więc też jest pozbawionych możliwości funkcjonowania. W związku z tym dzisiaj w mojej ocenie, jeśli mówimy o tych wszystkich instrumentach, to błąd jest taki, że wybieramy sobie PKD w zależności od tego, kto tam głośniej krzyknie i powie, że nie ma środków finansowych. W związku z tym moje pytanie jest takie: Czy nie należy wykorzystać doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej i zastanowić się nad jedną prostą formułą pomocy, czyli, mówiąc krótko, wyrównaniem (Dzwonek) poziomu przychodów każdego przedsiębiorcy np. w wymiarze 70%, jak to jest we Francji czy w Niemczech, rok do roku.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Klimczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Proste rozwiązania są najlepsze, to jest stara maksyma - nie tylko stara, ale i sprawdzona. Dlaczego rząd nie spróbuje właśnie w taki sposób podejść do konstruowania kolejnych tarcz, szczególnie biorąc pod uwagę to, że kiedy ogłaszana jest pomoc z kolejnej tarczy, zgłaszają się nowe rodzaje działalności gospodarczej, które nie są w niej uwzględnione, a tym samym są poszkodowane.

Okazuje się, że one także nie są uwzględnione w tarczy pomocowej. Czy rząd nie myśli, żeby przejść do takiej prostej zasady, że pomoc należy się tym wszystkim działalnościom gospodarczym, które notują określoną stratę?

I naczelna zasada: żadnych nowych podatków do końca pandemii, a przynajmniej przez najbliższe 2 lata. Dziękuję serdecznie. Zapraszam uprzejmie. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Okres pandemii jest to taki czas, który objął cały glob. Właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie obiecując, a realizując, wprowadził tzw. wsparcie dla branży turystycznej i polskich rodzin, które w wyniku pandemii mogły utracić czy mieć zmniejszone wpływy budżetowe - wprowadził bon turystyczny. Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 500 zł, które otrzymuje każde dziecko do 18. roku życia i, dodatkowo, jeżeli jest dziecko. Szanowna pani, pani pozwoli, że nie będę z mównicy z panią polemizować, a pani, siedząc w ławach poselskich, ze mną.

Tym bonem można opłacać m.in. wypoczynek, zarówno pobyt w hotelu. Ale nie obowiązuje ten bon turystyczny tylko i wyłącznie w tym momencie. Proszę powiedzieć, czy bon [[Dzwonek]] jest realizowany? Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jestem zawiedziona na całej linii tym, co pan powiedział, bo pytania od ludzi z branży są zupełnie inne. Pan na żadne pytanie nie odpowiedział. Chcę powiedzieć, że branża turystyczna przynosi naszemu krajowi 7% produktu krajowego brutto. Prawie 1 mln mieszkańców, Polaków, żyje z tej branży. Bardzo ważna działalność. Tymczasem miejscowości turystyczne, gdzie głównym źródłem dochodów są usługi turystyczne, znalazły się w dramatycznej sytuacji. Od 3 miesięcy nie mają z czego zapłacić ZUS-u, kredytów, zapłacić pracownikom, zapłacić za energię i pokryć innych kosztów. Mówienie ciągle o tarczy nr 6 to naprawdę jest jakieś wielkie nieporozumienie. Ona nie załatwia tych problemów w żaden sposób. Ludzie chcą pracować. Sezon turystyczny daje, przynosi największe dochody. Takie miasto jak Karpacz straci w tym roku 200 mln zł, podobnie Szklarska Poręba i inne.

Kiedy rząd na to odpowie? To jest temat do dyskusji, a nie zasłanianie się dziurawą tarczą. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Zapraszam, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać o całą branżę agroturystyczną. Zapomnieliście o branży agroturystycznej w tej tarczy, kolejnej tarczy, wcześniej nie było pomocy. Jest duży problem. Wielu rolników, którzy z wielu względów musieli wygasić produkcję rolniczą, było przekonywanych przez doradców, przez przedstawicieli ministerstwa rolnictwa, że przecież ze względu na położenie, akurat mówię o województwie podlaskim, gdzie powstało wiele takich gospodarstw agroturystycznych. Dolina Biebrzy, okolice Puszczy Białowieskiej - tam te gospodarstwa działają. Dzisiaj stoją puste, dzisiaj nie ma pomocy dla nich, a rolnicy, kiedy pytają ministerstwo rolnictwa, co dalej, są odsyłani do ministerstwa rozwoju, a z ministerstwa rozwoju oczywiście do ministerstwa rolnictwa. I tak piłeczka jest cały czas odbijana. Dużo się mówi chociażby o Podhalu, mało się mówi o województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, a takich kwater w ostatnim czasie powstało tam dużo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Żyjemy w trudnym czasie pandemii. Pan prezydent ją podpisał. To świadczy o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości reaguje na potrzeby przedsiębiorców, społeczne. Ale chcę państwu przypomnieć historycznie, że to dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości zostały uruchomione takie programy pomocowe dla naszych rodzin jak 500+, 300+, trzynasta emerytura. Mamy w tej chwili pandemię. Mamy środki, dalej utrzymujemy te programy pomocowe dla polskich rodzin, bo rodzina jest podstawą w polskim społeczeństwie. Szanowni Państwo! Na te wszystkie potrzeby, które zgłaszają przedsiębiorcy, rząd reaguje, można powiedzieć, z dnia na dzień. Tylko w momencie, kiedy państwo nie mówią z tej mównicy, tylko gdzieś przy mównicy, a złapie to mikrofon, mówicie, że jednak te tarcze są dobre dla społeczeństwa, dla przedsiębiorców. Myślę, że polski rząd na czele z panem premierem nie zostawi potrzebujących przedsiębiorców i będzie ich wspierał w miarą możliwości. Czy w związku z drugą falą pandemii grożą nam wzrost bezrobocia i masowe zwolnienia? Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Decyzja rządu: zamykamy restauracje, puby, hotele, baseny i centra fitness. Poszkodowane firmy otrzymują: 100% czynszu za 3 miesiące, 100% wynagrodzeń i opłat. Dla przedsiębiorców, którzy nas słuchają, mam niestety złą wiadomość. Ta pomoc dla firm, o której powiedziałam, to nie jest decyzja polskiego rządu. Tak gospodarce pomagają Czesi. Brawo. Szybko, prosto i sprawiedliwie. Myślicie, że oni mają te swoje ciepłe posadki w spółkach Skarbu Państwa, jak wasze rodziny? Restauracja to nie tylko właściciel. To są kelnerzy, kucharze, osoby sprzątające. To są ci, którzy dostarczają im mięso, pieczywo i warzywa. To są te pralnie, które piorą im obrusy. Tak naprawdę to, co PiS robi dla polskiej gospodarki, przypomina reperowanie telewizora marki Rubin w PRL-u. Trzeba było raz go puknąć z góry, raz z boku i zaczynał działać, ale na krótko.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jarosław Rzepa, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Uchwalając tarczę 6.0, po raz kolejny podzieliliście państwo społeczeństwo i gospodarkę.

W Warszawie zarejestrowanych jest 12 tys. legalnych taksówek.

Dziś w tej sytuacji masowo rezygnują z prowadzonej działalności, choć aby uczciwie prowadzić swój biznes, musieli zdobywać licencje, zdać egzamin z topografii. A państwo polskie dzisiaj, szanowni państwo, co robi? Pieniądze idą do Irlandii, do Holandii, a w polskim budżecie nie zostają podatki. Panie ministrze, pan o tym wie, a państwo przedłużacie wejście lex Uber. Taksówkarze oczekują, że od 1 stycznia lex Uber wejdzie w życie, a nie po raz kolejny państwo to przesuniecie. Szanowni Państwo! Nie można dzielić w ten sposób PKD. Strata. Strata jest tym elementem, który powinien wyznaczać to, która z tych branż powinna zostać objęta wsparciem.

Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Pandemia zaskoczyła cały świat, nie tylko Polskę. Wiele gospodarek bardziej rozwiniętych, bardziej zasobnych niestety poradziło sobie znacznie gorzej niż nasz rodzinny kraj. Dzięki działaniom Prawa i Sprawiedliwości udało się bardzo szybko wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców. Państwo tego nie widzicie, ale jednak trzeba świat ocenić takim, jakim jest. Ponad 165 mld zł trafiło do polskiej gospodarki po to, żeby uratować ponad 6 mln miejsc pracy. To jest wartość, którą powinniśmy wszyscy wspólnie cenić.

Szanowni państwo, są pewne ograniczenia, które nie pozwalają wspierać wszystkich w taki sposób, o którym państwo mówicie. Ja jeszcze chciałabym podkreślić jedno, że dzięki takim intensywnym działaniom obecnego rządu wskaźniki dotyczące naszej gospodarki są jedne z lepszych w Europie, a nawet świecie.

A więc myślę, że te działania rządu, które zostały podjęte, przynoszą [[Dzwonek]] konkretne skutki. Ale ja mam pytanie do pana ministra: Jakie są podstawowe ograniczenia pomocy sektorowej dla branż dotkniętych kryzysem? Czy pomoc nie zaciemni jednak relacji rynkowych? Dziękuję serdecznie. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Czy tą dyskusją udowadniacie jednoznacznie, że jesteście kompletnie oderwani od rzeczywistości? Pani poseł powiedziała, że przecież branża turystyczna dostała bon turystyczny, tylko zapomniała dodać, że hotele są zamknięte. Bonu będzie można użyć może latem, a do tego czasu masa właścicieli w tej branży po prostu zamknie swoje interesy. To jest właśnie ten chaos w gospodarce, którego nie potraficie albo nie chcecie zrozumieć. Pan Janusz, właściciel kilku punktów gastronomicznych, był u mnie, by walczyć o swoje prawa przedsiębiorcy, bo w gastronomii robicie taki sam chaos. Chcecie zmuszać właścicieli punktów gastronomicznych, które dzisiaj nie działają, by do końca roku wymienili kasy fiskalne na kasy fiskalne on-line. Ale po co mają ponosić jakieś koszty, skoro ich punkty dzisiaj generują jakieś minimalne przychody, z których wielkiego urobku dla państwa i tak nie ma, bo dla przedsiębiorców ledwo co starcza?

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Andrzej Grzyb na łączeniu. Na łączeniu jest albo go nie ma. Czekając na pana posła, poproszę w takim razie panią poseł Marzenę Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam panią do mnie, poprowadzimy razem. Niech pani sobie wyobrazi, że pan poseł w sposób grzeczny, miły i sympatyczny przysłał mi SMS, że rezygnuje. Proszę pani, ja panią informuję z wielką przyjemnością, gdyż po prostu świetnie mi się z panią współpracuje. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proponowałabym jednak posłankom i posłom Prawa i Sprawiedliwości zejść na ziemię, porzucić te wielkie liczby i ministerialne stołki i posłuchać ludzi na dole, [[Oklaski]] tych ludzi, którzy prowadzą swoje firmy. Szanowni Państwo! Napisała do mnie w dniu 29 października, a więc jeszcze przed drugim czytaniem tzw. tarczy 6.0, pani Monika z Jędrzejowa.

Ale ona założyła firmę dopiero w tym roku i niestety z tej pomocy nie skorzysta. Powiedzcie, czy tak jest, czy tak nie jest. Nie skorzysta, dlatego że z tej pomocy mogą skorzystać tylko firmy, które powstały tak naprawdę do listopada, ale roku ubiegłego, bo do tego czasu można porównywać spadek przychodów. Pani Monika wczoraj napisała do mnie, że jest załamana, że to jest niesprawiedliwe, że liczy na to, że państwo zmądrzejecie, bo to jest nieludzkie tak różnicować ludzi. Przygotowaliśmy poprawkę do drugiego czytania, później głosowaliśmy nad uchwałą Senatu i na sali głosowaliśmy - trzy razy państwo odrzucaliście poprawkę mówiącą o tym, żeby wsparciem objąć również te firmy, które powstały w tym roku, [[Dzwonek]] albo chociaż te, które powstały po listopadzie roku ubiegłego. Byliście głusi. A więc tak wygląda wasza pomoc. Zejdźcie naprawdę na ziemię. Przeproszę pana posła Jana Łopatę, bo pani posłanka Anna Kwiecień prosiła o głos, dlatego że ma posiedzenie komisji, więc. Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Szanowni Państwo! Słyszymy od kilku dni, że kolejne gospodarki się zamykają, że tak naprawdę Europa zaciąga hamulec, ponieważ okazało się, że państwa zdecydowanie lepiej rozwinięte również mają ogromne problemy z koronawirusem i z epidemią. Jak wiemy, szanowni państwo, Niemcy już trzecią dekadę zajmują pierwsze miejsce w polskim eksporcie i imporcie towarów oraz usług. Zagraniczny popyt na niemieckie towary i usługi, w których zawarty jest polski komponent, odpowiedzialny był za blisko 29% polskiego eksportu do Niemiec. Polski eksport jest niezwykle silnie powiązany z niemiecką gospodarką. Panie ministrze, mam pytanie: Jak w tej chwili przełoży się na naszą gospodarkę, właśnie na eksport, ten ogłoszony niemiecki lockdown, pełny lockdown? Czy państwo planujecie przeanalizowanie, które firmy kooperują z niemieckimi przedsiębiorcami, i czy będzie można zastanowić się nad tym, czy nie wesprzeć tych firm, których działalność niestety jest silnie powiązana [[Dzwonek]] z niemiecką gospodarką?

Bardzo dziękuję, panie marszałku. Można. Te wszystkie wycieczki polityczne, połajanki personalne, myślę, ani teraz, ani nigdy nie przynoszą efektu. Polaków, którzy być może, a nawet na pewno teraz słuchają nas i oczekują konkretnej odpowiedzi. Słuchają zapewne, bo większość firm niestety jest pozamykana i mają więcej czasu na to, by śledzić, co się dzieje wokół nich. Niestety nie dzieje się dobrze. Mówicie tu państwo o kolejnych tarczach, o tarczy nr 6, i natychmiast pojawiają się następni, którzy zgłaszają kolejną branżę. Ja też w tej chwili zgłoszę branżę, o której zgłoszenie mnie proszono, a mianowicie branżę zajęć edukacyjnych dodatkowych, PKD 85.52.Z.

Nie jesteśmy w stanie. Cały katalog PKD należałoby wpisać, bo dzisiaj jest taka sytuacja. Tak się nie da zrobić. To musi być kryterium obiektywne, ale ogólne, typu chociażby, nie wiem, przychody rok do roku. Trzeba wziąć [[Dzwonek]] przykład z innych państw i taki system wprowadzić, abyśmy ciągle nie mówili, że kolejna branża jest wyeliminowana. Zapraszam pana posła Piotra Borysa z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Trzeba naprawdę wyjść z gabinetu ministerialnego, z tych nowych aut, pojechać na południe Polski, porozmawiać z właścicielami pensjonatów, hoteli, restauracji, z których 80% nie pracuje - nie pracuje, po prostu branże zostały de facto zamknięte. Każde solidarne państwo, które zamyka w czasie pandemii branże, daje ekwiwalent utraconych korzyści, a przynajmniej pokrywa koszty działalności. Właściciele pensjonatów, hoteli nie mają możliwości uzyskania pomocy. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, która dokładnie w oparciu o kryterium utraty przychodów daje zabezpieczenie wszystkim tym, którzy dzisiaj stoją na skraju bankructwa. Dlatego żądamy, aby nasz projekt ustawy ratujący branże turystyczną i okołoturystyczną, choć nie tylko, był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu w czwartek i w piątek.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Anna Milczanowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Choćbyście państwo nie wiem jak zaklinali tę rzeczywistość i mówili do nas, żebyśmy zeszli na ziemię, my stąpamy bardzo mocno po ziemi w poczuciu odpowiedzialności, w poczuciu odpowiedzialności za państwo.

Panie Ministrze! Jak przedstawia się aktualna sytuacja w handlu zagranicznym? Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! A przede wszystkim: Panie Ministrze i Panie Posłanki z PiS-u! To, co wy mówicie, naprawdę jest z kosmosu. Mówicie, jakbyście żyli na innej planecie. Pandemia naprawdę pustoszy polską gospodarkę i naprawdę setki tysięcy przedsiębiorców mają ogromne problemy.

Naprawdę znam to środowisko bardzo dobrze. Chciałem zadać konkretne pytania, ponieważ ta wasza pomoc jest wprowadzana późno, jest chaotyczna, jest nieprzewidywalna i nierównomierna. Wszyscy wam to mówią.

Jest połowa grudnia, branże są pozamykane, rozporządzenia brak. Czemu dalej tak bardzo mało wiadomo o PFR 2.0? Czemu nie działają rozwiązania kredytowe?

Ostatnie pytanie: Czemu nie pozwalacie rozciągnąć ferii? Wszyscy wiemy, że część ludzi omija zakazy, przyjeżdża w jednym tygodniu, a tak mogliby przyjeżdżać przez 10 tygodni i pomóc branży działać w odpowiednim reżimie sanitarnym. Zejdźcie na ziemię i zacznijcie pomagać polskim firmom. Pani poseł Teresa Wargocka, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jest pani poseł? Jest. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Zatrzymano wzrost zachorowań. To góralka z Podhala mówi: tych dutków to my żeśmy trochę zebrali. Proszę mi dać dokończyć. Szanowni Państwo! Dzisiaj musimy się zastanawiać, co dalej.

Dzisiaj mamy możliwość wyjścia z tego kryzysu za pomocą szczepień. Mam pytania do pana ministra. Co z Krajowym Planem Odbudowy? Na jakie wsparcie może liczyć polska gospodarka w związku z nową perspektywą unijną, z nowymi pieniędzmi, które są potrzebne i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie? Dziękuję bardzo. Pani posłanka Monika Rosa, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tę pomoc udzieloną polskim przedsiębiorcom można opisać słowami: za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. Ponieważ to,

Czy szykują się kolejne zamknięcia, lockdowny?

Czy mają państwo przewidywania co do wzrostu skali upadłości polskich firm, czy nastąpi on już teraz, może na wiosnę, czy państwo czegoś takiego nie przewidują i wsparcie państwa nie będzie potrzebne? A jeśli będzie potrzebne, to jak to wsparcie będzie wyglądało, jakie to będą kwoty, jakie to będą narzędzia, jakie instrumenty?

Dziękuję serdecznie. Udało się uzyskać połączenie z panem posłem Grzegorzem Matusiakiem, o które zabiegaliśmy. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zanim przejdę do pytania, chciałbym przypomnieć posłom Platformy Obywatelskiej ich troskę o tzw. przedsiębiorstwa państwowe.

Szczególnie chodziło o ratowanie branży górniczej.

wręcz przeciwnie, starano się tę branżę pogrzebać. Dzisiaj, przypomnę, jeżeli chodzi o wsparcie branży turystycznej, że pomoc, jaką uzyskała branża turystyczna, to przede wszystkim pomoc z PFR - 5 mld, a 4 mld to: bon turystyczny, postojowe, zwolnienia z ZUS.

Jest przygotowywany następny pakiet wsparcia branży turystycznej. Która branża najbardziej ucierpiała i jak wsparto branżę turystyczną? Dziękuję bardzo. Czy pani poseł Barbara Dziuk jest na sali? A zwracam zawsze uwagę.

Proszę pani, po prostu przepraszam panią. Wielichowska, oczywiście. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Gospodarka gaśnie na naszych oczach, ofiarami koronawirusa są nie tylko osoby, które zaraziły się wirusem, ale też przedsiębiorcy. Wystarczy wysiąść z limuzyny albo przestać odwiedzać pusty - pełen propagandy zamiast pacjentów - Szpital Narodowy i porozmawiać z przedsiębiorcami, tak jak ja rozmawiam z panem Arkiem ze Stronia Śląskiego, z panią Anną z Kłodzka, z panem Wojtkiem z Nowej Rudy, z panem Adamem z Dzierżoniowa czy z panią Kasią z Ząbkowic.

Dziś nie wiedzą, jak ustrzec się przed upadłością. Czy rząd ma jakąś strategię, może jakiś plan chociaż albo jakiś mały planik?

Dziękuję serdecznie pani poseł Monice Wielichowskiej. I zapraszam pana posła Waldemara Andzela, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość rozmawia z wyborcami, rozmawia z przedsiębiorcami. Ja rozmawiam i z panem Arkiem, i z panem Mateuszem, przedsiębiorcą. Rozmawiamy. Nie przeszkadzajcie tu w tej sali. Prawo i Sprawiedliwość twardo chodzi po ziemi. Polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze na tle gospodarki całej Europy.

Mam pytanie do pana ministra: Jak wygląda produkcja przemysłowa, tak istotna dla generowania polskiego PKB? Na jakich podstawach oparte jest przekonanie, że w 2021 r. czeka nas wzrost gospodarczy? Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, panie pośle. Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za prawidłowe akcentowanie: Gramatyka, jestem pełen szacunku i pełen dumy z pana marszałka. Pani posłanka Leszczyna powiedziała, że jesteście bezradni wobec gospodarki w kryzysie. Ja powiem więcej: jesteście bezradni wobec gospodarki w ogóle. Nie wiem, czy pamiętacie państwo ten slajd: to są wasze cele na rok 2020. Gdybyście dobrze je realizowali, może dzisiaj nie byłoby tej dyskusji, może polska gospodarka byłaby w dużo lepszym stanie. Tylko trzy przykłady, bo na tyle pewnie starczy czasu. Dużych i średnich firm miało być ponad 22 tys., a z ostatnich danych GUS wynika, że jest ich 18 tys., czyli o 300 mniej niż wtedy, kiedy zaczynali państwo rządzić.

Jakoś trudno nazwać to sukcesem. Kapitał dla rozwoju, czyli wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do PKB, miał mieć poziom 25%, wyszło jak zwykle: na koniec roku 2019 ten wskaźnik wynosił 18 punktów procentowych. Proszę zwrócić uwagę, że to są dane sprzed pandemii. Z litości podaję dane sprzed pandemii. Przychodzi mi do głowy cytat z Budki, ale nie z Borysa Budki, tylko z Budki Suflera: To nie tak miało być, zupełnie nie tak. Tak rządzicie. Coraz rzadziej się śnią tęczowe mosty. Dziękuję. Myślę, że pan poseł Budka też doczeka się takiej chwili, że będą go cytowali z mównicy sejmowej. Tak że życzymy tego panu posłowi Budce. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wiele tutaj słów padło: nie chodzimy po ziemi, nie chodzimy wśród ludzi. Mieszkamy tak jak państwo gdzieś tam w swoich miejscach i do nas też się zwracają przedsiębiorcy ze swoimi kłopotami i zgłaszają problemy. Tak że to nie jest tak, że nie widzimy problemów, z którymi się zmagają przedsiębiorcy, szczególnie aktualnie branża turystyczna.

Ale pandemia się kiedyś skończy i mam w związku z tym do pana ministra pytanie: Czy ministerstwo przewiduje zmiany legislacyjne mające na celu ułatwienie działalności gospodarczej już w warunkach, kiedy COVID się skończy? Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że na początek wszyscy musimy zadać sobie pytanie, czy tę porażającą nieudolność rządu w sprawie pandemii, ten chaos, tę niepewność, którą rząd wprowadza, można usprawiedliwiać rządami sprzed 8, 10, 15 czy 30 lat, czy raczej posłowie PiS powinni tutaj przyjść i przeprosić Polaków za swój rząd, za to, że wprowadza taki chaos, taką niepewność i niszczy państwo. Niszczy gospodarkę, niszczy ludzi, którzy ciężko pracowali przez całe życie, żeby zbudować swój biznes. Za te nieodpowiedzialne działania, które firmujecie swoimi głosowaniami. Tymczasem są takie branże jak branża współpracy transgranicznej polsko-czeskiej, polsko-słowackiej, które nie mają PKD. Ale wy tego nie rozumiecie. Dzisiaj ta branża umiera, ale nie potraficie im pomóc. A to, co rząd PiS robi w branży turystycznej, zwłaszcza tym przedsiębiorcom, którzy działają w regionach turystycznych: w Beskidach, Wiśle, Szczyrku, Ustroniu, Brennej, Bystrej, to po prostu polityczny kryminał. Najpierw rząd PiS wprowadza lockdown miejscowości turystycznych w czasie ferii, a teraz zmienia bon turystyczny w taki sposób, że rozszerza go na imprezy jednodniowe.

I pytanie, czy rząd pójdzie po rozum do głowy i wreszcie stworzy albo przyjmie przygotowany przez Koalicję Obywatelską mechanizm wsparcia przedsiębiorców w miejscowościach turystycznych, bo oni dzisiaj tego potrzebują. Pani poseł Agnieszka Górska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, sytuacja firm, przedsiębiorstw, dzięki którym wytwarzany jest tak ważny dla gospodarki produkt krajowy brutto, jest bardzo trudna. Pandemia wymusza kolejne ograniczenia, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić odpowiednią pomoc dla polskich firm i przedsiębiorstw. Wszyscy doceniamy wielki wkład pracy całego rządu już od kilku miesięcy, od pierwszego dnia epidemii w ograniczanie negatywnych skutków COVID-19. Wszystkie rozwiązania do tej pory wprowadzone przez rząd względem gospodarki i przedsiębiorców są nieocenione w tym trudnym czasie. Niezależnie od tego, co mówi opozycja, to fakt.

To chociażby tzw. estoński CIT, specjalny fundusz inwestycyjny czy zmiany zwiększające limit przychodów dla zastosowania niższej stawki VAT-u. Przedsiębiorcy liczą po wprowadzeniu tych rozwiązań na uzyskanie płynności, tak potrzebnego czasu i stabilności dla swoich firm. Jak te zmiany wpłyną na naszą gospodarkę? I kolejne moje pytanie: Jakie jeszcze działania mające na celu przyspieszenie odbudowy gospodarki po pandemii wprowadza ministerstwo? Nadmienię również, że dużą szansą na rozwój są także środki z europejskiego funduszu gwarancyjnego, najnowszej wspólnej tarczy państw członkowskich (Dzwonek) przeciwko pandemii. Do przedsiębiorców ma trafić co najmniej 20 mld zł w ciągu najbliższych lat.

Głównym celem funduszu jest zapewnienie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez zwiększenie im dostępu do finansowania. Czy instytucje te już przygotowały odpowiednią ofertę? W tych działaniach uczestniczy również Bank Gospodarstwa Krajowego. Media już dziś w tym kontekście wskazują, że analizuje on aktualne oczekiwania sektora MŚP odnośnie do wsparcia leasingu, gdyż do tej pory nie było dedykowanego produktu gwarancyjnego dla tej formy finansowania. Po dzisiejszej dyskusji strach pomyśleć, co by się działo, gdyby Platforma z PSL-em dalej rządzili w kraju. Krzyk, awantury, granie na emocjach, nienawiść, dzielenie Polaków - to główne wasze rozrywki. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Katarzyna Lubnauer, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie i panowie posłowie! Panie Marszałku! Ja mam wrażenie, że tylko z okien limuzyn. Mówią też, że rozmawiają z przedsiębiorcami. Tak, przy pomocy policji. Policja rzeczywiście dość licznie przybywa na protesty przedsiębiorców, którzy - jak widać - protestują, bo są tak zachwyceni tym, jak rząd im pomaga. Ostatnio jechałam taksówką i taksówkarz powiedział, że jest to jego pierwszy kurs po czterech godzinach stania i czekania na to, że pojawi się jakikolwiek klient. Tak się składa, że branża taksówkarska nie została zamknięta. Dlaczego narzekają? No może dlatego, że jeżeli zamknięte są restauracje, do których nie ma po co wozić klientów, jeżeli zamknięte są teatry, kina, jeżeli ludzie nie urządzają hucznych imprez, ponieważ po prostu jest koronawirus, jeżeli nie ma ślubów, jeżeli nie ma wesel, jeżeli nie ma tego wszystkiego, co powoduje, że korzystamy z taksówki, to taksówkarze nie mają kursów. Najzwyczajniej w świecie oni muszą zapłacić dzierżawę za samochód, muszą zapłacić podatki, a nie otrzymują żadnych pieniędzy od klientów. On spytał wprost: Czy jedyną pomocą, którą otrzymają od państwa, ma być zwolnienie z ZUS-u na jeden miesiąc, na listopad? Jak on ma przeżyć? Jak on ma zapłacić ten ZUS w następnych miesiącach? Jak on ma zapłacić opłaty za samochód, albo ratę kredytu albo dzierżawy? Jak ma przeżyć z rodziną?

Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Adama Szłapkę, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z powodu pandemii rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje różne działania dotyczące gospodarki.

Dlatego pytam pana ministra bardzo konkretnie: Na podstawie jakich analiz, jakich badań, jakich rozmów, jakich konsultacji została zawieszona branża fitness w ostatnich tygodniach? Proszę o odpowiedź na piśmie. Jakie konkretne ekspertyzy, badania i analizy zostały przez rząd zamówione i przeprowadzone, które posłużyły jako podstawa do podjęcia tej decyzji? Czy wy wiecie, że w branży fitness są bardzo duże sieci, które zatrudniają wiele osób na umowę o pracę, i te firmy zostały pozbawione jakichkolwiek możliwości wpływów? Zgłaszają się do biur poselskich właściciele takich siłowni. Czy wy wiecie, że w ramach branży fitness działają trenerzy pracujący na umowę zlecenie w klubach i siłowniach? Czy wy wiecie, że są ludzie, trenerzy, którzy prowadzą działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i którzy też zostali pozbawieni jakiejkolwiek możliwości zarobkowania przez ten czas? Z dnia na dzień. Dlatego pytam konkretnie i proszę o przesłanie na piśmie tych analiz, tych ekspertyz i tych badań, na podstawie których wy podejmowaliście w tej sprawie decyzję. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Teresa Pamuła, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam panią poseł. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Branże nie zostały zamknięte, tak jak państwo tutaj mówicie. Gospodarka pracuje, dlatego jesteśmy tutaj. Oczywiście taksówkarze są w bardzo trudnej sytuacji, ale proszę państwa, te 150 mld, prawie 160 mld, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wpompował w gospodarkę, uratowało gospodarkę i nas wszystkich, Polaków. I nie chcemy, żeby państwo opowiadali tutaj nieprawdę, wmawiali Polakom nieprawdę.

Udało się dofinansować branżę sanatoryjną.

Nikogo nie zwolnili.

Wysoka Izbo! Jest takie powiedzenie: w zdrowym ciele zdrowy duch. Mówię to również jako syn polskiego olimpijczyka.

90% pracowników branży fitness zatrudnionych jest na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, najczęściej jest to umowa zlecenia. Przed wybuchem epidemii w Polsce działało prawie 3 tys. klubów fitness, do których uczęszczało nieco ponad 3 mln osób.

I to jest również przykład działań irracjonalnych.

To pokazuje, jak nieracjonalne były decyzje. Apeluję wprost: Panie ministrze, branża fitness czeka na czytelne regulacje, na realną pomoc, która musi zostać zaoferowana, i konkretną perspektywę, dotyczącą otwierania tych obiektów.

Dziękuję serdecznie. A mówił do państwa syn dwukrotnego medalisty olimpijskiego. Będziemy się łączyli z panią poseł. Witam serdecznie. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, aby w jak największym stopniu złagodzić jej negatywne skutki, zresztą dzisiaj moi przedmówcy bardzo celnie wskazywali, jak wielka to jest pomoc, jak bardzo jest w stanie wesprzeć wiele gałęzi i jak wielu przedsiębiorcom się tu pomaga. W perspektywie długotrwałego oddziaływania pandemii na gospodarkę. Nawet po wprowadzeniu w życie programu szczepień piętno pandemii będzie wciąż oddziaływać, np. na branżę gastronomiczną, taksówkarską i kilka innych.

Stąd pytanie, panie ministrze: Czy można przewidywać, jakie branże po epidemii będą musiały w największym stopniu przedefiniować swoje strategie biznesowe? Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości tak pięknie opiekuje się przedsiębiorcami, więc również ta strategia, wskazanie dziś, [[Dzwonek]] gdzie w przyszłości przedsiębiorcy mogą widzieć dla siebie możliwość realizacji swoich pomysłów, biznesowych koncepcji, na pewno bardzo im pomoże. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Panie Ministrze!

Pani poseł mówiła o empatii wobec ludzi.

Staramy się pomagać i dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości miał pieczę nad finansami państwa przez poprzednie 4 lata, potrafiliśmy doprowadzić do sytuacji, że budżet mógłby być w tym roku bez deficytu.

Po pierwsze, czy jest szansa, że dzieci wrócą do szkół? Ona skorzystała z tarczy, otrzymała pożyczkę, miała 15 pracowników, jednak w tym momencie nie ma prawie żadnych dochodów, więc większość zwolniła.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Agnieszka Soin, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszyscy doskonale wiemy, że tarcze antykryzysowe skutecznie ochroniły przed skutkami kryzysu i utrzymały wskaźnik bezrobocia na stałym poziomie. Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia na koniec października br. wyniosła 6,1%, co oznacza, że przez kilka miesięcy bezrobocie było na stałym poziomie. Pandemia COVID-19 jest poważnym wstrząsem dla gospodarki oraz może przyczynić się do znacznego zmniejszenia liczby miejsc pracy i wzrostu bezrobocia. Proszę pana ministra o informację, jakie są perspektywy rynku pracy na koniec 2020 r. oraz czy stabilizacja pracy utrzyma się również w przyszłym roku. Czy w najbliższym okresie powinniśmy spodziewać się wzrostu bezrobocia? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Andrzej Grzyb, klub parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że nikt nie kwestionuje faktu, że pieniądze publiczne z budżetu państwa zasiliły przemysł i usługi w okresie pandemicznym. Jest tylko pytanie, czy zasiliły w sposób równomierny. Czy wszystkie działy gospodarki, czy wszystkie typy działalności gospodarczej miały szansę na uzyskanie tej pomocy? Konserwatorzy urządzeń do rozlewania napojów, którzy są zarejestrowani w PKD jako inna działalność - gdyby byli zarejestrowani jako prowadzący działalność w branży metalowej, to mieliby szansę. Natomiast w innej działalności - nie mają. To są więc te kwestie, które wracają do nas jako do posłów do parlamentu. Ci przedsiębiorcy próbują znaleźć u nas zasadne skądinąd wsparcie, żeby nie przynależność do kryterium działalności gospodarczej PKD miała pomóc czy być podstawą do pomocy, ale przede wszystkim, żeby utrata przychodów w tych firmach była tym warunkiem. Jest to trudniejsze, zdajemy sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony wiemy też, że jeżeli chodzi o Polski Fundusz Rozwoju, planowana transza dla dużych firm to było 25 mld zł. Wykorzystanych będzie prawdopodobnie 10, ponieważ wiele firm się wykruszyło z własnej inicjatywy, ale z powodów obiektywnych, stwierdzonych przez organa publiczne. Stąd też istnieje pewna rezerwa w publicznych środkach, która mogłaby zasilić [[Dzwonek]] w szczególności małe i średnie firmy, w tym również te firmy, o których tutaj często mówiono: gastronomiczne, turystyczne, prowadzące działalność dietetyczną. Proszę państwa, do zakończenia dyskusji pozostało nam 10 minut, bo jak wiecie, 90 minut trwa ten punkt. Jest dwóch mówców - po 5 minut.

Panie Marszałku! To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to fakt, że dzisiaj nie widać, aby rząd - również pan minister - miał spójny pomysł, jak wygląda sprawa dzisiaj, jak ma wyglądać na najbliższe miesiące dla branży turystycznej i wszystkich branż, które z tą branżą są powiązane. To są dostawcy wszelkiego rodzaju dóbr. Nie widzimy również i nie zobaczyliśmy przez te wiele miesięcy wypowiedzi pana ministra, czy są jakieś realne analizy. Czy to nie jest nerwowe łapanie się za ścianę i decydowanie pod wpływem tego, że poprzedniego dnia w takim czy innym medium taki czy inny materiał prasowy, medialny się pojawił i: dawaj, zamykamy - tak jak to było przy okazji cmentarzy? Tak naprawdę państwo nie jesteście przyjaciółmi firm rodzinnych, bo wszystkie wasze rozwiązania nie uwzględniają firm rodzinnych w postaci spółek cywilnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, ale również spółek prawa handlowego, przypadków, kiedy mamy do czynienia z firmami, w których jest żona, mąż, ewentualnie dzieci, które pomagają w tym biznesie, właśnie w różnego rodzaju hotelach, pensjonatach, restauracjach, barach, bo tak naprawdę dajecie pieniądze na ochronę miejsc pracy w większych zakładach.

Nie pomagacie rodzinnym firmom, a z drugiej strony wprowadzacie takie zasady, które pozwalają kantorom wymiany walut czy kancelariom adwokackim występować o pieniądze na tzw. utrzymanie miejsc pracy, gdy właśnie rodziny popadają w potężne tarapaty finansowe nie tylko z tego powodu, że nie mają na bieżące rzeczy, że nie mają bieżącego wpływu ale to jest kwestia również opłacania leasingów, rachunków za dostarczone media, kredytów, które często są pobrane na inwestycje w ostatnich latach. To są realne pożyczki, to jest zawieszenie płatności ZUS dla wszystkich, którzy prowadzą dzisiaj działalność gospodarczą, zawieszenie rat kredytów, leasingów, pożyczek do czasu trwania ograniczeń, które zostały podjęte przez rząd. Dziś zakłady dystrybucji prądu zaczynają odłączać prąd różnego rodzaju pensjonatom. Chcecie przykłady tego, jak zadziałała pierwsza tarcza. Co robi dzisiaj? Musiał wypowiedzieć wszystkim pracownikom umowy o pracę, gdyż nie ma perspektywy na sezon, nie ma perspektywy na pomoc. Co to oznacza? Że zostały wydane pieniądze, które tak naprawdę zostały spalone w kominku. Może być i drugie tyle, tylko to jest tak jak zabawa dzieciaka, który do palącego się ogniska dolewa benzyny i cieszy się, że płomień na chwilę jest wielki. Jak nie dołożymy dzisiaj drewna, to tak naprawdę to ognisko bardzo szybko zgaśnie. Prosimy pana ministra o to, żeby pan na wszystkie nasze pytania odpowiedział na piśmie, bo na niewiele z nich dostaliśmy jakąkolwiek odpowiedź. Przecież wy nie macie własnych pieniędzy. Jeśli ci podatnicy zostaną teraz, dzisiaj zarżnięci, to nie będzie z czego oddawać. Nie będzie za co tego spłacić, bo przecież to nie są pieniądze, które wyjęliście panu Morawieckiemu z konta ani panu Kaczyńskiemu z szuflady, tylko to są pieniądze Polaków. Zadłużacie się, ale te długi ktoś będzie musiał spłacić. Nie wy, nie pan Kaczyński, tylko wszyscy Polacy. PFR dzisiaj tak naprawdę jest instrumentem, który za chwilę będzie oligarchizował polską gospodarkę. Upadające hotele będzie można za złotówkę odkupić czy przez PFR, czy przez Polski Holding Hotelowy - państwową firmę.

Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, panie ministrze. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pan minister Robert Tomanek. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję państwu za zgłoszone pytania, za uwagi. Wszystkie były notowane przez moich współpracowników i przeze mnie. Dyskusja była bardzo inspirująca i pouczająca dla mnie. Oczywiście na wszystkie państwa pytania zostaną udzielone odpowiedzi. Będą one opatrzone wyjaśnieniami przygotowanymi w oparciu o wiedzę, którą dysponuje resort.

Skala pomocy tarczowej to jest 8% polskiego produktu krajowego brutto. To, co otrzymujemy jako wsparcie z Unii Europejskiej, to jest niecałe 5%, licząc PKB roczne w całej perspektywie finansowej. Czyli 8% to jest naprawdę dużo. Musimy mieć świadomość, że jest to duży wysiłek całego społeczeństwa i państwa. Możliwość rozciągania tej pomocy na większą skalę jest ograniczona.

To jest duże ryzyko. Sygnalizują to sami przedsiębiorcy, zwracają na to uwagę, krytykując również instrumenty, których użyliśmy.

Siłą polskiej gospodarki jest przede wszystkim eksport. Osobiście pokładam bardzo duże nadzieje w systemach samoregulacji gospodarki. Większe - może to zabrzmi paradoksalnie - niż w instrumentach wspierania takich czy innych branż. W jaki sposób to skierować? Pomoc horyzontalna jest niedoskonała. Pomoc branżowa jest niedoskonała. Rząd musi dokonywać trudnych wyborów. To jest obowiązek rządu. Musimy liczyć się z krytyką, ale jesteśmy w stałym dialogu nie tylko z parlamentem, lecz także z grupami przedsiębiorców. Przedstawiciele branż, o których państwo mówiliście, są stałym gościem w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Trudno. Stało się tak z różnych powodów, różne są argumenty. Nie chciałbym się wdawać w dyskusję, bo nie jestem epidemiologiem.

Przepraszam, że nie zaspokoiłem wszystkich potrzeb informacyjnych. Obiecuję również jak najrzadziej korzystać z limuzyn. Nie cierpię tego. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.

Już raz rękę złamałem.

Proszę państwa, wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przechodzimy do następnego. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o rządowych projektach ustaw: - o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., - o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości ministra sprawiedliwości Tajwanu. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 837 i 838.

Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 687 i 796) Proszę pana posła Piotra Saka o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawiam sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zawarty jest w druku nr 687, zaś sprawozdanie komisji inkorporowane jest w druku nr 796. Przypominam, że 27 listopada skierowano rzeczony projekt do komisji, zaś 2 grudnia komisja obradowała na posiedzeniu komisji. W trakcie posiedzenia odbyła się wstępna, aczkolwiek dość ożywiona i pogłębiona, dyskusja na temat nowych konstrukcji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej oraz nowej usługi sieciowej umożliwiającej elektroniczne uzyskiwanie danych z Krajowego Rejestru Karnego, tak naprawdę taki nowy kanał uzyskiwania informacji z tego rejestru. Proponowane zmiany ukierunkowane są na zautomatyzowanie i odhumanizowanie uzyskiwania zaświadczeń wydawanych przez organy administracji publicznej. Odejście od tradycyjnych i nieco już archaicznych form umożliwi szybszy i sprawniejszy dostęp do uzyskiwania informacji zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. Te nowe rozwiązania racjonalizatorskie mają skutkować według deklaracji strony rządowej bardziej sprawnym, operatywnym, szybszym, bardziej dynamicznym uzyskiwaniem informacji. Ten czas ma być skrócony do jednego dnia. W trakcie rozpoznawania projektu wprowadzona została jedna poprawka, mająca charakter legislacyjno-redakcyjny. Pozostałe nie zostały przyjęte. Dziękuję na tym etapie za spokojną, wyważoną i merytoryczną dyskusję. Liczę na kontynuację tej atmosfery w dalszym czasie prac legislacyjnych. Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę panią poseł Barbarę Bartuś, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę serdecznie. Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 796. Mimo że nazwa projektu ustawy mówi o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego, to główną przyczyną opracowania projektu i omawianych zmian było, wydaje się, ogromne zapotrzebowanie na informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Obecnie procedura udzielania informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego uregulowana jest w ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. Z roku na rok do Biura Informacyjnego KRK wpływa coraz więcej zapytań i rocznie już dawno liczba tych zapytań przekroczyła 1 mln. Tymczasem sposób udzielania informacji nie zmienił się w swoich założeniach od utworzenia Krajowego Rejestru Karnego w 2000 r., kiedy zapotrzebowanie na informacje z KRK było kilkakrotnie mniejsze. Dotychczas podejmowane działania w celu usprawnienia pracy biura koncentrowały się na optymalizacji dostępnych zasobów ludzkich i technicznych, jednakże możliwości dalszego funkcjonowania biura w obecnym kształcie i przy wykorzystaniu posiadanych zasobów przestają być wystarczające. Dlatego z propozycją zmian rząd po raz pierwszy wystąpił już w ubiegłej kadencji. Powróciliśmy teraz. Nowe rozwiązanie dotyczące udzielania informacji ma zapewnić większy stopień automatyzacji procesu przetwarzania danych przez m.in. dostarczanie określonym podmiotom usługi sieciowej. Podmioty te w celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego nie będą musiały składać zapytania, ale za pomocą aplikacji, którymi już dysponują, będą mogły wysyłać do systemu Krajowego Rejestru Karnego żądanie udzielenia informacji. Na podstawie żądania nastąpi automatyczne przeszukanie i weryfikacja danych. Odpowiedź na takie żądanie zostanie udzielona synchronicznie, tzn. bez udziału pracownika, bez udziału osoby. Zaproponowane we wniosku rozwiązania mają szczególne znaczenie przede wszystkim dla sądów, prokuratury, Policji, służb specjalnych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość deklaruję poparcie dla tego rządowego projektu. Jednak aby usprawnić jeszcze, dopracować ten projekt składam na pana ręce poprawki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Tomasza Zimocha, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pod koniec listopada, kiedy rozpoczynaliśmy prace nad projektem tej ustawy, powiedziałem, że proponowane zmiany wydają się wskazane, choć zaufanie do wszelkich rządowych projektów i ich autorów zmalało niemal do zera. Miałem jednak nadzieję, że uchwalimy ustawę w trybie mini-max - minimum zbędnych słów, maksimum dobrego prawa. Obawy okazały się słuszne. Krótki projekt, tylko cztery artykuły, można było go dokładnie przygotować, a okazuje się, że to zadanie trudne jak zdobycie K2 zimą. Zgodnie z sugestiami Biura Legislacyjnego w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej zgłaszam poprawkę dotyczącą uszczegółowienia delegacji ustawowej dla ministra sprawiedliwości do wydania przepisów wykonawczych tak, aby rozporządzenie wydane na jej podstawie uwzględniało także specyfikę udzielania informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W czasie posiedzenia komisji Zjednoczona Prawica zgłosiła siedem poprawek. A chciałoby się, by szczególnie rządowe projekty były wyjątkowo dopieszczone. Ale i zgłaszane poprawki nie mogą być wadliwe, i to z dwóch powodów. Z powodu przekroczenia zakresu przedłożenia - poprawki nie dotyczyły przedmiotu nowelizacji przedstawianego w pierwszym czytaniu, to obejście trzech czytań, znaczące naruszenie procedury, chyba że państwo robią to celowo, by Trybunał Konstytucyjny przestał być bezrobotny. Poprawki nowelizujące kodeksy muszą mieć też szczególny tryb procedowania i pierwsze czytanie zmian kodeksu powinno się odbyć na posiedzeniu plenarnym, a tak nie było i nie jest. Rekomenduję zatem głosowanie przeciwko tym poprawkom, jeżeli one tak brzmią, a w przypadku ich przyjęcia - głosowanie przeciwko przyjęciu całej ustawy. Sejm nie może przyjmować ustaw z naruszeniem prawa. Sejmu na to nie stać. Chodzenie na skróty bardzo często powoduje zupełne zagubienie. Rządzący chodzą niestety w Sejmie na skróty. Apeluję o procedowanie w trybie mini-max - minimum błędów, maksimum dobrego prawa. Jeszcze prośba do przewodniczącego, do pana, panie pośle, by pracował pan w czasie posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej w trybie mini-max - minimum pogardy, minimum nieżyczliwości, a maksimum uprzejmości. Uprzejmości, czyli lepiej nie odmawiać posłom możliwości wykonywania normalnej pracy, choćby wtedy kiedy zapowiada pan, że poprawki przedstawi pan w stosownym czasie, bez możliwości zapoznania się z nimi przez członków komisji. Przewodniczy pan Komisji Nadzwyczajnej, ale ja proszę tylko o zwyczajne, normalne pana zachowanie. Nie namawiam do wejście zimą na K2, bo to dla pana nieosiągalne, ale osiągalne, panie pośle, są dla pana podstawowe zasady savoir vivre. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Roberta Kwiatkowskiego, klub parlamentarny Lewica. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powiało grozą po wystąpieniu posła Zimocha, zupełnie tak jak na K2 zimą, choć nie było mnie tam, ale spodziewałem się, mówiąc szczerze, nieco bardziej ciepłego przyjęcia tego rządowego przedłożenia, ponieważ jednak w odróżnieniu od poprzednika klub parlamentarny Lewicy ma stosunkowo pozytywne podejście do tego rządowego przedłożenia. Choć rzecz jasna diabeł tkwi w szczegółach i ta moja wypowiedź nie będzie wolna od akcentów krytycznych. Ale na początku przypomnijmy, że, tak jak mówiła o tym pani poseł Bartuś, właściwie to przedłożenie rządowe rozwiązuje ok. 80% problemów, jeśli za problem uznajemy konieczność obsłużenia i odpowiedzenia na idące w miliony pytania z różnych stron do Krajowego Rejestru Karnego, bo taka jest istota tego rządowego przedłożenia i tej nowelizacji.

No i świetnie, można powiedzieć. Może trochę szkoda tych pięćdziesięciu paru pracowników, którzy tym się do tej pory zajmują, ale wierzę, że administracja rządowa znajdzie dla tych ludzi inne miejsce i inną pracę, tym bardziej że wymiar sprawiedliwości po sławetnych reformach autorstwa Ziobry raczej cierpi na rosnącą przewlekłość postępowań, niż szczyci się tym, że jest tego coraz mniej i ludzie krócej czekają w sądach na rozpatrzenie ich spraw. Otóż najciekawsze, moim zdaniem, jest to, że resort sprawiedliwości i, zdaje się, cały rząd dalej uprawiają taką silosową filozofię działania.

Dlaczego resort sprawiedliwości nie doprowadził do sytuacji, w której ustawa o doręczeniach elektronicznych, bardzo potrzebna, rozwleczona w czasie... 9 lat, panie marszałku, 9 lat będziemy czekali na ostateczne sfinalizowanie kwestii doręczeń elektronicznych. Dlaczego resort sprawiedliwości nie zajął się tymi problemami, nie doprowadził do tego, że nie tylko Agencja Wywiadu i Służba Ochrony Państwa, ale też zwykły przedsiębiorca, który bierze udział w jakimś przetargu i potrzebuje zaświadczenia o niekaralności, nie może szybko, bezpiecznie i bezproblemowo uzyskać takiego zaświadczenia? Mogę formułować kolejne pytania, ale powiem na koniec, że zdaje się, że nasza dyskusja - odnoszę się do tego, o czym mówił szanowny przedmówca, pan poseł Zimoch - jest w wariancie mini-mini. To znaczy posłowie mogą sobie porozmawiać, a z rządu ani z Ministerstwa Sprawiedliwość, ani z resortu cyfryzacji czy, przepraszam, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo nowym ministrem cyfryzacji jest Mateusz Morawiecki, nie ma chyba na tej sali nikogo. Chyba że się mylę. Nie, nie mylę się niestety. Tak że w tej formule mini-mini, powtarzam raz jeszcze, mimo dość aroganckiego podejścia klub Lewicy będzie głosował za tym rządowym przedłożeniem. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam pana posła Krzysztofa Paszyka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Nieobecny Panie Ministrze Sprawiedliwości! W imieniu klubu Koalicja Polska podtrzymam pozytywną opinię co do istoty projektu rządowego zmieniającego Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie usprawnienia informatyzacji ważnego wycinka systemu sprawiedliwości, jakim jest Krajowy Rejestr Karny. Nie możemy dzisiaj, w XXI w., dalej hołubić zasady wymiany dokumentów papierowych, skoro można to usprawnić za pomocą systemów elektronicznych. Ale zgodzę się z przedmówcami, że po ostatnich latach praktyki i doświadczeń, jeśli chodzi o pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości, jest taka zasada przeniesiona z ruchu drogowego, zasada ograniczonego zaufania, i to jest fakt, wszyscy to odczuwamy.

Panowie, nie idźcie tą drogą, nie psujcie do końca tej legislacji, która tu w ostatnich miesiącach czy latach nie ma się najlepiej. Właśnie przez takie praktyki. Będziemy przyglądać się tym poprawkom, trzeba je dobrze przeanalizować.

Dziękuję panu serdecznie, panie pośle. Chciałem powiedzieć, bo chcę być uczciwy wobec wszystkich stron, że pan minister Marcin Romanowski słucha nas zdalnie. Oczywiście.

Panie Marszałku! Ja tym razem krótko. Jest to zmiana typowo techniczna i raczej powinna być dosyć oczywista. W oczywisty sposób należy usprawniać wszelki obieg dokumentów, a najlepiej się go usprawnia, właściwie likwidując dużą część z nich. Korzystając z okazji, że jest akurat dyskusja na ten temat konkretnie, akurat o dokumentach, chciałem państwu przypomnieć, bo często jest tak, że z mównicy sejmowej docierają pewne kwestie, że w tym momencie jest ustawowy obowiązek złożenia zaświadczenia o niekaralności w przypadku licencjonowanych pracowników ochrony, Straży Granicznej, pracowników kontroli skarbowej, doradców skarbowych, komorników, policjantów, nauczycieli, w tym także katechetów - jako nauczyciel z 15-letnim stażem nigdy tego nie rozumiałem, ale to jest na liście - prokuratorów, sędziów, agentów ubezpieczeniowych, detektywów. Myślę, że połowę tej listy można by z tej ustawy wywalić. Rozumiem, że wymóg niekaralności może funkcjonować u służb mundurowych, tych, które dbają o nasze bezpieczeństwo, czy w sądownictwie, natomiast cała reszta jest jednak sektorem prywatnym i w tym sektorze prywatnym tego typu ograniczeń nie powinno być.

Tak jak mówiłem, jest to projekt techniczny i dobrze, że chociaż coś będzie lekko usprawnione. Dziękuję bardzo. Czy jest pan poseł Michał Szczerba? Pan poseł Mirosław Suchoń? Też nie widzę. W związku z tym łączymy się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości panem Marcinem Romanowskim. Panie ministrze, czy pan jest? Jest pan. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak rzeczywiście zostało to zauważone przez szanownych państwa posłów, istotnym przedmiotem jest tutaj zmiana w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jeżeli chodzi o przesłanki, to obecnie, od kilku lat liczba zapytań, wniosków do Krajowego Rejestru Karnego łącznie - bo mamy tutaj do czynienia z jednej strony z Warszawą, z drugiej strony z punktami informacyjnymi w całej Polsce - wynosi 3 mln, od wszystkich podmiotów liczonych łącznie.

Zwrócę uwagę, że obecnie średni czas udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski wynosi prawie 19 dni.

Odpowiadając też na uwagę dotyczącą delegacji ustawowej, chciałbym zwrócić uwagę, że to było przedmiotem naszej pracy. To była uwaga czy też poprawka pana posła Zimocha.

Oczywiście tutaj można mieć inne zdanie, dyskutowaliśmy rzeczywiście nad tym na posiedzeniu komisji, ale w ostateczności myślę, że wspólnie z Biurem Legislacyjnym uzyskaliśmy tutaj wspólne stanowisko odpowiadające brzmieniu aktualnego przedłożenia. Tak że jestem przekonany, że ten projekt, jeżeli stanie się obowiązującym prawem, da możliwość opatrywania zaświadczeń kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i rzeczywiście umożliwi to pełne zautomatyzowanie procesu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie przedstawionego projektu. Bardzo dziękuję. Poseł sprawozdawca, pan poseł Piotr Sak, prosił jeszcze o głos. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Dziękuję serdecznie za wszelkie słowa, spostrzeżenia i uwagi, zwłaszcza te krytyczne. Dziękuję za wniesione poprawki. Oczywiście one będą ulegać dalszemu wartościowaniu, walidacji na dalszym etapie prac legislacyjnych. Muszę, mam wewnętrzny imperatyw, żeby odnieść się tutaj do słów pana posła Zimocha, który starał się mnie tutaj zmitygować, skonfundować swoją wypowiedzią.

I jak pan wie doskonale, moje poprawki odnosiły się do zapisów po art. 3 i dlatego była ta kwestia zasygnalizowana. Niezależnie od tego, panie pośle, zanim tak naprawdę te poprawki zostały przeze mnie ustnie zgłoszone, trafiły one już poprzez pracowników komisji do wszystkich posłów. Tym bardziej wypełniłem w tym zakresie obowiązek wynikający z art. 42 regulaminu Sejmu, który wskazuje, kiedy należy zgłaszać poprawki. Dlatego ta uwaga jest absolutnie zbędna, jałowa i niepotrzebna. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, na podstawie art. 95 ust. 2 regulaminu Sejmu kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu przedstawienia sprawozdania. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki nr 732 i 821) Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, druki nr 732 i 821.

Te poprawki nie uzyskały akceptacji komisji. Natomiast komisja w nosi o uchwalenie sądowego przedłożenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i Jako pierwsza zdalnie głos zabierze pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i

Ponieważ nie ma połączenia z panią poseł, głos zabierze pan poseł Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska. Nie ma pana posła. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, klub Lewica. Bardzo proszę pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Lewicy przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy Kodeks postępowania karnego, druki nr 732 i 821. Jak czytamy w przedłożeniu, projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt ustawy wprowadza zmiany do Kodeksu postępowania karnego, które uściślają i doprecyzowują obowiązujące już obecnie przepisy odnoszące się do gwarancji procesowych przysługujących osobom pokrzywdzonym. Konieczność wprowadzenia tych zmian wiąże się z wykonaniem zobowiązań wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego oraz Rady ustanawiających normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Zmiany te mają uwzględniać wnioski Komisji Europejskiej w związku z naruszeniem procedur dotyczącym niepełnego wdrożenia wspomnianych dyrektyw. W polskim prawie przepisy obecnie zawarte w Kodeksie postępowania karnego realizują już większość postanowień ze wskazanych wcześniej dyrektyw, m.in. prawo pokrzywdzonego do informacji o przysługujących mu uprawnieniach oraz do informacji na temat postępowania, prawa do tłumaczenia, w tym złożenia zawiadomienia o przestępstwie w języku, którym pokrzywdzony włada, do bycia wysłuchanym, do pomocy prawnej, do zwrotu poniesionych kosztów, do odszkodowania, do środków ochrony, a ponadto w Kodeksie karnym wykonawczym - w zakresie dotyczącym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Chodzi o zapewnienie środków pomocy dla pokrzywdzonych, w tym pomocy materialnej oraz niematerialnej w postaci porad prawnych oraz psychologicznej. Co prawda już sam sposób realizacji wspomnianych zapisów ustawowych pozostawia na dzień dzisiejszy wiele do życzenia, zwłaszcza chodzi tu o sposób dysponowania i cele, na jakie faktycznie przeznaczane są środki z tzw. funduszu sprawiedliwości, które - mówiąc delikatnie - są mocno kontrowersyjne. Raport NIK stwierdza wręcz wprost, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewniło adekwatnej i skutecznej pomocy ofiarom przestępstw. Wracając do przedłożenia, chcę powiedzieć, że w odniesieniu do kolejnej z dyrektyw jej przepisy również znajdują odzwierciedlenie w szeregu ustaw, w tym w Kodeksie karnym w zakresie dotyczącym przestępstw na tle seksualnym czy w Kodeksie postępowania karnego w odniesieniu do praw pokrzywdzonych dzieci, w tym co do szczególnego trybu przesłuchania, nagrywania takich przesłuchań czy ich fakultatywności, a także w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizującej zapisy tzw. konwencji antyprzemocowej. Wiele z obecnie obowiązujących w naszym kraju przepisów daje wsparcie niezbędne z perspektywy osób pokrzywdzonych. To wsparcie i ochronę, dziś gwarantowane prawem, które mogłyby się wydawać czymś oczywistym i podstawowym, zyskaliśmy dzięki dostosowaniu polskiego prawa do prawa unijnego właśnie. Dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej poprawia się nie tylko stan naszej infrastruktury drogowej, kolejowej, zyskują nie tylko dofinansowane gminy, nie tylko docieplone, rozbudowane szkoły, ale też nasze prawo staje się lepsze, a w tym konkretnym przypadku - osoby poszkodowane przestępstwem zyskują lepszą ochronę prawną. Polska w Unii Europejskiej to nie tylko dodatkowe środki finansowe na ochronę zdrowia, jak te z Funduszu Odbudowy, czy na środowisko z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to nie tylko znane wszystkim, chociażby ze słyszenia, dopłaty dla rolników, ale to też to, o czym czasem zdajemy się zapominać na co dzień: lepsza ochrona naszych praw, praw człowieka, ochrona praworządności. Ponieważ proponowane zmiany w przepisach zmierzają do pełniejszego wykonania prawa unijnego, a w konsekwencji - do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych, klub Lewicy popiera niniejsze przedłożenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Czy pan poseł Krzysztof Paszyk jest na sali?

Czy głos będzie chciał zabrać podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Marcin Romanowski? Bardzo proszę sprawozdawcę komisji pana posła Marka Asta. Wysoka Izbo! Chciałbym przede wszystkim podziękować za rzeczową dyskusję w ramach komisji. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, więc nie wzbudzał kontrowersji. Jeszcze raz serdecznie wszystkim członkom komisji dziękuję. Dziękuję za uwagi do projektu, wszystkie głosy i oczywiście w imieniu komisji wnoszę o uchwalenie przedmiotowego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam teraz 10 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druki nr 809 i 835) Bardzo proszę panią poseł Iwonę Arent o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, druk nr 809 i druk nr 835. Marszałek Sejmu skierował do naszej komisji przedkładany projekt. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po przeprowadzeniu pierwszego czytania rozpatrzyła projekt. Podczas rozpatrywania zostały zgłoszone poprawki. Poprawka nr 2 wynika z konieczności uzupełnienia projektowanych przepisów o ministra właściwego do spraw geologii w związku z wyodrębnieniem tego działu administracji rządowej ustawą z dnia 20 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Poprawka nr 3 to poprawka wynikająca z konieczności doprecyzowania terminu wydawania opinii, o której mowa w przepisie. Poprawka nr 4 jest związana z uchyleniem pkt 23 w art. 77 ust. 5. Poprawka 5. służy poprawnemu wyrażeniu początkowej woli projektodawcy.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Janusz Kozik, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, druk sejmowy nr 809, jest wykorzystanie potencjału Bałtyku w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z wiatru oraz stworzenie norm prawnych, które w perspektywie wielu lat pozwolą na realizację projektów inwestycyjnych oraz budowę nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Chciałbym podkreślić znaczenie przedkładanego projektu nie tylko dla sektora energetycznego, ale szerzej - i dla całej gospodarki, w szczególności w okresie odbudowy naszego potencjału gospodarczego po pandemii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło we wrześniu zaktualizowany projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Jednym ze strategicznych i priorytetowych kierunków wskazanych w tym dokumencie jest program inwestycyjny budowy morskich farm wiatrowych o wartości ok. 130 mld zł, który doprowadzi do uzyskania ok. 11 GW mocy zainstalowanej do 2040 r. w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej w obszarze Bałtyku oraz powstania ok. 77 tys. nowych miejsc pracy. Kluczowe jest to, aby morskie farmy wiatrowe powstały z jak największym udziałem polskich przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw, w szczególności przedsiębiorstw branży stoczniowej i portowej. Szacowana wartość projektowanych inwestycji nie ma precedensu w historii, co oznacza duże korzyści dla gospodarki, a także wpływy do budżetu państwa. Największymi beneficjentami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej będą stocznie, porty, przemysł stalowy i metalowy, przemysł maszynowy, sektor transportowy i usługowy. Wiele z nich już teraz bierze aktywny udział w zagranicznych projektach budowy morskich farm wiatrowych, ale też są takie, które dopiero planują włączyć się do tego obszaru działalności.

Model wsparcia przewidziany w ustawie opiera się na wypróbowanej w polskich realiach gospodarczych koncepcji tzw. dwustronnego kontraktu różnicowego, który z powodzeniem jest stosowany w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wsparcia OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy wejdą do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie różnicy między rynkową ceną energii a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Jeśli mogę jeszcze, pani marszałek, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, druki nr 809 i 835, bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy, po doręczeniu ich posłom. Do przedstawienia wniosku zostałem upoważniony. Bardzo proszę, pan poseł Sławomir Neumann. Przepraszam, pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Rząd nie zauważył, że przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować i budować morskie farmy wiatrowe, mają problemy z planem zagospodarowania obszarów morskich, że postępowanie związane z pozwoleniem na budowę sztucznych wysp trwa i są problemy, że są problemy z przyjęciem warunków przyłącza i z całym procesem administracyjnym związanym z wydawaniem decyzji, który się przedłuża.

Dziś Polska potrzebuje rozwoju dużych niskoemisyjnych źródeł wytwórczych zwiększających udział OZE w miksie energetycznym.

Bardzo proszę, pan poseł Sławomir Neumann, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Już kilka miesięcy temu podpisano list intencyjny między (Dzwonek) władzami samorządowymi, naukowcami, biznesem dotyczący tego, żeby, korzystając z tej ustawy, móc wprowadzić tę politykę jak najszybciej i zarabiać. To jest element zarabiania, nie tylko tańszej energii dla Polaków, ale też zarabiania przez polskie firmy dobrych pieniędzy w dobrym, nowoczesnym biznesie. Chciałbym, pani marszałek, zgłosić sprzeciw. Poprawki, które zostały złożone, powinny trafić do komisji. Tam też pewnie będą poprawki, więc nie ma powodu podchodzić do tego w taki sposób. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Beata Maciejewska, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jest to długo oczekiwana, bardzo potrzebna ustawa dotycząca rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. To jest bardzo ważny moment dla rozwoju, budowania nowoczesnej energetyki w Polsce.

Przypomnę, że Polska ma największy potencjał, jeśli chodzi o energetykę wiatrową na Bałtyku.

Przede wszystkim ma wpływ na to, co stało się kilka dni temu, a mianowicie na to, że Unia Europejska wyznaczyła nowy, 55-procentowy cel redukcji emisji

Nie może być tak, że Polska, mając tak ogromny potencjał polskiego wiatru na Bałtyku, może sobie odpuścić te kwestie i pozostać z tyłu. Jako Lewica będziemy głosowali za tym projektem. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Szanowny Panie Ministrze! Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze wspierało rozwój energetyki odnawialnej. To rząd, który współtworzyliśmy, i nasz minister gospodarki wpierw Waldemar Pawlak, później Janusz Piechociński przygotowali kluczową dla rozwoju branży ustawę o odnawialnych źródłach energii. Jak tylko władzę przejęła obecna władza, zaczęła niszczyć te podwaliny dla rozwoju OZE, które my budowaliśmy przez lata. Za naszych rządów energetyka wiatrowa rozwijała się w Polsce jak nigdzie indziej w Europie, szanowni państwo. Nowe projekty nadal nie mogą być rozwijane przez tzw. ustawę odległościową. Tysiące ludzi wtedy straciło pracę.

To te farmy wiatrowe, które powstały, nieprzerwanie produkują prąd, chroniąc nasze środowisko naturalne, zmniejszając kary, które Polska musi płacić za niespełnienie umów, na jakie się zgodziliśmy.

Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Procedowana ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ma swoje wady. Wiemy o tym doskonale, bo rozmawiamy z inwestorami. Ale wiemy od nich także, że jeżeli jej dzisiaj nie uchwalimy, to możemy zapomnieć o energii elektrycznej z farm na Bałtyku za 5 lat, a zatem i o transformacji energetycznej, i o pieniądzach z Unii. A nasza gospodarka bardzo tej energii potrzebuje. I potrzebuje też tych miliardów, miliardowych inwestycji w farmy na morzu, bo one dadzą rozpęd polskim przedsiębiorstwom, które już od lat eksportują produkty i usługi na rynki, gdzie energetyka wiatrowa rozwija się bez takich barier, jakie wy, państwo, u nas stworzyliście. Gdybyście w 2016 r. nie zaczęli walki z wiatrakami, tylko kontynuowali to, co my zaczęliśmy budować, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. W oparciu o inwestycje w Polsce rozwijałby się dalej krajowy łańcuch dostaw.

Ale tego czasu nie mamy. Inwestorzy jak najszybciej muszą wiedzieć, w jakich ramach mają działać, a to określają rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Odpowiednie wnioski muszą zostać złożone do prezesa URE do końca marca przyszłego roku, szanowni państwo. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za gospodarkę naszego kraju w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej informuję, że będziemy głosować za. Bardzo proszę, abyśmy tę ustawę jak najszybciej przyjęli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja.

Dziękuję bardzo, panie pośle.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po pierwsze, powstaje nowy gigant, do którego trzeba będzie dopłacać tak samo jak do Centralnego Portu Lotniczego, który być może nigdy nie powstanie. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, tu Lewica mówi, że się tworzy miejsca pracy. Gdyby zamiast hutnictwa zrobić dymarki, to ilość miejsc pracy by wzrosła jeszcze bardziej. Jeszcze raz: celem gospodarki jest zmniejszenie ilości miejsc pracy, a nie zwiększenie ilości miejsc pracy.

Powiedzcie tutaj Polakom, o ile drożej będziemy płacili za energię elektryczną, dlatego że ona nie jest z węgla czy nie jest z atomu, tylko jest z farm wiatrowych, oczywiście o ile one kiedykolwiek powstaną, bo na pewno powstanie przedsiębiorstwo, które je będzie robiło, i będą w nim pensje, premie itd., to jest oczywiste. Polak powinien wiedzieć, ile to będzie nas kosztowało. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Minuta na zadanie pytania. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak wygląda plan zagospodarowania Morza Bałtyckiego? Dlaczego firmy, które mamy w wykazie. Tak naprawdę ta ustawa jest szyta pod te firmy. Część z nich zdecydowała się na inwestycje w pasie przygranicznym ze Szwecją, co straszliwie wydłuża proces akceptacji, uzgodnienia środowiskowe itd. Czy mamy wolne przestrzenie dla firm innych i czy będziemy wpuszczać na teren Morza Bałtyckiego również firmy spoza Unii Europejskiej, z określonym kapitałem, po to żeby zrealizować cel 55%? Jak wygląda spięcie finansowe tych inwestycji, które są w tej chwili realizowane przez podmioty, które są związane z tą ustawą? Jak będzie wyglądało wsparcie coroczne opłaty OZE właśnie dla energetyki [[Dzwonek]] wiatrowej? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Muszę powiedzieć, że jak żywo mam przed oczami obraz sprzed 5 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość de facto zabijało energetykę wiatrową, przyjmując absolutnie niekorzystne przepisy w tym względzie. Dzisiaj na sali nie widzę nikogo, kto wtedy tutaj wychodził i bardzo stanowczo stał za projektem, który niszczył ten ważny sektor, który z jednej strony stanowił o gospodarce, ale z drugiej strony zapewniał bezpieczeństwo energetyczne. No tak, no to jest właśnie hipokryzja i całkowite pomieszanie po tej stronie rządowej.

Natomiast co z firmami prywatnymi, niezależnymi, które by chciały wejść na ten rynek? Widać wyraźnie, że jest tutaj jednak [[Dzwonek]] wsparcie wyłącznie dla tych, którzy są powiązani prawdopodobnie z większością. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Te 11 GW w przyszłości z wiatru na morzu to jest to, na co czekaliśmy. Kiedy 5 lat temu spytałem ministra odpowiedzialnego za sprawy energetyki, jak wyobraża sobie odnawialne źródła energii, kogenerację, to on odpowiedział mi w ten sposób: wiecie państwo, chcielibyśmy mieć w jednym ręku wytwarzanie, przesył i regulację. Od tamtego czasu przeszliśmy kawał drogi w kierunku prawidłowego rozwoju energetyki, tego miksu energetycznego i za to, mimo że są spóźnienia, dziękuję.

W związku z tym mam pytanie: Czy sieci, które są w chwili obecnej, planowane wiatraki, są wystarczające, żeby ten przesył był sprawny, żeby można było to przesłać? Po drugie, jest też oczywiście pytanie dotyczące planowanej energetyki atomowej. Czy to nie jest w kolizji? Czy moce, czy możliwości przesyłowe są wystarczające, żeby lokalizować dwa typy energii: wiatrowej na morzu i energetyki potencjalnie atomowej, która jest w naszych planach? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przemawiam tu jako energetyk. W związku z tym wiem, że kluczową sprawą w systemie energetycznym naszego kraju są właśnie sieci przesyłowe i sieci dystrybucyjne, na co zwrócił uwagę mój przedmówca. W związku z tym mam pytanie do pana ministra: Czy za tym ambitnym planem budowy elektrowni wiatrowych na morzu nadążą inwestycje polskich sieci energetycznych? Bo wiemy, że dzisiaj to jest kluczowa sprawa, żeby tę energię do polskiego systemu można było wprowadzić. Rzecz druga. Czy rząd planuje w tym zakresie przygotowanie projektu tzw. ustawy korytarzowej? Bo energetycy borykają się z wieloma problemami dotyczącymi zgód, dotyczącymi wszystkich planów itd. Jeżeli tego w jakiś sposób nie skrócimy, to będzie niestety w ogóle problem ze skorelowaniem i z wybudowaniem (Dzwonek) farm na morzu i z wprowadzeniem tej energii do systemu przesyłowego i później dystrybucyjnego w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Skoro jest refleksja, to ja chciałbym zapytać o krok dalej.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Gdyby tak się pokusić o nazwanie czy ocenę polityki PiS wobec OZE, to przychodzi tylko jedno do głowy: walka z wiatrakami.

Chcecie zwyczajnie osiągnąć ten efekt OZE w postaci spalania polskich lasów. Tak samo jesteście nieskuteczni w walce z polityką Unii Europejskiej w zakresie (Dzwonek) odnawialnych źródeł. Najpierw walczyliście z celem 40-procentowej redukcji, a teraz zgodziliście się na 55-procentowy. Tylko jak go chcecie osiągnąć? Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Paweł Papke, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy mówi o precyzyjnym rozdzieleniu pierwszej i drugiej fazy systemu wsparcia.

Wyróżniono dwa sposoby przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda. Czym podyktowana jest ta data? Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dlatego mam pytanie: Jak zmieni się rynek pracy po wprowadzeniu tej ustawy? Ile powstanie nowych miejsc pracy? Pragnę również dopytać przy okazji tej ustawy o znakomity program, bo mam wrażenie, że opozycja całkowicie o tym zapomina, o program „Mój prąd” Energia wiatrowa będzie miała swój udział w miksie energetycznym. A jak na dzień dzisiejszy wygląda realizacja tego programu? Jaki jest dzisiaj udział w miksie energetycznym prądu wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne, bo widzimy, że praktycznie w tej chwili na co drugim - może przesadzam - ale na bardzo wielu budynkach montowane są panele? Mam też pytanie: Jak to wyglądało za czasów [[Dzwonek]] naszych poprzedników? Pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska.

Ale, panie ministrze, pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw OZE. Kiedy pierwszy prąd popłynie właśnie z tych farm wiatrowych? Jak będziemy realizować ten wskaźnik, który został narzucony, którzy sami sobie narzuciliśmy - 21% OZE do 2030 r. Kolejne pytanie. Obiecaliście Polakom, że będą rekompensaty za prąd. Chciałbym pana zapytać, czy Polacy, którzy liczyli na to, którym obiecywaliście [[Dzwonek]] rekompensaty za podwyżkę prądu, energii elektrycznej, otrzymają tę rekompensatę, a jeśli tak, to kiedy. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Niestety w 2016 r. wykończyliście w Polsce energetykę wiatrową.

Niestety Polska jest na szarym końcu. W Danii mamy 41% energii z energetyki wiatrowej, w Niemczech - 21%, w Polsce - zaledwie 8%. Teraz próbujecie się za to zabrać i coś tam poprawiać. Natomiast zgodnie z założeniami tej unijnej dyrektywy podmioty, które będą chciały skorzystać z tej ustawy, będą musiały złożyć wnioski do 31 marca. To jest wyjątkowo mało czasu. Chciałbym zapytać, dlaczego tak późno zabraliście się za procedowanie nad tą ustawą i czy taki termin na składanie wniosków nie wpłynie negatywnie na powodzenie tej ustawy. Czy może tak naprawdę chodzi o to, żeby przyszli przedsiębiorcy nie złożyli tych wniosków i żeby dalej opierać się na węglu? Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowni Państwo!

Czy państwo jako wnioskodawcy przewidzieli rozwiązanie też tego problemu? Jeśli tak, to w jaki sposób? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie ministrze, udało mi się dobiec i słyszałem, jak koleżanka z PiS-u pytała pana o nowe miejsca pracy. A ja zapytam o stare miejsca pracy.

To jest fabryka, która miała w swoim zamiarze budować fundamenty pod farmy, podwodne farmy wiatrowe. Czy ona jest również w tym projekcie zawarta i czy wreszcie ludzie zaczną w niej pracować, bo jest to majątek, potężny majątek, za potężne miliony, który stoi pusty? Drugie pytanie.

Również był pan w Świnoujściu, rozmawiał pan o rozwoju portu świnoujskiego jako dedykowanego do wiatraków. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie dotyczące konkurencyjności polskiej gospodarki, mianowicie ogromną częścią kosztów przemysłu są koszty energii elektrycznej.

Pragnę również przytoczyć pewien przykład, zły przykład, ale niestety miało to miejsce. Mianowicie prezydent Warszawy pan Rafał Trzaskowski niedawno, jakiś czas temu wybrał koreańskie tramwaje zamiast tramwajów z bydgoskich, polskich zakładów PESA. Pragnę zapytać, czy ten sam sposób doboru, wyboru będzie premiowany przy budowie farm wiatrowych. Czy po prostu będą to budować polskie firmy, czy koreańskie, [[Dzwonek]] czy niemieckie? Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii pan Ireneusz Zyska. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Chciałbym również podziękować wszystkim państwu posłom za pracę w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w dniu wczorajszym. To też świadczy o wadze tego projektu, znaczeniu dla polskiej gospodarki. Mam niewiele czasu, a było bardzo dużo pytań, na które chciałbym odpowiedzieć.

Nie ma tutaj ograniczeń.

Pierwsza i druga faza wsparcia, pomocy publicznej, kontrakt różnicowy. Dlaczego do 30 marca, a decyzję prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wydać tylko do 30 czerwca? Wynika to bezpośrednio z treści dyrektywy RED II, która wskazuje, że od połowy przyszłego roku może obowiązywać tylko i wyłącznie system konkurencyjny w ramach aukcji OZE, podobnie jak ma to miejsce teraz w energetyce, jak stosujemy to w energetyce lądowej, różnych technologiach odnawialnych źródeł energii. Stąd też udzielanie pomocy publicznej w trybie administracyjnym może się zakończyć decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki tylko do 30 czerwca przyszłego roku. Są wśród nich również projekty z udziałem spółek Skarbu Państwa, ale także prywatnych podmiotów.

Myślę, że zadaje to kłam tym tezom, które państwo posłowie z opozycji próbowali przedstawić. Odnośnie do pytania pani poseł Anny Kwiecień powiem bardzo króciutko, bo nie dotyczy to samej ustawy. Drodzy państwo, nie zgadzam się z tezą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy z wiatrakami. Po pierwsze, w ramach aukcji OZE, które zostały przeprowadzone w roku 2018, roku 2019 i roku 2020, właśnie przed chwilą się skończyły, 3 grudnia, zostało zakontraktowane 4,2 GW mocy. w elektrowniach wiatrowych na lądzie.

Do tego dochodzi program „Mój prąd”, o który pytała pani poseł. Przekroczyliśmy 3,5 GW mocy zainstalowanej we wrześniu tego roku w instalacjach fotowoltaicznych. Do tego, drodzy państwo, jest ponad 360 tys. prosumentów.

Dzisiaj, proszę państwa, zbliżamy się do 400 tys. Proszę sobie porównać te wielkości. Tak że ta informacja lansowana przez państwa, że walczymy z wiatrakami, jest absolutnie nieprawdziwa. Powiem, drodzy państwo, co również jest bardzo ważne, że w 2016 r. były inne technologie.

To wielkie instalacje, które będą zasilać polską gospodarkę. Pan poseł Paweł Rychlik pytał o konkurencyjność. Dostęp do dużej mocy (Dzwonek) zainstalowanej, wytwarzającej tzw. zieloną energię poprawi sytuację polskich spółek produkujących, polskich podmiotów gospodarczych, które będą mogły eksportować na najbardziej lukratywne rynki europejskie i światowe polskie produkty z udziałem właśnie zielonej energii. Pani Marszałek! Nie wiem, czy byłaby zgoda, żebym jeszcze mógł kilka sekund przedłużyć.

Polska ma ogromny potencjał.

Myślę, że w kolejnych latach, pod koniec lat 20., na początku lat 30., wszystkie porty - zarówno zespół portów Szczecin-Świnoujście, jak i zespół portów Gdańsk-Gdynia, mniejsze porty takie jak Władysławowo, Ustka, które mogą być portami serwisowymi - będą miały swoją wielką szansę na realizację tych projektów, żeby obsługiwać morskie farmy wiatrowe.

Ma powstać również ponad 77 tys. nowych miejsc pracy, głównie na Pomorzu Środkowym, ale nie tylko.

Osiągniemy cel odnawialnych źródeł energii, cel OZE na rok 2030. Pomoże nam to również w osiąganiu celu związanego ze zmniejszaniem emisyjności gospodarki. Nawet rozumiem też głosy trochę uszczypliwe czy krytyczne ze strony opozycji, ale jak wszyscy podkreślali, jest to ustawa dobra, potrzebna dla Polski, dla naszego systemu energetycznego, dla polskiej gospodarki. Dziękuję za te pozytywne głosy. Bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie tego projektu ustawy w głosowaniu wraz z poprawkami, które zostały zgłoszone dzisiaj przez pana posła z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Miałem okazję, siedząc tutaj w ławie poselskiej, zerknąć na te poprawki. Uważam, że one są ze wszech miar pożądane i godne poparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono poprawki oraz wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 828, 828-A i 836) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. To bardzo proszę, ale nie zgłosił pan do sekretariatu. To bardzo proszę, panie pośle. Nie był pan zgłoszony, dlatego nie mam pana na liście. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie zmian w przedmiotowej ustawie wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania kolejnych sektorów gospodarki oraz wprowadzenia rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organów państwa. W art. 1 zmiany dotyczą kwestii wynagradzania pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zmiana w art. 15 wprowadza możliwość wypłacania świadczenia postojowego osobom, które dotychczas nie korzystały z tego świadczenia. Nowelizacja umożliwia utrzymanie ważności certyfikatów lotnisk w okresie obowiązywania stanu pandemii oraz nowych uprawnień dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tym okresie. Kolejne zmiany umożliwiają przekazywanie wsparcia operatorom kolejowych przewozów pasażerskich oraz przewoźnikom przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz przedłużenia okresu obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych. Nowe przepisy umożliwiają przekazanie środków finansowych w kwocie 120 mln zł na wsparcie branży kinematograficznej. Wprowadzone zmiany dotyczą także obniżenia wysokości kosztów pozaodsetkowych kredytów w czasie pandemii. W art. 4 wprowadzono zmiany dotyczące wojskowych komisji lekarskich. W art. 7 zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgłosił do omawianego projektu ustawy poprawki, które komisja zaopiniowała pozytywnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Teraz pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Sprawdziłem, jak było z tymi ustawami COVID-owymi w ostatnim czasie. 26 listopada br. słyszeliśmy takie słowa: Dzisiaj wdrażamy tarczę 2.0. Dodał, że pomoc ma objąć m.in. turystykę, gastronomię i kulturę. 10 grudnia, zaledwie 2 tygodnie później, padły kolejne zapowiedzi: Dla przedsiębiorców najbardziej zagrożonych branż proponujemy nowe instrumenty wsparć.

Nie znalazłem tarczy 3.0, nie znalazłem tarczy 4.0, nie znalazłem tarczy 5.0. Ale nie o tarczę tutaj chodzi. Tutaj chodzi tak naprawdę o to, czy jest realna pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych drugą falą epidemii koronawirusa, poszkodowanych wyłączeniem całych sektorów gospodarki decyzjami administracyjnymi rządu. Tego wsparcia po prostu nie ma. Opowiadacie państwo o kilkudziesięciu miliardach pomocy, która tak naprawdę jest tylko w przekazie propagandowym polityków Prawa i Sprawiedliwości, a w rzeczywistości nie istnieje. Natomiast co mamy w tej tarczy, w tej ustawie COVID-owej, bo trudno ją nazwać tarczą, która została złożona do Sejmu? To oczywiście z COVID-em nie ma nic wspólnego, ale pokazuje, że państwo po prostu wykorzystujecie każdy taki element do tego, aby cokolwiek, co leży w szafkach ministerialnych, w gabinetach ministerialnych, wykorzystać i wrzucić do tego jednego wora, bo wiadomo, że jest to przyjmowane w specjalnym trybie. Realnego wsparcia jest faktycznie 120 mln zł: na kinematografię, na stypendia, na promocję filmów, na dokończenie produkcji filmów, które zostały uruchomione. Tak naprawdę to jest jedyny element wsparcia dla sektora kultury, który w tej tarczy został uwidoczniony. Reszta to bliżej niedookreślone finansowanie. Co prawda ustawa daje możliwość przyznania rekompensat dla PKP PLK za obniżone dochody z tytułu korzystania z infrastruktury kolejowej, co prawda jest możliwość przekazywania dotacji na przewozy kolejowe czy dopłaty do przewozów autobusowych, ale gwarancji finansowej tutaj nie ma.

Przecież to jest niepojęte. W czym gorsi są ci, którzy świadczą usługi na rzecz samorządów?

Dlatego dzisiaj złożyliśmy na ręce pani marszałek konkretny projekt ustawy, która jest realnym wsparciem dla tych, którzy są najbardziej pokrzywdzeni, która pokazuje możliwości finansowania szeregu przedsięwzięć, w szczególności w zakresie ochrony miejsc pracy. Dodatkowo do przedłożenia rządowego, do ustawy, o której jest mowa, składamy kilka poprawek. Te poprawki dotyczą gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z poręczeń czy gwarancji spłaty kredytu. Wprowadzamy możliwość. Naprawdę to nie jest czas i pora, aby podmioty, które borykają się z gigantycznymi problemami, dzisiaj zajmowały się tym, aby mieć kasę fiskalną od 1 stycznia. I wreszcie również wprowadzamy poprawką możliwość odsunięcia w czasie, możliwość wliczania w koszty nietrafionych pożyczek, tak jak to mają banki, tak jak to mają SKOKI.

Dlatego to jest pakiet naszych poprawek do tej ustawy. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, chcąc poprawić los ludzi przynajmniej w tym zakresie, te poprawki uwzględnią, o co bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Widać, że święta za pasem, bo rząd zaserwował nam projekt ustawy, który jest jak bigos - pełen rozmaitości. Tutaj nawet kwestia trwającej pandemii nie jest żadnym spoiwem łączącym poprawki, łączącym te nowele, bo niektóre w ogóle nie dotyczą kwestii związanych z potrzebą dostosowania przepisów do tej szczególnej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Nawet Biuro Legislacyjne zwracało uwagę na wyjątkowy rozrzut tematyczny tych regulacji. W tym krótkim wystąpieniu chciałabym zwrócić uwagę na trzy kwestie z wielu poruszanych w tej ustawie. Kwestia pierwsza. Odrzucono na posiedzeniu komisji nasze poprawki, które uniemożliwiały używanie nadzwyczajnych przepisów do manipulowania czasem pracy i wskazywania miejsca odpoczynku dla pracowników. Pod przykrywką pandemii chcecie zamienić Polakom miejsca pracy w obozy pracy. To niedopuszczalne. Lewica stoi i zawsze będzie stała po stronie pracowników, i nigdy nie zgodzi się na takie prawo. Czy naprawdę chce pan pozbawić polskich pracowników praw i godności? Jeżeli tak, to proszę to powiedzieć dzisiaj Polkom i Polakom prosto w oczy tutaj, na tej sali. Lewica zgłosiła w tej sprawie wniosek mniejszości. Kwestia druga. Zgłaszaliśmy poprawki wstrzymujące eksmisje w czasie pandemii i również je odrzuciliście.

W czasie pandemii ludzie muszą czuć się bezpiecznie. Jeśli władza chce teraz kogokolwiek wywłaszczać, to powinna mieć obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego o tym samym metrażu i w tym samym standardzie. I wreszcie kwestia trzecia dotycząca przewozów autobusowych. Myślę, że to dobrze, że wreszcie dostrzeżono potrzebę dofinansowania tej gałęzi publicznego transportu. Szkoda tylko, że państwo znowu zrobiliście to po swojemu, bez konsultacji ze specjalistami. Oparliście dopłaty na dofinansowaniu utrzymania linii komunikacyjnej, co według ekspertów doprowadzi do sztucznego utrzymywania linii z jednym połączeniem w tygodniu w celu otrzymania dopłaty.

Nie ma informacji, co z nowymi liniami, które wcześniej nie funkcjonowały. Czy dostaną wsparcie, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Składamy teraz na ręce pani marszałek w tym zakresie poprawkę. Sensowne wsparcie dla tej branży jest potrzebne, bo pomoże przetrwać przewozom autobusowym, których funkcjonowanie będzie konieczne także do tego, by realizować „Narodowy program szczepień” Bo jak już program ruszy, to osoby z mniejszych miejscowości, zwłaszcza starsze, muszą mieć jakąś możliwość dojechania na szczepienie, a autobus to często jedyne połączenie komunikacyjne, które jest dostępne dla tych mieszkańców. Apeluję w tym miejscu do większości parlamentarnej. Bardzo proszę, przyjrzyjcie się zgłaszanym poprawkom, bo one są po prostu korzystne dla Polek i Polaków. Dziękuję. Dziękuję za poprawkę. I bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! W pierwszych słowach chciałbym się odnieść do tego, nad czym procedujemy, czyli do druków nr 828 i 828-A.

Podzieliśmy ich, szanowni państwo, czym? A dzisiaj życie pokazuje, że w wielu obszarach, szanowni państwo, dzieją się ludzkie tragedie. Z dobrych słów, które mogę powiedzieć, szanowni państwo, jeżeli chodzi o ten wniosek - dobrze, że wreszcie państwo pomyśleliście o transporcie kołowym, o przewozach autobusowych.

Myślę, że to jest przeoczenie, może jeszcze będziecie mogli państwo to naprawić. Dobrze, że mówicie o kolejach, mówicie o lotniskach.

Zostały zamknięte hotele, uzdrowiska, z wielu małych sklepików przesunęliśmy się do dyskontów, Biedronki, Lidla, nie wiadomo gdzie jeszcze, a te hurtownie, szanowni państwo, zatrudniają ludzi, ba, mają umowy z rolnikami, które są obwarowane odbiorem towarów w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie. Dlatego, szanowni państwo, w imieniu klubu Koalicja Polska składamy szereg poprawek, które uwzględnią te obszary funkcjonowania naszego państwa, które państwo pominęliście, nie wiem, czy z chytrości, zawiści, ale to również są nasi przedsiębiorcy, którzy każdego roku w normalnych warunkach płacą podatki, inwestują, chcą się rozwijać, ale chcą również myśleć o przyszłości.

Ludzie masowo likwidują swoje firmy.

Dlatego, szanowni państwo, pozwolę sobie jeszcze raz w imieniu Koalicji Polskiej złożyć poprawki do przedłożonego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Nikt już nie pamięta, która to jest już nakładka i na którą tarczę.

Z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że od ostatniego wystąpienia na ten temat w czasie poprzedniej sesji, w którym wyliczałem kraje w Europie, które zdążyliśmy już przegonić pod względem liczby zmarłych na COVID, przegoniliśmy kolejnego rywala, czyli Holandię, a więc tak jak mówiłem od początku, ostatecznie wszyscy osiągniemy podobne wyniki, tylko niektórzy kosztem większym, a niektórzy mniejszym. Cała ogromna ofiara poniesiona przez gospodarkę, przez bankrutujących obywateli na wiosnę służyła tylko odwlekaniu tego nieuchronnego, a w ostateczności zapewne wyjdzie na to samo.

Rząd dostrzega oczywiście uzasadnione potrzeby własnych organów przy opróżnianiu lokali przejmowanych na cele publiczne, kiedy tymczasem właściciele prywatnych lokali muszą często latami bujać się z niepłacącymi lokatorami, bo rząd często bardziej chroni intruza niż właściciela. Widać, że odległość od ucha ministra ma znaczenie. Zresztą przy okazji widać też, że gospodarka nakazowo-rozdzielcza, którą wszyscy od lat budują w naszym kraju, w trudnych sytuacjach jest po prostu niewydolna i wymaga natychmiastowych, ciągłych zmian regulacji, bo bez tych zmian, bez nowych ustaw wszystko by się poprzewracało w okolicznościach, których rząd nie przewidział. To jest też przestroga, że wszelkie sztywne regulacje w nieprzewidzianych okolicznościach powodują tylko problemy, a rządowi często wydaje się, że wie wszystko o tym, co próbuje uregulować, a w rzeczywistości jego wiedza jest zazwyczaj niewielka.

Pasażer w komunikacji bardziej przeszkadza, niż pomaga, i tak większość pieniędzy pochodzi z dotacji od miasta, a nie z biletów, więc akurat pomaga się tym, którzy najmniej tego potrzebują.

Naprawdę zwątpiłem w sens istnienia tej komórki.

Po co? Na koniec: w uzasadnieniu bardzo ucieszyło mnie to, że dostrzega się, że w kwestii gospodarki niepewność co do działań rządu tę gospodarkę paraliżuje, że rząd zauważa to, że jego trudne do przewidzenia ruchy powodują, że ludzie nie chcą inwestować, boją się inwestować, nie wiedzą, co ich czeka za chwilę, co rząd zamknie, a co rząd otworzy. Z tego powodu cała gospodarka cierpi. Proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Wysoka Izbo! Natomiast zwracam uwagę, że to, co robi rząd, z reguły daje skutki dokładnie odwrotne, niż rząd by chciał.

Póki my tracimy przez aktywność rządu w gospodarce, tracimy na to paręset miliardów rocznie, dzięki temu, że rząd coś robił w gospodarce, paręset miliardów, to tutaj giną ludzie. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwsza pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Komunikacja miejska, która jest współfinansowana przez samorządy, jest w bardzo trudnej sytuacji. Spółki miejskie, które zajmują się komunikacją, mają ogromne straty, a samorządy nie są w stanie im pomóc finansowo, bo COVID zrujnował tak naprawdę finanse samorządowe. Moje pytanie: Dlaczego - bo nie ma racjonalnego uzasadnienia - w tym projekcie ustawy komunikacja miejska została pozostawiona bez żadnego wsparcia, bez żadnej pomocy? Proszę o konkretną odpowiedź, żeby można było samorządowcom odpowiedzieć, dlaczego rząd tak postępuje. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście jest tak, że te kolejne tarcze w zasadzie nie wiadomo dlaczego są tak numerowane, bo te numery jakoś wyłamują się z kolejności i pojawiają się coraz wyższe, co nie odpowiada rzeczywistości. Ale rozumiem, że takie są prawa propagandy. Kwestia eksmisji. Panie ministrze, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego - wszyscy wiemy, że tam głównie chodzi o to, że ci, którzy zajmują wysokie stanowiska, kasują niezłe pieniądze. Natomiast wy chcecie wprowadzić przepisy, które w ramach epidemii będą pozwalały wywłaszczyć tych ludzi, którzy oczekują godnego traktowania i godnych odszkodowań. Druga rzecz - bon turystyczny. Rozszerzają państwo definicję tego bonu tak, że będą mogły z tego korzystać osoby w ramach imprez 1-dniowych, czyli np. organizatorzy pielgrzymek, ale uderzacie tym w miejscowości turystyczne oparte właśnie na pobycie. Dlaczego tak bardzo nie lubicie miejscowości turystycznych i co zrobicie dla przedsiębiorców z tych miejscowości, z Beskidów, z Tatr, żeby im pomóc? Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! To jest i tak mniej, niż wnioskował. Wskazujecie państwo w tej ustawie, że również przewoźnicy kolejowi i autobusowi mają otrzymać podobne wsparcie, przy czym nie ma kryteriów, które mogą - że tak powiem - pokazać tym firmom, jak to wsparcie miałoby wyglądać. Natomiast pominięta jest zupełnie sprawa lotnisk, które przeżywają duże trudności, i to niekoniecznie nawet z powodu tej sytuacji, ale również z powodu pewnych zaszłości, chodzi np. o odszkodowania z tytułu uznania, że lotniska są strefą, która wpływa na obniżenie wartości nieruchomości wokół strefy lotniskowej. Wydaje mi się, że te lotniska - np. lotnisko w Poznaniu - wymagają pilnej pomocy, bo jeżeli nie zatrzyma się w sposób ustawowo [[Dzwonek]] uregulowany tej sprawy, to może się okazać, że poziom roszczeń, toczące się sprawy plus odsetki spowodują, że to lotnisko, ten port lotniczy po prostu zbankrutuje. Bardzo proszę, pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie o szczegółową kwestię, mianowicie o oparcie dopłat dla branży autobusowej o dofinansowanie utrzymania linii autobusowej. Linia” daje bardzo wąskie pole do interpretacji, jako że odnosi się de facto do trasy przejazdu autobusu, a „sieć komunikacyjna” odnosi się do układu linii komunikacyjnych na danym obszarze. Jeśli w ramach sieci może dochodzić do zmian tras przejazdu, skróceń czy wydłużeń linii komunikacyjnych, to możemy wtedy nadal mówić o utrzymaniu tejże sieci, np. poprzez porównanie pracy eksploatacyjnej, tj. łącznej liczby wykonanych kilometrów. Skąd więc taki wybór, który przecież z perspektywy przewoźników, z perspektywy mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego jest niekorzystny? Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To jest kolejna ustawa dotycząca walki z pandemią czy zabezpieczenia polskich przedsiębiorstw w związku z pandemią. Jest tutaj wiele bardzo ważnych rozwiązań, natomiast mam pytanie: Dlaczego to jest kolejna ustawa, która pomija branżę gastronomiczną i branżę fitness? Codziennie pojawiają się informacje o tym, że zamykane są kolejne restauracje, że zwalniani są kolejni ludzie. Tej pomocy bardzo brakuje. Przecież obie te branże są gotowe do tego, żeby wprowadzić obostrzenia, restrykcje. Nie trzeba ich zamykać, nie trzeba zawieszać ich działalności, żeby były bezpieczne. Widać wyraźnie, że rząd w podejmowaniu decyzji o zamykaniu czy wyłączaniu tych branż nie oparł się na ekspertyzach, tylko [[Dzwonek]] jakichś bliżej nieuzasadnionych kryteriach. Pan poseł Maciej Lasek, Koalicja Obywatelska. Nie widzę pana posła. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Ta propozycja, którą przedstawiliście państwo, dotyczy również publicznej służby krwi. Chciałbym więc zadać pytanie, czy te rozwiązania, które dokonują zmian w tym zakresie, są wystarczające.

Czy były odpowiednie konsultacje z tą branżą? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Pierwsze moje pytanie jest takie: Dlaczego nie mogliście wszystkich tych regulacji i programów przyjąć w jednej ustawie, tak jak się robi w innych państwach europejskich, tylko musicie non stop coś poprawiać, zmieniać, kombinować? Dzisiaj pani poseł Pamuła z tej mównicy powiedziała, że nie ma w Polsce żadnych branż zamkniętych, żadnych branż wyłączonych. Pani poseł pluła dzisiaj tym wszystkim ludziom w twarz, twierdząc, że wszystko jest świetnie i wszystko jest otwarte. Wracając do ustawy: zakłada ona pomoc dla branży kinematograficznej, nomen omen też zamkniętej. Tak jak sugeruje np. prof. Simon, jest już przypuszczalnie między 4 mln, 6 mln a 10 mln ozdrowieńców, którzy mogliby bez żadnych rygorów sanitarnych z tego korzystać, dla reszty można by było wprowadzić jakiś reżim sanitarny. Skoro otwarte są kasyna i kościoły, a. Proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek, poseł niezrzeszony.

Wysoka Izbo! Ta ustawa jest napisana niechlujnie, a w dodatku krzywdzi ludzi.

To jest po prostu fatalny pomysł i ja bardzo proszę o wycofanie się z niego. Bardzo proszę, pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Chciałem zaprotestować przeciwko sformułowaniu, które pada z ust rządzących, o pomocy dla przedsiębiorców. Otóż przedsiębiorcy nie potrzebują żadnej pomocy, przedsiębiorcy potrzebują tego, żeby państwo im nie przeszkadzało, i wtedy doskonale sobie poradzą. Niestety państwo od lat przeszkadza im gąszczem biurokracji, regulacji, horrendalnymi podatkami, nakazami, zakazami, a w ostatnich miesiącach przeszkadza im w sposób wyjątkowo dotkliwy chaotycznymi, absurdalnymi obostrzeniami i faktycznym lockdownem. Rząd powinien wziąć za to odpowiedzialność i udzielić przedsiębiorcom rekompensaty, a nie pomocy. Zacznijcie uczciwie mówić o rekompensatach, a nie pomocy, nie róbcie z siebie łaskawców, nie róbcie z przedsiębiorców żebraków. Bo wy nie jesteście łaskawcami, jesteście winowajcami tej sytuacji, jak mówił Kisielewski: to nie kryzys, to rezultat, rezultat waszych decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja.

Wysoka Izbo! Jak już mówiliśmy ja i kolega Sośnierz, działania rządu nie przynoszą na ogół nic dobrego, a czasami nawet szkodliwe rzeczy, natomiast tracimy na tym miliardy, ale teraz chodzi o życie ludzkie.

W tej chwili ludzie nie umierają na COVID, na COVID umiera średnio mało ludzi, natomiast na inne choroby umiera o 1 tys. osób więcej niż normalnie. To wasze działania, to działania rządu.

Musicie coś robić. To wy macie krew na rękach.

Wysoka Izbo! Twierdzenie, że projekt nowelizacji ustawy COVID-owej nie zawiera żadnych konkretnych przepisów, które niosą za sobą rekompensaty negatywnych skutków pandemii, to nieprawda.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Dziękuje bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj znowu się zdziwiłem, bo muszę powiedzieć to samo, co koledzy z Konfederacji. Nie mówcie o żadnej pomocy, bo żadnej pomocy przedsiębiorcom nie dajecie.

Za to, że zrobiliście z tych ludzi nędzarzy, a oni harowali po 12, 14, 16 godzin w swoich małych firmach.

Jeszcze raz powiem: w Polsce padają wszystkie branże, bez względu na to, jaki [[Dzwonek]] mają numer, oprócz spożywczej, monopolowej i aptek. To będzie pierwsza prawdziwa pomoc. To będzie prawdziwa pomoc.

Panie i Panowie Posłowie! Trudne czasy epidemii, jakie dzisiaj mamy, to nie są czasy na wyrzucanie ludzi z domów z jakiegokolwiek powodu, a już tym bardziej z powodu jakichś megalomańskich inwestycji premiera Morawieckiego. Dlatego w szeregu poprawek, jakie złożyliśmy do tej ustawy, jedną z kluczowych jest ta, która wykreśla możliwość wyrzucania ludzi z domu w trakcie epidemii z powodu tego, że chcecie budować Centralny Port Komunikacyjny. Druga bardzo ważna poprawka dotyczy gastronomii.

Wszystkim jest bardzo ciężko.

Panie i Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Zawsze podczas dyskusji nad projektami ustaw, które są związane z pandemią koronawirusa, państwo z lewej strony sali staracie się wygłosić jakąś - co jeden, to mocniejszą - filipikę. Wysoka Izbo! Widać, jak niektórych to bardzo interesowało.

Świetnie. Jeżeli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, bo wokół tego się koncentrowała większa część tej dyskusji. Szanowni państwo, oczywiście wy zawsze macie świetne pomysły. To znaczy zawsze uważacie, że macie świetne pomysły. Oczywiście wychodząc na mównicę, tego powiedzieć nie możecie.

Bardzo proszę o spokój na sali.

Prawdą, której nie usłyszymy do was, jest to, że recesja w Polsce oczywiście jest, jest na całym świecie, ale w Unii Europejskiej jest najniższa właśnie w Polsce, szanowny panie. Tak, gratuluję zdrowego rozsądku przy takich wypowiedziach. Realna pomoc, której podobno nie widać. Tak jej nie widać, że ponad 160 mld już poszło na pomoc dla przedsiębiorców, ale tylko wyście jej nie zauważyli.

Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej i jesteśmy gotowi natychmiast rozpocząć tę pomoc.

Nie wiem, czy wiecie państwo, że w CEIDG od stycznia do grudnia tego roku zarejestrowanych zostało ok. 200 tys. nowych działalności. Co zaś się tyczy taksówkarzy, o których tutaj pytano, oczywiście, że zostali uwzględnieni, tylko - tak jak to już ktoś powiedział - państwo nie macie czasu przeczytać ustaw, państwo musicie się zajmować innymi rzeczami. Gdybyście przeczytali te ustawy, wiedzielibyście, że zwolnienie z ZUS dla nich zostało przygotowane. Niestety to z waszej strony padały te pytania.

A więc te wszystkie mechanizmy są w tym wypadku wdrożone. Czemu służy twierdzenie, że [[Dzwonek]] jakoby te ustawy są nieprzygotowane, że ciągle coś trzeba zmieniać? Miało być cały czas wszystko zamknięte? To chcecie państwo powiedzieć? To podajcie dobre przykłady. Podajcie przykłady krajów, w których wszystko zostało świetnie zrobione i na których moglibyśmy się wzorować. Bo wszyscy są w takiej samej sytuacji. Tylko jakoś nikomu dużo lepiej to nie wychodzi niż nam w Polsce.

Bardzo proszę pana ministra Andrzeja Bittela o udzielenie odpowiedzi na pytania. Ale jak sam pan minister zwrócił uwagę, ustawa została podpisana wczoraj, a problem z pomocą dla przedsiębiorców jest już prawie rok, niedługo będzie rok, więc dosyć późno ta pomoc przychodzi. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Pierwsza kwestia, którą chciałem poruszyć, to sprawy związane z pomocą dla sektora transportu zbiorowego i brakiem pomocy dla komunikacji miejskiej, jak tutaj zostało stwierdzone. Państwo pewnie wiecie, jestem o tym przekonany, że ustawa o ulgach, do której się odwołujemy w tych przepisach, nie dotyczy komunikacji miejskiej. Państwo wiecie, że samorząd terytorialny prowadzący komunikację miejską prowadzi własną politykę związaną z ulgami i ją finansuje. A więc z tych dwóch prostych i oczywistych powodów nie można tych zasad tutaj dopisywać i to jest oczywiste dla każdego, kto ma elementarną znajomość przepisów w tym zakresie. Zwracam uwagę, że rozszerzamy pomoc tam, gdzie są umowy związane z służbą publiczną, również o gminne i powiatowe linie - państwo tego nie dostrzegli, a warto to dostrzec - w transporcie kolejowym. Kryteria tej pomocy są znane i opisane w ustawie i trudno mi się zgodzić, że ich brakuje.

A więc warto to dostrzec. Ona nie jest zapisana w OSR. Tam w ustawie jest OSR, taka tabelka, tam dalej, gdzie jest mowa, że te pieniądze są zabezpieczone w budżecie na 2021 r., i zapewne państwo o tym wiecie już, bo budżet jest przecież przedmiotem obrad Wysokiej Izby. Szczególnie bolesne dla mnie osobiście, ale myślę, że dla każdego, kto ma elementarne poczucie odpowiedzialności za słowo i elementarną znajomość przepisów prawa, które są stosowane w przypadku procedur związanych z prowadzeniem inwestycji celu publicznego, z prowadzeniem inwestycji liniowych czy kubaturowych, ale przede wszystkim liniowych, bo o tych tutaj mówimy, są słowa o jakiejś zmianie, zabraniu prawa ludziom, których majątek ma być rzekomo odebrany. Może należałoby znać obecne brzmienie przepisu art. 15zzu, który mówi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Przepis ten był uchwalany przed okresem ochronnym. Jest okres ochronny, nie wolno ludzi wyrzucić na bruk w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego.

Zwykle rozwiązuje się to na wcześniejszych etapach.

Myślę, że pani marszałek pozwoli, bo to ważne. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, odrzucona propozycja lokalu zastępczego, odszkodowanie wypłacone w całości. Następny przykład, odrzucona propozycja lokalu zastępczego, odszkodowanie wypłacone w całości. Warszawa (Dzwonek), właścicielce zaproponowano refundację lokalu zastępczego, wypłacono zaliczkę w wysokości 70% wysokości odszkodowania. Ludzie mają prawo oczywiście domagać się słusznego odszkodowania, ale też trzeba realizować procesy inwestycyjne, tu nie ma kwestii masowej skali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, mówię do pana ministra Bittela, który teraz zmierza w kierunku wyjścia. Przecież my mówiliśmy wyraźnie, że chodzi o Centralny Port Komunikacyjny. Wie pan, co tam się dzieje w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego? To wie większość rządząca, cała opozycja, ale i chyba cała Polska. Tam głównie wysocy urzędnicy kasują co miesiąc bardzo wysokie wynagrodzenia, i to się dzieje w CPK.

To tam się dzieje i to jest przykre, i ja tego nie rozumiem, bo to pozwala (Dzwonek) stwierdzić, że rząd wykorzystuje sytuację, trudną sytuację.

Przepraszam, panie ministrze, może pani poseł, a potem pan minister, żeby już za jednym zamachem było. Bardzo proszę. Panie ministrze, komponent kolejowy CPK będzie dotyczył całej Polski, prawie wszystkich województw, więc co pan tutaj nam wciska, że to nie będą masowe eksmisje? Dziękuję. Bardzo proszę, pan minister Bittel zabiera głos. Dziękuję bardzo. Wiedziałem, że państwo będziecie oczywiście odnosili się do komponentu kolejowego i w ogóle do inicjatywy CPK, bo jej nie akceptujecie. Natomiast, jeżeli państwo chcecie powiedzieć, że wprowadzenie tego wyjątku spowoduje, że. Może pan poseł oceniać, że to jest inwestycja prowadzona tak czy inaczej. To jest pana prawo. Każdy ma prawo do swojej oceny, tak. Jeżeli piszemy przepisy, to staramy się pisać przepisy kompleksowo. Państwo tutaj namawiacie do pisania przepisów spójnych, kompleksowych. Stosujemy tych pięć ustaw specjalnych.

Tak samo wie to pani poseł i to jest odpowiedź na pani pytanie. W związku z tym, że w drugim czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Sprzeciwu nie słyszę.

Proszę panią poseł Annę Milczanowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!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 Komisje: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. wnoszą: Wysoki Sejm raczy uchwalić projekt ustawy z druku nr 822 bez poprawek.

Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Arkadiusz Mularczyk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Wysoka Izbo! Odbyła się dyskusja, zostało przedstawione przez właściwych ministrów uzasadnienie proponowanych tutaj zmian. I trzeba podkreślić, że komisje pozytywnie odniosły się do tych proponowanych zmian, zastrzeżeń czy też do wycofania jednego zastrzeżenia. Chcę podkreślić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, że my w całości popieramy proponowane zmiany dwóch zastrzeżeń oraz wycofanie jednego zastrzeżenia. W naszej ocenie te korekty wskazują na postęp w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej, a pozytywnym efektem tych korekt czy tych zmian będzie poszerzenie świadomości w zakresie środków ochrony oraz działań podejmowanych celem wyeliminowania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Zajmijcie się wreszcie na poważnie problemem przemocy domowej w Polsce, żeby ktoś za kilka lat nie wywiesił podobnych plakatów z twarzami właśnie pobitych kobiet i dzieci, z podobnym hasłem: Bo w Polsce rządził PiS. Każdy, kto dzisiaj kwestionuje konwencję antyprzemocową, staje po stronie tych, którzy biją i mordują. Staje po stronie sprawców przemocy domowej. Wysoka Izbo! Obecna władza właśnie zdobywa szczyty Himalajów hipokryzji. Z jednej strony rząd modyfikuje w tej ustawie zastrzeżenia, które Polska złożyła do konwencji antyprzemocowej kilka lat temu, ale z drugiej strony robi bardzo konkretne kroki w celu wypowiedzenia całej konwencji. Najpierw minister sprawiedliwości składa konkretny wniosek, potem premier odsyła konwencję do tzw. Trybunału Konstytucyjnego.

To się dzieje w sytuacji, kiedy prawie 700 tys. Polek każdego roku doświadcza różnych form przemocy domowej. Wysoka Izbo, ale czego można się spodziewać po obecnej władzy? Ta walka z konwencją antyprzemocową prowadzona przez obecną władzę właściwie nie powinna dziwić. Widzimy od kilku tygodni, jak traktowane są Polki. Obecna władza nienawidzi kobiet. To w państwie PiS zmusza się kobiety do rodzenia śmiertelnie chorych dzieci. To w państwie PiS kobiety są napadane w trakcie pokojowych protestów przez zamaskowanych sprawców z pałkami teleskopowymi. To w państwie PiS kobiety atakowane są bez powodu gazem. To w państwie PiS 19-letniej kobiecie służby łamią rękę, a politycy obecnej władzy nie widzą w tym nic zdrożnego, nic złego. Wysoka Izbo! Apeluję dziś do polityków obozu władzy: skończcie wreszcie z prześladowaniem kobiet, powstrzymajcie tę falę brutalnej przemocy, której doświadczają pokojowo protestujące kobiety na ulicach polskich miast, i powstrzymajcie wreszcie tych polityków prawicy, z Ziobrą na czele, którzy otwarcie domagają się i dążą do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. Apeluję dziś do tego rządu: przestańcie wreszcie podważać miejsce Polski wśród cywilizacji Zachodu, podważać zachodnioeuropejskie standardy ochrony praw obywateli. Wycofajcie wniosek z tzw. Trybunału Konstytucyjnego dotyczący konwencji i powstrzymajcie niszczenie praw kobiet w Polsce. Już zniszczyliście miejsce i szacunek do naszego kraju w Unii Europejskiej.

Bardzo proszę, pani poseł Katarzyna Ueberhan, klub Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Obniżcie VAT na wieszaki. Protesty się odbywają, bo nie organizuje ich Sasin. Mefedron ma lepszy skład niż rząd. Nie, to nie są hasła polityczne ani hasła reklamowe, to cytaty z transparentów. Tak, również państwa wyborców manifestujących na ulicach polskich miast, co myślą o rządach prawicy i piekle kobiet, które na polityczne zamówienie z Nowogrodzkiej zafundował nam trybunał niekonstytucyjny. Nie tylko feministkom, nie tylko nam, lewaczkom, ale nam wszystkim, obywatelkom, w tym również tym, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. Zbliża się koniec roku kalendarzowego. To dobry moment na podsumowania, po roku od wyborów parlamentarnych, a w pierwszym roku nowej kadencji. Cóż, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zmienić definicję przemocy, ale nie uzupełniając ją o inne formy - jak choćby ta ekonomiczna, co byłoby zgodne z konwencją - lecz poprzez wykreślenie z definicji wyrażenia: „jednorazowe” Niedoszły projekt przemoc+ na wzór kremlowski zakładał pierwsze pobicie w rodzinie za jeszcze nie przemoc. Ministra rodziny pytana o wypowiedzenie konwencji stwierdziła, że Polska nie może pozwolić na narzucanie sobie jakichkolwiek treści ideologicznych niezgodnych z konstytucją. Cóż, pani minister, akurat równość kobiet i mężczyzn wprost z tej konstytucji, z naszej konstytucji wynika. Wiceminister sprawiedliwości domagał się wcześniej wypowiedzenia genderowego bełkotu, dziś na posiedzeniu komisji poinformował o niezmienionym stanowisku Solidarnej Polski, która chciałaby wypowiedzenia konwencji, tylko że uniemożliwia jej to prawo.

I tak mija nam rok 2020, w którym rządząca prawica, w imię źle rozumianej tradycji, ze strachu przed diablicą gender, rozjeżdża walcem prawa kobiet. Władza dopuszcza się przemocy, najpierw tej instytucjonalnej, ograniczając nam, kobietom, prawa, a w reakcji na falę słusznego sprzeciwu w imię prawa staje się oprawcą. Na polecenie ministra ds. własnego bezpieczeństwa w ruch idzie gaz, policyjne pałki, a protestującym łamie się nie tylko prawa, ale i kości. Będą konsekwencje, ukaranie winnych, usłyszymy: „przepraszam” czy jak od klasycznego przemocowca usłyszymy, że to nasza, kobiet wina, same się prosiłyśmy? Bije funkcjonariusz? Może to nie jest przemoc. Tak wygląda przestrzeganie prawa i wymierzanie sprawiedliwości w państwie Prawa i Sprawiedliwości końca 2020 r. Państwo z prawej strony izby, za wszystko, [[Dzwonek]] co nawarzyliście w tym roku, przyjdzie wam zapłacić polityczną cenę w przyszłości.

Bardzo proszę, pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów i Konserwatyści mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule w dniu 11 maja 2011 r. Rządowy projekt dotyczy zmiany, wycofania i modyfikacji zastrzeżeń złożonych przez Polskę do konwencji stambulskiej. Procedowany projekt ustawy jest potrzebny, wynika bowiem ze zmiany prawa polskiego. Konwencja Rady Europy z 2011 r. ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Wiemy, jak wiele kontrowersji i ideologicznych dyskusji wzbudza. Jako Koalicja Polska apelujemy i uważamy, że żadne skrajności nie powinny tu mieć miejsca. Przemoc wobec kobiet nie jest ideologiczna, nie ma barw politycznych. Niezależnie od narodowości, wyznania, statusu materialnego i społecznego kobiety w naszym kraju powinny czuć się bezpiecznie, a zwłaszcza dzisiaj, w dobie pandemii, kiedy kryzys ekonomiczny i stres nasilają agresję. Do mnie, jako do posłanki, zgłaszają się kobiety z różnymi problemami, często niestety też te, które doświadczają przemocy domowej lub przemocy w środowisku pracy. Mam apel i pytanie do rządu: Czy należycie monitoruje i zapobiega on przemocy, czy wykorzystuje narzędzia, jakie posiada, czy nie należy wzmocnić kontroli państwa w tym zakresie? Jak funkcjonuje „Niebieska Karta” Jak są dzielone środki z Funduszu Sprawiedliwości? Czy faktycznie ten fundusz pomaga osobom pokrzywdzonym i doświadczonym przestępstwem, czy środki z funduszu nadal będą przeznaczane przez pana ministra na inne cele, często niezwiązane z przeciwdziałaniem przemocy? Czy jest wystarczająca współpraca rządu z samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie? Jakie rząd podjął działania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 6 konwencji? Drodzy Państwo! Każda forma zapobiegania przemocy wobec kobiet będzie popierana przez klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego rekomenduję Wysokiej Izbie (Dzwonek) tę ustawę. Dziękuję.

Wysoka Izbo!

Czy tylko retorycznie możecie się przerzucać w ramach swoich walk wewnętrznych, ale jak przychodzi co do czego, to już nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek zrobić? Konwencja stambulska powinna zostać wypowiedziana i to nie dlatego, że ma w sobie komponent antyprzemocowy, bo wszyscy z nas się zgadzają, że ktokolwiek bije dzieci czy kobiety, zasługuje na potępienie, zasługuje na karę, i to w polskim prawodawstwie powinno być implikowane, jak najbardziej. Chodzi o to, że konwencja stambulska została oparta przede wszystkim na ideologicznych założeniach.

Po drugie, zakłada, że konstrukty te zostały nam narzucone na przestrzeni dziejów w wyniku dialektycznej walki płci, nierównych stosunków władzy. W związku z powyższym konwencja stambulska błędnie pojmuje przemoc: nie jako wynik patologii życia społecznego - no tak, przemoc to jest patologia życia społecznego, która powinna być karana - ale jako zjawisko strukturalne, gdzie mężczyźni z góry są ustawiani w pozycji tych złych, którzy zawsze biją. To jest ingerencja w rodzinę, to jest ingerencja w to, jak pojmujemy rodzinę. Celem konwencji jest zatem daleko idąca inżynieria społeczna, sięgająca podstawowych struktur społecznych. Świadczą o tym zarówno sam tekst konwencji, jak i działalność organu powołanego do jej monitorowania. Nie jest możliwe stosowanie konwencji stambulskiej z pominięciem ideologicznych założeń. Dlatego my jako Konfederacja przygotowaliśmy dzisiaj projekt uchwały, w którym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do wszczęcia formalnej procedury wypowiedzenia konwencji stambulskiej, ponieważ to jest jedyna droga, żeby zapobiec tej ideologicznej, lewicowo-liberalnej projekcji wprowadzenia do polskiego prawodawstwa właśnie przesunięcia. przesunięcia naszego prawodawstwa i uznania tego wszystkiego.

Państwo naprawdę nie potrafią tego robić. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu. Panie pośle, proszę zająć swoje miejsce i nie przeszkadzać. Szanowny Panie Marszałku! Pani poseł, momencik. Przepraszam bardzo, czy można. Czy jest szansa, aby umożliwić pani poseł zabranie głosu? Dziękuję. Wysoka Izbo! Ze sprawami kobiet w Polsce jest jak z wyborami premiera Sasina: niby są przepisy, a tak naprawdę nikt nikogo nie ściga.

Nowych zastrzeżeń złożyć nie możemy, ale możemy żonglować istniejącymi. I tak rząd PiS żongluje właśnie teraz prawami kobiet. W tym projekcie tak naprawdę chodzi jednak o utrzymanie w mocy jednego z zastrzeżeń o fundamentalnym znaczeniu. Wytłumaczę treść tego prostymi słowami. Rząd miga się od ścigania z urzędu tzw. naruszenia nietykalności cielesnej, czyli np. pobicia, szarpania, popychania, uderzania, spoliczkowania, targania za włosy, przygniatania kolanem do podłogi, aktów codziennej przemocy, które w Polsce musi znosić, zgłosić ofiara mieszkająca pod jednym dachem z oprawcą. I często potem to zgłoszenie wycofuje pod wpływem gróźb. Tymczasem właśnie naruszenie nietykalności to jedna z najczęstszych kwalifikacji czynów wobec kobiet padających ofiarami przemocy. Tym samym rząd przyznaje, że od 5 lat nie zrobił nic, by to państwo, nie ofiara, ścigało domowych oprawców, sadystów. A tego wymaga od nas konwencja. Naruszenie nietykalności i ściganie na mocy art. 217 Kodeksu karnego z oskarżenia prywatnego nazywa się w Polsce drobnym przestępstwem. Samo w sobie jest to już skandalem. Dziś na posiedzenie komisji sprawiedliwości zaniosłam poprawkę, która kończy to piekło, i od pana ministra Romanowskiego dowiedziałam się, że ściganie przemocy domowej z urzędu to za dużo roboty dla polskiej Policji. Dobrze państwo usłyszeliście. Witajcie w kraju, w którym z oskarżenia publicznego ściga się obrazę uczuć religijnych, ale nie damskich bokserów, w kraju, gdzie 600 policjantów strzeże domu jednego prezesa, a brakuje ich do ratowania katowanych kobiet, gdzie minister sprawiedliwości otwarcie przyznaje, że skala przemocy domowej przekracza możliwości służb i państwa. To hańba, że ofiary przemocy domowej ciągle mogą liczyć w Polsce tylko na siebie. Dlatego proszę Wysoką Izbę o poparcie wniosku mniejszości, dzięki któremu to państwo, a nie ofiary, będzie zobowiązane do zakończenia domowego piekła kobiet.

Na tym lista osób przedstawiających stanowiska klubów parlamentarnych i koła została wyczerpana. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj o fundamentalnych prawach człowieka, o czymś, co możemy nazwać - aż to dziwnie brzmi - cywilizacyjnym osiągnięciem, czymś, co jest oczywiste, a jednak cały czas musimy o to walczyć.

Chciałbym to usłyszeć z tej mównicy sejmowej od przedstawiciela rządu. To po pierwsze. Po drugie, Polska ma jednak bardzo poważny problem systemowy z walką z przemocą w rodzinie.

Chciałbym, żeby przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej [[Dzwonek]] odciął się od haniebnych słów, które padły z ust przedstawiciela tego rządu pani Beaty Szydło, która chwaliła Zakopane za to, że nie przyjęło lokalnego programu zwalczania przemocy domowej. Pytanie zada pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Konwencja stambulska jest niezwykle ważnym aktem prawnym dającym kobietom ofiarom przemocy domowej możliwość natychmiastowej izolacji od sprawcy. Bite kobiety, maltretowane dzieci nie muszą czekać miesiącami, a czasami latami na wyrok sądu, aby policja mogła odseparować sprawcę. Niezwykle martwi jednak fakt, że tak ważny akt prawny jest kwestionowany przez polityka, który powinien stać na straży każdego prawa wspierającego ofiary przemocy i być przeciwko sprawcom. Minister sprawiedliwości powinien stać po stronie ofiar. Niestety zostało wszczęte postępowanie w sprawie wypowiedzenia konwencji, a także została skierowana sprawa do Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni państwo, jeśli chce się bronić kobiet, ofiar przemocy domowej, [[Dzwonek]] to jest się za konwencją. Jeśli jest się przeciw konwencji, to gdzie się jest, pytam. Dziękuję bardzo. Proszę teraz panią poseł Małgorzatę Tracz o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zastrzeżeniu tym Polska uznaje, że obowiązek wszczynania postępowania z urzędu nie dotyczy drobnych przestępstw. Takimi drobnymi przestępstwami są według Kodeksu karnego występki naruszenia nietykalności cielesnej, które są w Polsce ścigane z oskarżenia prywatnego. Naruszenie nietykalności cielesnej to nic innego jak uderzenie, spoliczkowanie, kopnięcie, szarpanie, popychanie, przytrzymywanie czy ciągnięcie za włosy. To jest nic innego niż podstawowy katalog przemocy fizycznej w ramach przemocy domowej. Konwencja stambulska zobowiązuje nas do ścigania takich przestępstw z urzędu, natomiast nie działa to w Polsce, bo Polska nie zmieniła tej sytuacji przez ostatnich 5 lat, zasłaniając się omawianym zastrzeżeniem. Stąd moje pytanie do ministra sprawiedliwości.

Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę teraz panią poseł Katarzynę Lubnauer o zadanie pytania. Panie i Panowie Posłowie! Panie Marszałku! Właściwie chciałabym się zwrócić do posłów PiS, ale jak widać, temat ich nie interesuje, dlaczego są takimi tchórzami. Tchórzliwie zabrali poprzez Trybunał Konstytucyjny podstawowe prawo kobiety do aborcji w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu, a w tej chwili po raz kolejny przy pomocy tego samego Trybunału Konstytucyjnego chcą wypowiedzieć konwencję stambulską, mimo że Trybunał Konstytucyjny nie ma uprawnień do badania tego, czy ta konwencja i jej tłumaczenie są ze sobą zgodne.

A tak naprawdę to każdy cywilizowany kraj powinien wprowadzić jej zapisy.

Dziękuję bardzo. Proszę teraz panią poseł Katarzynę Marię Piekarską o zadanie pytania. 16 lipca pani minister Maląg: przygotowujemy się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Pan Marcin Horała: jeśli analiza różnych aspektów prawnych wykaże, że można konwencję stambulską wypowiedzieć, to tak się stanie. Dlatego pytam: Czy ofiary przemocy domowej mogą spać spokojnie, czy raz na zawsze powiecie państwo, że nie wypowiecie tej konwencji, i czy nie będzie tak, że przed kolejnymi wyborami, kiedy będziecie rywalizować o głosy z Konfederacją, jednak tę konwencję wypowiecie? Czy organizacje pozarządowe, które od lat pomagają ofiarom przemocy domowej, mogą liczyć na wsparcie finansowe na swoją działalność ze strony rządu, np. z Funduszu Sprawiedliwości?

Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Mirosława Suchonia o zadanie pytania. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Myślę, że podstawowe pytanie, które musimy sobie dzisiaj zadać i na które każdy powinien sobie odpowiedzieć. Przepraszam, panie pośle. Czy panowie posłowie mogą przenieść dyskusję poza salę? Bardzo dziękuję, panie marszałku. Czy rząd powinien dbać o bezpieczeństwo ofiar przemocy, czy powinien pomagać tym ofiarom, zapewnić im bezpieczeństwo, czy też powinien dbać o dobre samopoczucie sprawców tych przestępstw? Wydaje się, że racjonalnym, zdroworozsądkowym i realnym w całym cywilizowanym świecie postępowaniem jest dbanie o ofiary przemocy i jak najbardziej krytyczne podejście do tych, którzy stosują przemoc.

I to przedstawicielka ministra sprawiedliwości broniła tego stanu rzeczy.

I drugie pytanie: Czy zostawi konwencję w spokoju? Ona gwarantuje właśnie to, że państwo jest zobowiązane do dbania o ofiary przestępstw, a nie o dobre samopoczucie sprawców. Dziękuję.

Wysoka Izbo! Rozmawiamy o konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale symboliczne jest również to, że dzisiaj z tej mównicy wiceminister Maciej Wąsik powiedział w sprawie złamania ręki 19-letniej Aleksandry, że na tym etapie nie ma powodów do tego, żeby uważać, że policjanci bezprawnie użyli środków przymusu.

Jest to symboliczne. Druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy realnie walczyć z przemocą wobec kobiet, z przemocą domową, to potrzebne są również środki. Przez lata takie organizacje pozarządowe jak Centrum Praw Kobiet otrzymywały środki z Funduszu Sprawiedliwości. Cały Fundusz Sprawiedliwości został w tej chwili przekierowany na autopromocję polityków Solidarnej Polski. Pamiętacie państwo, jak Andrzej Duda ułaskawił ojca pedofila. Wtedy było pytanie, jak tej rodzinie, jak tej matce, jak tej córce pomagało państwo polskie.

Pan poseł Aleksander Miszalski zada teraz pytanie. Wysoka Izbo!

Czy wy wiecie, z czego wynika ta różnica? W Szwecji każdy przypadek fizycznej przemocy wobec kobiet jest ścigany z urzędu, co automatycznie zwiększa wykrywalność przestępstw. Panie Pośle Mularczyk! Niech pan spróbuje sobie wyobrazić, że jest pan kobietą, mieszka w małej miejscowości, nie pracuje, prowadzi dom i jest pan finansowo zależny od swojego partnera. Myśli pan, że taka kobieta, czyli pan, wtedy zgłosiłaby się do policji? Rozumiem, że ostatnio nie jest wam za bardzo po drodze z kobietami. Powiedzcie, dlaczego nie chcecie wykonać w stronę kobiet tego drobnego gestu.

Czy mógłbym prosić o odpowiedź na piśmie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zadanie pytania panią poseł Monikę Rosę, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Kobiety w Polsce umierają w zaciszu swoich domów. 500 kobiet rocznie umiera w wyniku kobietobójstwa albo samobójstw powodowanych przemocą domową. Ile dokładnie, nie wiemy, ponieważ rząd nie prowadzi danych, statystyk w tej sprawie. Potrzebujemy bardzo mocno zmiany funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, nowelizacji tej ustawy, zmiany funkcjonowania „Niebieskiej karty” Szanowni państwo, państwo ministrowie, kiedy to się stanie? Potrzebujemy wpisania definicji przemocy ekonomicznej do polskiego prawa. Kiedy to się stanie? Potrzebujemy zmiany definicji gwałtu w polskim prawie. Kiedy to się stanie? Potrzebujemy nowego krajowego programu przeciwdziałania przemocy domowej - wieloletniego. Państwo planujecie ten program tylko na najbliższy rok. W ciągu roku nie uda się skutecznie przeprowadzić takiego programu. Dlaczego tylko na rok? Wciąż czekamy na to, aż wszystkie gminy w Polsce będą miały gminne programy przeciwdziałania przemocy domowej. Kiedy to się stanie? Państwa obowiązkiem jest nadzorować, [[Dzwonek]] żeby gminy miały takie programy. Wciąż czekamy na informację, kiedy zespół monitorowania przemocy zostanie powołany. Miał być z końcem października. Wciąż takiego zespołu nie ma. Pytanie zada pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister, która łączyła się z nami z rządowej limuzyny! Fakty są takie, że 25 lipca minister Ziobro złożył oficjalny wniosek o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej - konwencji, która zawiera szereg mechanizmów, które pozwalają skuteczniej niż polskie prawo chronić kobiety, m.in. rozszerzają definicję przemocy domowej czy klasyfikują przemoc ekonomiczną. A co robi rząd? Kładzie na szali bezpieczeństwo kobiet, i to w tak krytycznym momencie, jakim jest pandemia, kiedy większość z nas przebywa w izolacji. Tylko jedna z organizacji, Centrum Praw Kobiet, której zresztą odebraliście środki na funkcjonowanie, odnotowała blisko 50% więcej połączeń telefonicznych na numer interwencyjny i ok. 20% więcej zgłoszeń mailowych. Kobiety zamknięte z oprawcami w domach potrzebują realnej pomocy, realnych narzędzi prawnych, a takie właśnie zapewnia im ta konwencja. Perfidnie igracie bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem milionów kobiet w Polsce. Sprzedajecie bajki o ideologicznym wymiarze tej konwencji. Dziś dyskutujemy nad kwestiami wykonawczymi. Pozwala to więc mieć nadzieję, że te nieludzkie pomysły pana Ziobry wylądowały na śmietniku. Czy możecie w końcu dać nam gwarancję, że nie podniesiecie ręki na konwencję antyprzemocową i polskie kobiety? Miliony kobiet oczekują na tę odpowiedź. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Michała Krawczyka, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 13 maja br. wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski napisał o konwencji antyprzemocowej, cytuję: chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot. W odpowiedzi na moją interpelację, którą natychmiast skierowałem, pan minister podtrzymał to, że Solidarna Polska jest za wypowiedzeniem konwencji. 16 lipca na antenie jednej z rozgłośni radiowych minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg stwierdziła, że Polska szykuje się do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. Wówczas znów skierowałem interpelację, domagając się wyjaśnień. Pani minister napisała, cytuję: Rada Ministrów nie podjęła decyzji o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej przez Polskę, zostawiając oczywiście w ten sposób furtkę do podjęcia takiej decyzji w przyszłości i nie określając jednoznacznie stanowiska polskiego rządu. W związku z tym pytam panią minister: Czy są prowadzone jakiekolwiek działania, które mają doprowadzić do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej przez Polskę? Proszę wyjść i odważnie to powiedzieć tutaj, z tej mównicy, i zakończyć tę schizofrenię polskiego rządu. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Franciszka Sterczewskiego, Koalicja Obywatelska, do zadania pytania. Wysoka Izbo! Nie mogę uwierzyć, że w dniu, w którym z powodu epidemii zmarło ponad 600 osób, rząd znajduje czas, żeby po raz kolejny wdawać się w spory z kobietami. Konwencja stambulska nie pasuje wam od początku. To przedstawiciele waszego rządu mówili o konwencji rzeczy haniebne. Ale to nieprawda. Konwencja dotyczy zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zapamiętajcie to sobie raz na zawsze. Prawa kobiet, prawa antyprzemocowe to nie ideologia, lecz fundamentalne prawa człowieka. W wyniku przemocy domowej co roku ginie w Polsce ok. 500 kobiet, ok. 700 tys. jest bitych i prześladowanych. Dlaczego zatem polski rząd nie realizuje postanowień konwencji stambulskiej? Dlaczego stajecie po stronie oprawców? Czy możecie z tej mównicy zadeklarować, że [[Dzwonek]] polski rząd wbrew deklaracjom ministra Ziobry nie wycofa się z konwencji stambulskiej? Oczekuję jasnej i konkretnej odpowiedzi. Przestańcie być tchórzami. Dziękuję bardzo. Pytanie teraz zada pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Rzeczywiście 17 lipca pani minister Maląg zadeklarowała, że rząd szykuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, i później wielokrotnie to oświadczenie dementowano. I teraz właśnie pytanie: Czy to znaczy, że rząd nigdy się nie szykował do wypowiedzenia tej konwencji i pani Maląg kłamała - a jeśli kłamała, to jaka odpowiedzialność polityczna i karna ją z tego tytułu spotkała, bo składanie fałszywych oświadczeń w imieniu rządu publicznie jest chyba czymś skrajnie nieodpowiedzialnym - czy też rząd szykował się, ale się przestał szykować i w takim razie czemu znowu narobił w zbroję i zrezygnował z tego, co obiecywał? To jest tylko świstek papieru. Nikt nie został skazany ani tym bardziej nie powstrzymał się od przemocy z powodu konwencji stambulskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie mów nikomu, co się dzieje w domu - oraz: zły to ptak, co swe gniazdo kala. To według mnie dwa najgorsze przysłowia w języku polskim. Niestety często to właśnie w rodzinach dzieje się najwięcej przemocy, a te przysłowia namawiają do tego, żeby to zło ukrywać i by ofiary cierpiały w milczeniu. Często przemoc w rodzinie jest nieudokumentowana. Przecież tam nie ma kamer ani dziennikarzy, ale jest autentyczne cierpienie ofiar. Dlatego cieszę się, że Polska - przynajmniej jak dotąd - nie wypowiedziała konwencji stambulskiej, której podpisanie gwarantuje także, by kultura czy religia nie były usprawiedliwieniem dla przemocy w rodzinie. Niestety ten rząd, nie zważając na ten fragment, dodał nowe powiedzenia: co się dzieje na plebanii, nie rozpowiadaj ani ani albo: jesteś pedofilem w sutannie, sprawiedliwość cię nie dopadnie. A może najwyższa pora na zupełnie nowe przysłowie: wzajemny szacunek i rozmowa to polska tradycja domowa? Dziękuję. Proszę pana posła Artura Łąckiego, Koalicja Obywatelska, o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! A ja się cieszę, że PiS grzebie w konwencji stambulskiej. Róbcie tak dalej. W październiku wasz prezes kazał pani Przyłębskiej rozwalić kompromis, który może nie był dobry, ale funkcjonował. Teraz, grzebiąc w tym, ponownie wyciągnięcie kobiety na ulice i mam nadzieję, że to kobiety posprzątają po was w polityce i was posprzątają. Co wy w ogóle macie do kobiet? Czy wy jako dzieci, nie wiem, byliście bici przez matki? Albo was zamykały w ciemnym pokoju ze strasznymi lalkami, takimi szmacianymi i do tej pory nie potraficie się z tego otrząsnąć?

Proszę panią poseł Magdalenę Biejat, Lewica, o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trzymajmy się faktów. Według oficjalnych danych, danych Policji 75% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety. Według tych samych danych 90% sprawców przemocy to mężczyźni. Przemoc ma płeć. Płeć ma znaczenie, kiedy mówimy o przemocy w rodzinie. Nic więc dziwnego, że każda zapowiedź o możliwym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej, każda zapowiedź składania zastrzeżeń do konwencji antyprzemocowej wywołuje popłoch i przerażenie wśród kobiet, właśnie kobiet. Kiedy minister Maląg zapowiedziała wypowiedzenie konwencji i składanie zastrzeżeń, wraz z grupa posłów i posłanek Lewicy złożyłam interpelację w tej sprawie. Pani minister Maląg przez 3 miesiące nie odpowiadała. Kiedy wreszcie odpowiedziała, użyła oczywiście bardzo ogólnych określeń, ale jedno szczególnie chciałabym zacytować: W razie stwierdzenia niezgodności postanowień konwencji z Konstytucją RP wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie miał skutek derogacyjny.

Czy znowu chcecie tylnymi drzwiami, umywając ręce, wprowadzić kolejne ograniczenia praw kobiet? Domagam się jasnej deklaracji, jaki jest stosunek rządu do konwencji przemocowej. Proszę panią poseł Małgorzatę Prokop-Paczkowską, klub parlamentarny Lewicy, o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy kilka lat temu walczyliśmy, my, kobiety i mężczyźni, o ratyfikację konwencji, Platforma bardzo długo tej ratyfikacji nie podejmowała, podarowałam prezydentowi Komorowskiemu koszulkę z wielkim napisem: Tak dla konwencji. Prezydent ją obejrzał i odpowiedział mi: Ale dlaczego pani mi to daje? Obojętność i niezrozumienie tematu - to było wtedy. Dziś jest jeszcze gorzej, bo dziś rządzi nami skrajna prawica. Ktoś z Konfederacji przed chwilą powiedział, że przemoc bierze się z patologii. Mam więc pytanie: Czy obwinianie kobiet za to, że zostały zgwałcone, bo miały krótką spódniczkę, bo piły alkohol, bo za słabo się broniły albo że za cicho krzyczały, bo taki wyrok niedawno (Dzwonek) zapadł, tak uzasadniony, to patologia? Tak, to patologia. Bo koalicja rządząca jest przemocowa i patologiczna. Mam pytanie do ministra Czarnka: W jaki sposób w nowych podręcznikach, które już szykuje, z nową podstawą programową, będzie walczył z przemocą wobec kobiet?

Proszę teraz panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę o zadanie pytania.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Czas lockdownu jest szczególnie trudny dla ofiar przemocy domowej. Zamyka się nas w domach i wszystkie frustracje i problemy za tymi zamkniętymi drzwiami po prostu narastają. Szacuje się, że wzrost interwencji z tytułu przemocy domowej sięga nawet 90%.

Na taką deklarację czekają polskie kobiety. Dziękuję. Pytanie zada pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Liczba aktów przemocy domowa rośnie, a w ostatnim czasie - zwłaszcza w tym roku - jest to wzrost lawinowy. Rząd nie dostrzega problemu, a nawet go lekceważy. Hierarchowie kościelni ironizują na ten temat. Tymczasem w okresie pandemii, kiedy rodziny są zamknięte w domach razem z oprawcami, dzieją się straszne sceny. Chciałam zapytać: Jakie środki finansowe zabezpieczył rząd w budżecie państwa na rosnące gwałtownie potrzeby w zakresie pomocy ofiarom przemocy?

Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania panią poseł Bożenę Żelazowską, Koalicja Polska. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ideologizowanie przemocy nie ma sensu. Każda przemoc wobec każdej osoby jest po prostu bandytyzmem. Jednak to rząd posiada narzędzia, które mogą przeciwdziałać przemocy. Wiele z pytań, które chciałabym teraz zadać, zawarłam w moim wcześniejszym wystąpieniu, ale mam pytanie do pani minister: W jakim zakresie - czy w wystarczającym - rząd współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi, aby przeciwdziałać przemocy?

Dziękuję bardzo. Czy na sali jest pani poseł Gabriela Lenartowicz? Bardzo proszę o zadanie pytania.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Tymczasem Fundusz Sprawiedliwości, który ma pomagać osobom pokrzywdzonym w przestępstwach oraz osobom najbliższym, wydaje pieniądze np. na projekty Fundacji Czyste Serce, które mają wspierać jak największą liczbę kobiet i mężczyzn, aby osiągnęli szczęście w miłości, i podejmuje działania, aby każde małżeństwo było sakramentalne, a jak największa liczba dziewcząt i chłopców rozpoczęła życie seksualne po ślubie. Padło tu dzisiaj stwierdzenie, że przemoc bierze się z patologii.

Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zadanie pytania panią poseł Katarzynę Ueberhan, Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z raportu rzecznika praw obywatelskich wynika, że wiele jednostek samorządu terytorialnego w Polsce nie przeprowadziło lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie. Co z powiatami, gminami, które nie przyjęły programu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, pomimo że mają ustawowy obowiązek? Czy i jak organy administracji państwowej sprawują wynikający z ustawy nadzór nad gminami w tym zakresie? Jak rozdzielane są publiczne środki, w tym te z tzw. Funduszu Sprawiedliwości? Czy polskie prawo zacznie rozpoznawać inne formy przemocy niż ta fizyczna? Co z definicją gwałtu? Co z „Krajowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Obecny program właśnie się kończy, a projekt jego kontynuacji na kolejne lata nie został jeszcze przedstawiony. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie zada teraz pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Dyskusja z wami na ten temat nie ma najmniejszego sensu, bo wasze słowa nie mają żadnego znaczenia. W grudniu 2016 r. minister pracy Elżbieta Rafalska powiedziała: jestem za wypowiedzeniem przez Polskę konwencji stambulskiej. Resort sprawiedliwości potwierdził, że rozpoczyna w tej kwestii prace. Co jakiś czas zapowiadaliście wypowiedzenie.

Mam więc pełne nadziei pytanie: Czy możemy liczyć na taką samą wieloletnią opieszałość w realizacji waszych zapowiedzi dotyczących podwyżek podatków? W trybie sprostowania głos zabierze teraz pani poseł Katarzyna Lubnauer. Pan poseł Sośnierz powiedział, że to nie jest tak, że kobiety żyją kwestią konwencji stambulskiej. Przytoczmy liczby.

I dlatego również takie zdania jak pana i jak pan kolegi są nieodpowiedzialne. Konwencja stambulska jest jednym z dokumentów, który pomaga rządowi podejmować słuszne decyzje.

Na tym lista posłów zapisanych do pytań została wyczerpana. Proszę teraz panią Annę Schmidt, która jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej o zabranie głosu.

Jakby pan za chwilę użył nazwiska pani poseł, to znowu ona by się chciała odnieść i byśmy tak mogli siedzieć do rana. Proszę panią minister o zabranie głosu, a pana posła proszę uprzejmie o zejście z mównicy i zajęcie miejsca tam, gdzie powinni zasiadać posłowie. A ja panu jeszcze raz mówię, że pana bardzo grzecznie proszę o zejście z mównicy, bo już raz pan dał popis zdziczenia obyczajów, wpadając w ławy opozycji i wymachując rękami do kobiet. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo na mównicę, pani minister. Co to jest za bezczelne odzywanie się? Co to jest za demagogia? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W tej części, która dotyczy resortu rodziny oraz mojego wystąpienia na porannym posiedzeniu. Panie pośle, proszę usiąść na swoje miejsce i nie prowokować posłów opozycji.

Postaram się odpowiedzieć na większość pytań, które tutaj dzisiaj padły, nawiązując też do mojego wystąpienia na porannym posiedzeniu połączonych komisji. Po pierwsze, chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałam rano i co już wielokrotnie padało. Powtórzę to jeszcze raz: ani Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ani rząd wedle mojej wiedzy, mam nadzieję, że gruntownej, nie prowadzi żadnych działań ani żadnego postępowania, które zmierza do wypowiedzenia konwencji. Jak państwo doskonale. Pani poseł, proszę mi pozwolić skończyć.

W związku z tym premier uznał, że taki wniosek należy tam skierować. Czekamy, aż zostanie uruchomiona procedura w Trybunale Konstytucyjnym i ten wniosek zostanie poddany analizie. To wszystko, co mam do powiedzenia, po raz kolejny zresztą, szanowni państwo posłowie, jeśli chodzi o zakres prac związanych z konwencją stambulską. Jeśli chodzi o pytanie pana posła Szłapki dotyczące wykrywalności przestępstw, to ja jestem przekonana, że tutaj pan minister Romanowski będzie chciał zabrać głos.

Z danych, które zresztą były prezentowane, jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonywania ustawy o zapobieganiu przemocy - tydzień temu toczyła się na ten temat debata w Senacie - wynika, że w istocie wzrosła wykrywalność tych przestępstw, tzn. ilość powiadomień w ramach „Niebieskiej Karty” Czego to dowodzi?

Jeśli chodzi o pytanie jednej z pań posłanek - tutaj odniosę się do wypowiedzi pani posłanki, przedstawicielki klubu Lewicy - to, o ile dobrze sobie przypominam, pani poseł uczestniczyła w porannym posiedzeniu połączonych komisji. Jeśli nie, to przedstawicieli Lewicy zachęcam do odtworzenia tego posiedzenia. Zadziwia mnie, szczerze powiedziawszy, i zdumiewa stwierdzenie, że pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, czyli moja skromna osoba, ja - rzekomo, bo tu takie stwierdzenie padło z ust pani poseł - nie wie, co się dzieje w sprawach konwencji stambulskiej. O ile sobie dobrze przypominam, a pamięć mnie chyba jeszcze nie zawodzi, to właśnie ja rano wspólnie z ministrem Wawrzykiem i z ministrem Romanowskim, odpowiadając na pytania parlamentarzystów, którzy wzięli udział w posiedzeniu komisji, odpowiadałam na te pytania i motywowałam, tłumaczyłam, jaka jest zasadność wniosku i zastrzeżeń, które Polska składa w takiej formule, w jakiej one zostały złożone, a więc, jak państwo wiecie, dwa zostają nieco zmienione, jedno podtrzymane, a jedno wycofane. Będziecie państwo wiedzieć, jakie jest stanowisko rządu, jaka jest zasadność przedłożenia tych zastrzeżeń i jakie jest również stanowisko w tej sprawie, a raczej wiedza, bo do tego wypowiedź pani poseł się odnosiła, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania.

do procedury „Niebieskie karty”, która jest podawana właśnie przez przedstawicieli GREVIO, i nie tylko, przez Unię Europejską jako wzorcowy przykład rozwiązań, które zresztą zostały wdrożone już, jak państwo wiecie, wiele lat temu. Jeśli chodzi o pytanie - trochę tutaj wejdę w kompetencje ministra Romanowskiego, ale chciałabym się odnieść do tego - dotyczące tego, jakie rząd podejmuje działania, żeby zabezpieczyć szczególnie w okresie COVID-u ofiary przemocy, to przypomnę państwu, że niedawno przeprocedowaliśmy w polskim parlamencie ustawę autorstwa ministra sprawiedliwości, która w sposób natychmiastowy i skuteczny nie procedurami sądowymi, o jakich mówi konwencja stambulska, tylko procedurą szybkiej reakcji służb, w tym przypadku służb Policji, wprowadziła zapisy dotyczące natychmiastowej izolacji i wykluczenia z gospodarstwa domowego, z mieszkania, w którym przebywa ofiara, sprawcy tej przemocy.

To są kraje, które ratyfikując konwencję, zgłosiły zastrzeżenia do art. 55 wynikające z niczego innego jak właśnie z tego, że taki jest kształt prawa i art. 217 dotyczącego nietykalności cielesnej.

to pozwoli pani, że przekażę teraz głos oczekującemu na swoją wypowiedź panu ministrowi Romanowskiemu. Stwierdzę pod koniec swojej wypowiedzi tylko tyle, że chciałabym zwrócić uwagę państwa posłów, przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, że w momencie, kiedy konwencja stambulska była ratyfikowana, a więc 24 kwietnia 2015 r., to państwa ekipa rządziła, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to państwa ekipa zgłosiła zastrzeżenia, w tym do art. 55, wynikające z brzmienia art. 217, a ministrem wtedy był pan Cezary Grabarczyk, a po nim pan Borys Budka. A zatem rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy w ślad za tym, jaki jest obecnie obowiązujący kształt art. 217, jedynie to zastrzeżenie podtrzymał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kontynuując wypowiedź pani minister i nawiązując właśnie do art. 217, chciałbym też jeszcze dodatkowo zauważyć, że nie jest prawdą, że to ten przepis służy do kwalifikacji zjawisk związanych z przemocą domową. To jest przepis bardzo ogólny, który dotyczy całego spektrum lekkich przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej, a nie przeciwko życiu i zdrowiu, na co wskazuje umiejscowienie w rozdziale 27, a nie w rozdziale 19.

Wszystkie te wskazane czyny zabronione są ścigane z urzędu.

Jeżeli chodzi o statystyki, bo tutaj były pytania, ale było też wiele fałszywych, jak się wydaje, informacji, to nie obserwujemy - mówię o perspektywie ostatnich lat - jakiegoś istotnego wzrostu tego typu przestępczości, na co wskazują statystyki policyjne.

Chciałem zauważyć, że to przestępstwo miało miejsce w tym czasie, więc proszę skierować to pytanie do kogoś innego.

W naszej ocenie konwencja w wymiarze normatywnym nie wnosi nic do standardu ochrony, bo on już w momencie jej ratyfikacji był równy albo wyższy, jeżeli chodzi o rozwiązania krajowe, a w naszej ocenie, którą wielokrotnie wyrażaliśmy, może nie będę jej szczegółowo powtarzał, w warstwie ideologicznej ona jest niebezpieczna, bo np. błędnie identyfikuje przyczyny przemocy, właśnie wskazując na tradycję, role płciowe, a nie w patologie w postaci alkoholu, narkotyków i uprzedmiotowienia roli kobiety, przez co również ma znaczenie kontrfaktyczne.

To jest dobre porównanie, bo według standardów konwencyjnych ofiara musiała pozostawać ze sprawcą przemocy średnio przez 142 dni, bo tyle wynosił czas wydawania orzeczeń przez sądy.

Jesteśmy tutaj w dobrym towarzystwie, bo to są Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa i Łotwa.

Pierwsze tygodnie działania ustawy o natychmiastowym nakazie policyjnym właśnie to pokazują, że ofiary przemocy mogą rzeczywiście czuć się bezpiecznie, bo nie muszą pozostawać ze sprawcą przemocy przez 140 dni pod jednym dachem albo nie muszą uciekać z domu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.

Bardzo proszę, pani minister, o udzielenie tej odpowiedzi. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Rzeczywiście program został przyjęty nie w perspektywie wieloletniej, tylko na rok. Wynika to z faktu, o czym już mówiłam na porannym posiedzeniu połączonych komisji, że ministerstwo rodziny szykuje zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pojęcie, które funkcjonuje od wielu lat w ustawie, jest pojęciem zawężonym. Polskie prawo do tej pory stanowi o pojęciu przemocy w rodzinie, mamy świadomość i zdajemy sobie sprawę z tego, że przemoc obejmuje wszelkie rodzaje przemocy w tzw. gospodarstwie domowym, również w związkach nieformalnych, związkach partnerskich, a więc nie tylko w tradycyjnym ujęciu rodziny jako związku małżeńskiego.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu (druki nr 831 i 838) Bardzo proszę pana posła Arkadiusza Mularczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dwóch połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych, które dotyczy właśnie projektu ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Spraw Zagranicznych po wysłuchaniu głosów w dyskusji pozytywnie zaopiniowała przedłożoną inicjatywę i wnosi o jej uchwalenie przez Wysoką Izbę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi za przedstawienie sprawozdania. Przystępujemy teraz do prezentacji stanowisk klubów i koła.

Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni Państwo! Przedstawiając stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość na temat rządowego projektu ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu, chciałbym podkreślić, że ten rządowy projekt ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowań karnych w tego rodzaju sprawach i umożliwia przekazanie do Polski obywatela polskiego odbywającego na Tajwanie długoterminową karę pozbawienia wolności. Klub Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie opiniuje rządowy projekt. Dzięki przedmiotowej ustawie, która określa zasady funkcjonowania porozumienia, łatwiejszy będzie kontakt w sprawach karnych między odpowiednimi do tych spraw organami centralnymi Polski oraz Tajwanu. Dziękuję uprzejmie, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Tomasza Lenza o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja

Wysoka Izbo! Procedujemy nad projektem ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu. To właśnie przedstawiciele strony tajwańskiej zwrócili się do polskiego rządu z prośbą o rozmowy dotyczące podpisania tego porozumienia, zwracając uwagę, że Polska jest wykorzystywana szczególnie jako miejsce popełniania oszustw internetowych, a opóźnienia w wykonywaniu wniosków o pomoc prawną załatwianych obecnie na zasadzie wzajemności utrudniają postępowanie w zakresie ścigania przestępców. Dotyczy to właśnie zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni. Polska strona zwraca uwagę, że zakres podmiotowy porozumienia jest stosunkowo szeroki i obejmuje nie tylko kwestię cyberprzestępczości, bo obejmuje wzajemną pomoc prawną, ekstradycję, przekazywanie osób skazanych, udzielanie informacji o prawie i praktyce jego stosowania oraz udzielanie informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom. Porozumienie dotyczy także spraw karnych należących do właściwości sądów i prokuratury. Użyte w polskim tekście pojęcie „dochodzenie” należy wykładać autonomicznie, jako każde postępowanie mające na celu ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo, kto jest jego sprawcą, jaką odpowiedzialność powinien ponosić. Jak widzimy, to porozumienie, które jest bardzo szeroko opisane w ustawie, ono ma ponad 24 strony, obejmuje ważne kwestie dotyczące relacji prawnych w ramach ścigania przestępców. Natomiast zwracam uwagę na fakt, że zacieśniamy relacje polityczne, relacje prawne z Republiką Chińską, bo tak nazywa się w oficjalnych dokumentach Tajwan, który nie jest uznawany przez Chińską Republikę Ludową. Jak państwo wiedzą, Chiny cały czas domagają się powrotu Tajwanu do Chin kontynentalnych, protestując przeciwko relacjom międzynarodowym. Przepraszam bardzo. zapobiegając jakimkolwiek relacjom międzynarodowym, dyplomatycznym Tajwanu z jakimikolwiek krajami, więc na pewno strona chińska bacznie przygląda się zacieśnianiu tych relacji na kolejnych płaszczyznach.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi i przepraszam jednocześnie. To wyłączenie przypadkowe, nie miało charakteru recenzowania pana opinii w tej kwestii. Proszę bardzo pana posła Andrzeja Szejnę, który przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo! Procedowany projekt ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu, ma przede wszystkim transponować instrument o współpracy w sprawach karnych do polskiego porządku prawnego. Jest to więc ustawa, która umożliwia stosowanie uzgodnień porozumienia zawartego między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanego dnia 17 czerwca 2019 r. Art. 1 ustawy transponującej wskazuje bowiem, że współpraca z Tajwanem prowadzona jest na podstawie porozumienia, a więc w trybie i na zasadach w nim określonych, w tym określających chwilę jego wejścia w życie. Odnosząc się zatem do procedowanej ustawy, należy mieć na względzie właśnie to porozumienie, które określa zasady m.in. wzajemnej pomocy prawnej, ekstradycji, udzielania informacji o prawie i praktyce jego stosowania oraz udzielania informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosowane będą przepisy właściwego prawa krajowego, w przypadku Polski oczywiście będzie to Kodeks postępowania karnego. Strona tajwańska, która była inicjatorem podpisania porozumienia, wskazywała, że terytorium Polski jest miejscem niestety wykorzystywanym do oszustw internetowych. Długi czas rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy prawnej utrudnia postępowanie karne, szczególnie w zakresie cyberprzestępczości, kiedy szybki czas reakcji organów ścigania może doprowadzić do zatrzymania sprawców, natomiast zwłoka najprawdopodobniej będzie skutkować uniemożliwieniem wymierzenia sprawiedliwości.

Stosowanie postanowień porozumienia przyspieszyłoby i uprościło prowadzenie postępowań karnych w tego rodzaju sprawach wszczętych zarówno przez polskie, jak i przez tajwańskie organy ścigania. Ponadto na mocy art. 5 określającego zasady przekazywania osób skazanych umożliwiłoby sprowadzenie obywatela Polski, o czym była już mowa, odbywającego obecnie karę pozbawienia wolności w tajwańskim zakładzie karnym.

Wysoka Izbo! W wymiarze międzynarodowym przyjęcie ustawy transponującej umożliwi intensyfikację kontaktów polsko-tajwańskich. Klub parlamentarny Lewica popiera procedowany projekt ustawy ze względu na zdecydowane uproszczenie i przyspieszenie postępowania karnego w sprawach między RP i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości (Dzwonek) ministra sprawiedliwości Tajwanu. Apelujemy o wzmożone kontakty międzynarodowe zmierzające do jej zniesienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów i Konserwatyści przedstawi pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest to dokument dość kuriozalny począwszy od tytułu, bo mówi się o tym, że jest to projekt ustawy o zasadach współpracy między Rzecząpospolitą Polską - to wszyscy rozumieją - i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości ministra sprawiedliwości Tajwanu.

Jednocześnie, żeby było zabawniej, jeśli tak to można określić, my mamy polskie biuro w Tajpej, a Tajwan ma swoje biuro w Warszawie. Szef tego biura ma status ambasadora. Może jest ambasadorem tytularnym.

To jest dość, powiedziałbym, nietypowe. Z pewnym zdumieniem dowiedziałem się, że Polska jest centrum przestępstw w cyberprzestrzeni, które dotykają Tajwanu.

Chińczycy nie uznają Tajwanu za osobne państwo, ale podpisują z nim umowy międzynarodowe.

Klub PSL - Koalicji Polskiej - Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów zagłosuje za. Dziękuję bardzo panu posłowi. Bardzo proszę, panie pośle. Nie mam zastrzeżeń co do samej ustawy. Nie ma tam chyba niczego kontrowersyjnego, co nie byłoby znane z innych tego typu ustaw, poza jedną rzeczą - poza hipokryzją. Dokonujemy jakichś logicznych szpagatów w tytule, żeby nie nazwać Tajwanu państwem, tylko terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości ministra sprawiedliwości Tajwanu. Skoro jednak przyjmujemy do wiadomości, że istnieje minister sprawiedliwości Tajwanu i kontroluje sytuację na jakimś terytorium, to chyba przyjmujemy też do wiadomości, że istnieje Tajwan i właśnie to terytorium zajmuje.

Chin do siebie nawzajem, do władzy nad całością. Uznawanie komunistycznych Chin i nieuznawanie Tajwanu jest jakąś formą legitymizacji urojeń chińskich komunistów dotyczących władzy nad Formozą. Tajwan nie pyta nikogo, czy mu wolno wyciąć kornika gdzieś w lesie, Tajwan nie daje się upokarzać, nie tłumaczy się przed innymi z reform sądownictwa we własnym kraju, nikt mu nie grozi procedurami sprawdzania praworządności. Tajwan nie opowiada swoim obywatelom, że ich pomyślność zależy od tego, że się gdzieś zapiszą i jak będą grzeczni, to dostaną dotacje. Tajwan rozwinął się dużo lepiej niż Polska bez żebractwa, tylko dzięki pracy i w miarę wolnemu rynkowi, bez jakiejś idealizacji, ale - jak widać - tyle wystarczyło. Co więcej, Tajwan rozwija się mimo skrajnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, gdy tymczasem nasi tchórzliwi, na zewnątrz sterowni politycy mówią, że Polska nie może sobie na niepodległość pozwolić, bo leży między wschodem i zachodem, przecież zupełnie inaczej niż inne kraje, które nie mają nikogo na wschodzie ani na zachodzie. Ba, w czasie kiedy cała Unia Europejska potyka się o własne nogi w swojej nieudolnej polityce w zakresie walki z pandemią, Czyli Tajwan radzi sobie 2053 razy lepiej niż Polska. Zamiast więc oglądać się na wytyczne z Brukseli, czyli stolicy państwa, które ma najwyższy wskaźnik śmierci na 1 mln mieszkańców, może spytajmy ekspertów z Tajwanu, jak to się robi. Tak czy inaczej jest niedorzeczne, że Polska nie uznaje niepodległości Tajwanu, a oczekuje uznania własnej, której ma mniej. Tak więc uznajmy niepodległość Tajwanu, zanim oni przestaną uznawać naszą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym wystąpienia klubowe zostały zakończone. Do pytań zapisało się trzech panów posłów. Bardzo proszę. Jeżeli nie, to zamykam listę, ustalając czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Chciałem zapytać o kwestię kary śmierci, ponieważ w tej konwencji, w tej umowie nie ma nic na ten temat. Pytanie: Czy rząd w ogóle w jakikolwiek sposób rozmawiał o tym i próbował wprowadzić do tego porozumienia kwestię np. zakazu wykonywania tego wobec osób, które zostały na podstawie art. 4 poddane ekstradycji, na terytorium Tajwanu w związku z popełnieniem przez nie przestępstw? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Andrzeja Szejnę, klub Lewica, o zadanie pytania. Wysoka Izbo! Wiem, że on się zapatrzył na Tajwan, bo tam akurat jest możliwa kara śmierci.

Przed chwilą mieliśmy do czynienia z dyskusją o konwencji stambulskiej, o prawach kobiety. Otóż Sąd Rejonowy w Kielcach oddalił, umorzył postępowanie, które było wszczęte przeciwko dyrektorce mojego biura, feministce, Małgorzacie Marenin, która protestowała przed katedrą kielecką w walce pod hasłem: stop pedofilii w Kościele w czasie pandemii, twierdząc, że jej działanie jest zmotywowane szlachetnymi pobudkami, panie pośle. Tak jak pan nie rozumie szlachetnych pobudek pań posłanek, które występowały w imieniu Lewicy, broniąc praw kobiet, broniąc ich w obliczu przemocy, broniąc ich godności, szacunku, tak nie zrozumie pan oczywiście tego, co uczynił sąd w Kielcach, broniąc prawa do szlachetnej demonstracji przeciwko pedofilii w Kościele, tak nie zrozumie pan innych kwestii, które są związane z prawami człowieka, ale będę dążył (Dzwonek) do tego, żeby pana do tego przekonać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana posła Tomasza Piotra Nowaka o zadanie pytania. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

Rozumiem, że ona rośnie w tej chwili.

Zanim udzielę głosu panu ministrowi Romanowskiemu, w trybie sprostowania głos zabierze pan poseł Dobromir Sośnierz. Niestety, pan poseł Szejna już wyszedł i. To proszę przekazać.

Chciałem zapytać, skoro mówimy o tym, że. Bo pan oskarżył mnie o to, że ja nie rozumiem tego wysiłku, tego szlachetnego wysiłku posłanek, które walczą tutaj o konwencję stambulską. Chciałem zwrócić uwagę, że pani Lubnauer weszła tu i powiedziała, ile to kobiet było tutaj pobitych w ostatnich miesiącach. W związku z tym ta konwencja stambulska nie działa. W związku z tym właśnie uważam, że jest to działanie iluzoryczne i niepotrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ja także nie rozumiem w takim razie. Co pan chce sprostować, skoro nie zrozumiał pan wypowiedzi pana Szejny?

Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, w zakresie kary śmierci jest to oczywiście uregulowane za pośrednictwem tego przepisu, do którego odwoływał się pan poseł, a mianowicie przepis mówi o stosowaniu odpowiednio prawa krajowego, prawa polskiego, natomiast nasz Kodeks postępowania karnego w art. 604 § 1 pkt 6 jako niedopuszczalność wydania, jako negatywną przesłankę ekstradycji wskazuje właśnie uzasadnioną obawę, że w państwie żądającym wydania wobec osoby wydawanej może zostać orzeczona lub wykonana kara śmierci.

Jeżeli chodzi o relacje polsko-tajwańskie, to pewnym obrazem tego.

A więc tak wygląda ta skala współpracy prawnej w zakresie prawa karnego. Jeżeli chodzi o inne relacje, o inne porozumienia, które regulują ze stroną tajwańską tego typu zagadnienia, to tak jak już wcześniej wspomniał pan poseł Bartoszewski, również Chińska Republika Ludowa zawarła takie porozumienie, tak samo jak Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi natomiast w ogóle o regulacje dotyczące przeciwdziałania cyberprzestępczości, to może nie jestem tutaj specjalistą, tym bardziej od regulacji dalekowschodnich, ale one mają dość podobny charakter i stan rozwoju, jeśli można się tak wyrazić, jak nasze regulacje, co zresztą wiemy na podstawie współpracy, właśnie tej prawnej, między naszymi organami ścigania.

Dzięki temu w sposób kompleksowy, tak samo zresztą jak inne państwa wcześniej wspomniane, będziemy mieli uregulowane nasze relacje w zakresie stosowania prawa karnego w obrębie działania sądów i prokuratur. Warto tu jeszcze dodać, że oczywiście to nie jest klasyczna umowa międzynarodowa.

Rzeczywiście jest tak, że Tajwan ma specyficzny status prawny, stąd właśnie to narzędzie, które już wcześniej było wykorzystywane do transpozycji prawa zapewniającego unikanie podwójnego opodatkowania.

Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Ponieważ na sali nie ma sprawozdawcy komisji, zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o rezerwach strategicznych, druk nr 839. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o rezerwach strategicznych (druki nr 829 i 839) Bardzo proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W imieniu sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przedstawiam sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o rezerwach strategicznych, druk sejmowy nr 839. Sejm na 23. posiedzeniu w dniu wczorajszym na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. W trakcie wnikliwej, prawie 3-godzinnej debaty komisyjnej zgłoszone zostały liczne poprawki merytoryczne i legislacyjne, których większość komisja uwzględniła w załączonym do sprawozdania projekcie ustawy o rezerwach strategicznych. Ustawa ta powołuje Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na bazie istniejącej Agencji Rezerw Materiałowych w celu usprawnienia rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony do sprawozdania komisji projekt ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Otwieram dyskusję.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące rządowego projektu ustawy o rezerwach strategicznych. Miniony rok, nieprzewidywalna sytuacja związana z epidemią koronawirusa, nadzwyczajny kryzys społeczno-gospodarczy obnażyły ułomność wielu instytucji, warunków, w jakich dotychczas one funkcjonowały, pomimo że szczególnie skutecznie powinny pracować właśnie w takich trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach. To dotyczy tak kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków instytucji, jaką jest Agencja Rezerw Materiałowych, która mocą procedowanej ustawy będzie nosiła nazwę: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Chcąc skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, jakie postawiła przed nami rzeczywistość, nieść pomoc Polakom, zapewnić im realne bezpieczeństwo, agencja, która stanowi istotny element całego systemu wsparcia krytycznego państwa, powinna być instytucją sprawnie i szybko reagującą na pojawiające się kryzysy. Temu służą zmodyfikowane zapisy określające nowe, szersze zasady działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wprowadzone modyfikacje wynikają z nabytych doświadczeń związanych z walką z epidemią koronawirusa i niewydolności dotychczasowych rozwiązań prawnych. Stąd też przyjęcie tej ustawy jest nie tylko oczekiwane, ale wręcz pożądane, bo jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze w zarządzaniu państwem ceniliśmy sobie skuteczność i realny wymiar podejmowanych działań w przeciwieństwie do wielu naszych politycznych konkurentów, w przypadku których liczył się PR i przekonanie, że jakoś to się potoczy. Ustawa wprowadza zmiany mające na celu bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży niektórych towarów i dóbr na rynku oraz popycie na nie, ma zabezpieczyć życie i zdrowie obywateli. Jej celem jest uproszczenie i uelastycznienie procedur, w oparciu o które działa Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Znamy, szanowni państwo, stanowiska polityków Platformy Obywatelskiej i Lewicy, którzy bardzo często czy to na posiedzeniu komisji, czy w debacie w czasie posiedzenia na sali plenarnej, podkreślali, podnosili argumenty, jakobyśmy nie powinni przyjmować tej ustawy w tym momencie, pytali, po co ją przyjmujemy. Przepraszam bardzo, ale na co mamy czekać? Sugestie, by odłożyć w czasie wejście w życie tej ustawy, są antypaństwowe, są sprzeczne z polską racją stanu, interesem obywateli, i tak naprawdę wpisują się w narrację tych, którzy życzą naszej ojczyźnie jak najgorzej. Projektowana ustawa reguluje przede wszystkim zagadnienia z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych, a także ich finansowania. Rozbudowany zostaje także zakres zadań realizowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, dla których realizacji tworzone są rezerwy strategiczne, poszerzono również katalog asortymentu niezbędnego do osiągania celów określonych w art. 3 przedmiotowej ustawy, co pozwoli lepiej reagować na szybko zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze-polityczne. Nowa ustawa zapewnia lepszą koordynację działań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która będzie podlegała prezesowi Rady Ministrów jako organowi nadzorującemu, co jest uzasadnione i potrzebne z uwagi na to, iż to właśnie premier jest koordynatorem zarządzania kryzysowego na szczeblu centralnym, będąc jednocześnie przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. To również premier będzie organem właściwym do wydawania decyzji dotyczących udostępniania rezerw. Szereg przepisów zawartych w projekcie ustawy umożliwia szybsze i sprawniejsze działanie agencji, m.in. poprzez odformalizowanie procedur zakupowych czy zasad tworzenia rezerw lub zawierania umów związanych z przechowywaniem rezerw, zawsze jednak będzie to się odbywało z zastosowaniem przejrzystych, niedyskryminacyjnych i konkurencyjnych warunków wyłaniania kontrahentów. Takie rozwiązanie będzie sprawdzać się szczególnie w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Ustawa poszerza zadania agencji o nowe obszary, w szczególności o usługi transportowo-logistyczne, a także zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami, których właścicielem jest agencja lub które znajdują się w jej posiadaniu, co przyczyni się do większej operacyjności i efektywności jej działań. Projekt reguluje także katalog osób objętych obowiązkiem w zakresie ograniczenia prowadzenia działalności oraz składania okresowych oświadczeń o stanie majątkowym, co zapewni większą przejrzystość działania. Zabezpieczy to również Skarb Państwa przed ewentualnymi nadużyciami finansowymi ze strony pracowników agencji. Wszystkie działania są i będą transparentne, a podejmowane w interesie obywateli są i będą również konieczne. A więc, szanowni państwo, jawnie, przejrzyście, sprawnie i zgodnie z prawem działają instytucje pod kierunkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, w przeciwieństwie do instytucji działających pod kierunkiem tych, którzy w Polsce już przecież rządzili przez 8 lat i chętnie chcieliby nadal działać ukradkiem, po cichu, pod stołem, od czasu do czasu naradzając się na cmentarzach lub parkingach. Wysoki Sejmie! Ustawa jest nie tylko potrzebna, ale przede wszystkim jest oczekiwana. Klub Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy i rekomenduje jego przyjęcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę pana posła Sławomira Neumanna, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Ale jeżeli uważacie, panowie i panie z PiS-u, że nadzór bezpośredni premiera będzie jakąś czarodziejską różdżką, która usprawni działanie tej agencji, to jesteście w błędzie, bo do tej pory premier podejmował decyzje polityczne o zakupie węgla przez Agencję Rezerw Materiałowych. To premier podejmował decyzje, że spółki Skarbu Państwa będą kupować maseczki czy inny sprzęt ochrony osobistej. Tempo prac jest kompletnie nieprzystające do materii tej ustawy i do rzeczywistych potrzeb, bo jak mówię, większość tych wszystkich zapisów znajduje się w innych ustawach i z nich korzystacie. Ta ustawa nie daje wam żadnych dodatkowych uprawnień. Czy uważacie, że zapisanie możliwości kupowania poza ustawą o zamówieniach publicznych coś przyspieszy lub coś wam ułatwi? Przecież dzisiaj takie rozwiązania są zawarte w ustawach COVID-owych, przecież przez cały okres pandemii kupowaliście właściwie z pominięciem procedur mnóstwo różnego rodzaju materiałów, sprzętu.

Do dzisiaj tych respiratorów nie ma, pieniędzy też nie ma, pieniądze przepadły. Jeżeli tak naprawdę wyciągacie wnioski z tych prawie już kilkunastu miesięcy pandemii, to powinniście działać dokładnie odwrotnie, czyli nie zdejmować tych procedur i tego kagańca procedur z siebie, tylko działać dokładnie odwrotnie, czyli przestrzegać procedur, żeby one były jasne, czytelne, procedury zakupowe. Tu jest jak zwykle w tej ustawie zapisane, mówicie mniej więcej tak: dajcie nam wolną rękę, my wydamy miliony czy miliardy bez żadnych ograniczeń, kupimy wszystko tam, gdzie nam się podoba i gdzie będzie taka ochota. To jest błędne myślenie. Jedyną zmianą, żeby takie zakupy robić, jest to, że rzeczywiście teraz agencja będzie podlegała pod prezesa Rady Ministrów. Można będzie powiedzieć, że ludzie od Morawieckiego będą kupować, a nie ludzie od Szumowskiego czy od Sasina. No to będzie duża zmiana, rzeczywiście. Tylko czy po to, żeby zmienić ekipę, która będzie tych zamówień dokonywać, trzeba zmieniać całą ustawę, trzeba zmieniać system zarządzania tą agencją w czasie pandemii, kiedy ta agencja naprawdę powinna być przydatna państwu i pomagać Polakom? Wy teraz ciężko pracujecie, żeby trzecia fala pandemii była dla was także zaskoczeniem, bo pierwsza fala pandemii zaskoczeniem była, druga zaskoczeniem jest, trzecia pewnie będzie, bo wy zamiast myśleć o tym, jak zabezpieczyć Polskę, jak zabezpieczyć Polaków na trzecią falę pandemii, zajmujecie się teraz gierkami organizacyjnymi, jak tu zmienić podległość agencji, żeby ktoś inny decydował o zakupach, żeby ktoś inny decydował o władzach tej agencji. To jest wprowadzanie zamieszania i bałaganu do instytucji, która i tak z jakiejś superorganizacji nie słynie. Więc pytanie jest: Po co to robicie dzisiaj w takim momencie, kiedy rzeczywiście powinno to działać znacznie, znacznie lepiej? Czy nie lepiej zamiast przepychać się o to, kto będzie robił i nadzorował nową agencję, nie powinniście powiedzieć Polakom, że ta agencja już np. zakupiła czy zamówiła 70 mln strzykawek, bo tyle będzie potrzebne do zaszczepienia Polaków szczepionką COVID-ową? Jest niezliczona ilość konferencji prasowych premiera czy ministra zdrowia mówiących o tym, jak jesteście superprzygotowani do szczepienia Polaków szczepionką na COVID, ale nie słyszeliśmy, żeby rzeczywiście zabezpieczyć te 70 mln strzykawek, bo tyle będzie. Dzisiaj pan minister mówi o tym, że w każdej gminie będzie punkt szczepień. Czy agencja już zamówiła te lodówki, żeby dostarczyć tym gminom, żeby mogły spokojnie przechowywać te szczepionki? My tylko słyszymy o tym, że należy zmienić nazwę agencji na rządową. I tak dobrze, że nie narodową, bo to mogła być jeszcze narodowa agencja rezerw materiałowych - wtedy by na pewno się wszystko udało. Więc uważam, że w tym przypadku ustawa jest niepotrzebna, zbędna w tej chwili i szkodliwa, i nie ma co przeszkadzać w tak trudnej sytuacji tym ludziom w pracy. Dlatego składamy wniosek o jej odrzucenie.

Dziękuję bardzo panu posłowi za wystąpienie i złożenie poprawek. A teraz głos zabierze pan poseł Wiesław Szczepański, który przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie nasze stanowisko odnośnie do projektu ustawy o rezerwach strategicznych, zawartego w drukach nr 829 i 839. Debatujemy dziś nad ustawą w iście ekspresowym tempie. W środę otrzymaliśmy projekt ustawy, we wtorek było pierwsze czytanie, dzisiaj jest drugie czytanie i uchwalenie ustawy. W ostatnim okresie mieliśmy mnóstwo konferencji prasowych, informacji o zakupach, wyprzedażach z agencji, że jesteśmy gotowi na COVID, mamy zapasy, a potem okazało się, że król jest nagi. Chciałbym zapytać: Jak agencja jest przygotowana, o czym mówił mój przedmówca, do masowej skali szczepień? Czy mamy zapasy strzykawek, igieł, innego sprzętu, ale również sprzętu chłodniczego? Po co ta zmiana w ogniu walki z COVID-em? Czy nie należałoby z tym poczekać do momentu odejścia wirusa? Zastanawiam się, czy w świetle obecnych działań rządu w ogóle ta agencja jest potrzebna.

Agencja zmienia dzisiaj tylko nazwę. Czy zmiana nazwy będzie lekarstwem na jej złe działanie? Czy jest to brak zaufania do ministra aktywów państwowych, że podchodzi ona pod nadzór premiera?

Mimo że procedowana ustawa ma wpływ na wiele podmiotów, szacuje się, że z prawie 100 tys. przedsiębiorstw, samorządami, Strażą Graniczną, strażą pożarną, z tymi podmiotami w ogóle nie była konsultowana. Domniemam, że tak szybka zmiana może mieć na celu ukrycie niektórych nieprawidłowości, które miały miejsce w tej agencji. Chciałbym zapytać, panie ministrze: Ile ta agencja zakupiła węgla, a właściwie miału w ostatnich latach? Ile z tego sprzedała? Ile wydała na to milionów i ile leży jeszcze w tej agencji niezagospodarowanych? Obchodzimy tą ustawą, jak mówili moi koledzy, również ustawę o zamówieniach publicznych. Ustawa określa m.in. zasady tworzenia, utrzymania, udostępnienia, likwidacji oraz finansowania rezerw strategicznych, a także zadania i organizacje dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ale chciałbym zapytać również o kwestie kadrowe. Otóż czytam tę ustawę i mamy tam napisane, że prezesa agencji powołuje premier, ale prezes ma zastępcę lub zastępców. To chciałbym się dowiedzieć ilu: dwóch, trzech, pięciu czy też, powiedzmy, tylu, ile będzie potrzebnych stanowisk, dlatego że państwo nie określiliście maksymalnej liczby zastępców, tylko pojawiło się określenie „zastępców”, czyli jeden będzie, nie wiem, od paliw, drugi będzie od węgla, trzeci będzie od strzykawek, czwarty będzie jeszcze od czegoś innego. Chciałbym dowiedzieć się, jak wielka będzie liczba tych zastępców. O ile jeszcze dodatkowo wzrosną koszty funkcjonowania tej agencji? Chciałem powiedzieć, że mój klub wstrzyma się podczas głosowania nad tą ustawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi za przedstawienie stanowiska klubu parlamentarnego Lewica.

Przepraszam bardzo. Pana ministra też przepraszam. Jeszcze chwila. Jeżeli nie ma więcej chętnych posłów, to zamykam listę, ustalając czas na zadanie pytania na 1 minutę. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Tomasz Piotr Nowak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie ministrze, respiratory są na razie w Agencji Rezerw Materiałowych. Proszę powiedzieć czy te respiratory są z certyfikatami i jaka jest historia tych przesyłek, które doleciały wielkim Antonowem i zostały przyjęte przez Agencję Rezerw Materiałowych. Panie ministrze, drugi rząd robicie. Premier Morawiecki chce przejąć tę agencję, pewnie będzie miał apetyt na wiele innych agencji. Czy to wynika z tego, że jest niedowład, jakiś brak efektywnego zarządzania, kierowania tymi ministrami?

Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Proszę o zadanie pytania. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście przez lata rząd PiS wykorzystywał rezerwy strategiczne do tak naprawdę pewnych ruchów politycznych.

Mam proste pytanie, test na prawdę, panie ministrze. Ile poświęciliście środków przez ostatnich 5 lat na realizowanie takich propagandowych projektów, jak np. zakup węgla czy zakup respiratorów od handlarza bronią itp. Jeżeli państwo przyjdą do parlamentu, wyspowiadają się z tych grzechów, to być może zaczniemy wierzyć w to, co tu przedstawiacie. A na razie to czysta propaganda. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Gadowskiego, Koalicja Obywatelska, o zadanie pytania. Panie Ministrze! Czy uważa pan, że dzisiaj, w tej sytuacji gospodarczej, w sytuacji pandemii to jest właściwy moment na wprowadzenie tej ustawy w życie?

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego, Prawo i Sprawiedliwość, o zadanie pytania. Wysoki Sejmie! Obecnie poprzez Agencję Rezerw Materiałowych rząd dokonuje zakupów środków medycznych oraz wszystkich innych, związanych z kryzysem zdrowotnym, z obecną pandemią. Panie ministrze, czy i w jakim zakresie ta ustawa usprawni walkę z pandemią? Dlaczego w ogóle działania strategiczne państwa w związku z tą ustawą będą sprawniejsze? Obecna sytuacja to nie jest już poligon, to jest realny sprawdzian w boju możliwości państwa. Chciałbym także w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyć wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o rezerwach strategicznych, druki nr 829 i 839, bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu, po doręczeniu ich posłom.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak tak posłuchać relacji rządu, jak sobie radzi z pandemią, to od sukcesu - do sukcesu.

Wtedy, kiedy jedna z koleżanek chciała złożyć poprawkę wymagającą zabezpieczenia gwarancji bankowych od kontrahentów - to będzie bez przetargu, bez zamówień publicznych, ale chociaż z gwarancją bankową - usłyszeliśmy, że nie jest to potrzebne, bo są inne instrumenty. Po co gwarancje bankowe, skoro można się zabezpieczyć np. kamizelkami kuloodpornymi?

Mam pytanie.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jednocześnie Agencja Rezerw Materiałowych była słynna na początku roku, gdy skupowała węgiel do magazynu w Ostrowie Wielkopolskim.

Kto jest odbiorcą tego węgla? Mamy wrażenie, że wam już Sejm jest.

Dziękuję bardzo. Jako ostatni pytanie zada pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podczas dyskusji nad projektem ustawy widać bardzo wyraźnie, bardzo dobitnie, jaką logiką kierują się przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, którą niestety trzeba nazwać totalną opozycją. Otóż logika ta mówi: im gorzej dla Polski, tym lepiej dla opozycji.

Chciałbym zapytać: W jaki sposób ustawa wpłynie na usprawnienie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, dostępu Polaków do najważniejszych materiałów i towarów? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym lista posłów zapisanych do pytań została wyczerpana.

Chciałbym rzeczywiście odnieść się do kilku pytań.

To, jak bardzo ważny jest, okazało się właśnie w czasie pandemii. Nie przygotowaliśmy tej agencji do walki z pandemią - ani my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, ani wy - rząd Platformy Obywatelskiej, ani wcześniej rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Tak naprawdę ta ustawa jest kolejnym etapem zmian, które są wprowadzane. Tak, były.

Podobne zmiany, gdzie agencje tego typu są przesuwne pod ośrodek premierowski, mają miejsce w Danii, w Rumunii i w innych krajach, które wyciągnęły wnioski z pandemii. Dlaczego? Dlatego, że Agencja Rezerw Materiałowych zajmuje się tak szeroką gamą problemów i jej zadania idą w poprzek tylu różnych resortów, że rzeczywiście zasadne jest umiejscowienie jej w centrum rządu. To jest taka uwaga natury ogólnej.

Sytuacja wygląda w ten sposób. My nie kupujemy lodówek do każdej gminy. Pan zarzuca nam z jednej strony, że za dużo mówimy o przygotowaniach do programu szczepień, bo premier czy któryś tam minister wychodzi i o tym opowiada. A mówimy o tym dlatego, że dzisiaj w całej Europie wszystkie rządy starają się jak najwięcej mówić o programie szczepień, i to jest nasze wspólne zadanie. Mówię o całym parlamencie. Chodzi o to, żeby przekonywać obywateli do tego, że szczepienia są potrzebne, że wszyscy powinni się zaszczepić, że ten proces przygotowań jest transparenty i dobrze zaplanowany, bo tylko wtedy, gdy Polacy będą mieli poczucie bezpieczeństwa, będą chcieli się zaszczepić, a to jest w naszym wspólnym narodowym interesie.

To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia jest taka.

Właśnie o tym, jak ta agencja była traktowana, świadczy też to, gdzie była, bo ona była już pod nadzorem ministerstwa gospodarki, ministerstwa energii, ministerstwa klimatu i Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Proszę państwa, te przepisy, które proponujemy - a które wyłączają zakupy tylko w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, bo przecież wszystkie inne zakupy, które robi agencja, są normalnie poddane przepisom o zamówieniach publicznych - wprowadzamy po to, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji jak w czasie COVID-u, gdy musieliśmy na szybko wprowadzać przepisy na czas pandemii, na czas walki z COVID-em. Tu chcemy zadziałać wyprzedzająco.

Zgłoście taką poprawkę, a my bardzo poważnie się nad tym zastanowimy, dlatego że rzeczywiście to jest jeden z takich elementów funkcjonowania państwa, co do którego powinniśmy unikać sporów politycznych. Jeśli to ma wzbudzić wasze zaufanie do tych zmian, to uważam, że warto rozważyć taką poprawkę. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Krótko pan poseł Sławomir Neumann. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Myśmy się nie zrozumieli. To jest oczywiste, że należy zachęcać do szczepień. Każdy rozsądny człowiek będzie zachęcał do tego, żeby zaszczepiło się maksymalnie dużo Polaków. Czy to w programie narodowym, ogólnopolskim, nieważne jak nazwanym. Ja tylko mówię, że jeżeli ma być to skuteczne, to musimy zaszczepić miliony Polaków. Zresztą państwo też o tym mówią. Mówicie, że właściwie jesteśmy gotowi zaszczepić wszystkich. Czyli trzeba mieć 70 mln strzykawek i trzeba mieć odpowiednią ilość punktów szczepień, żeby nie szczepić przez 10 lat, tylko szybko.

Trochę więcej w miastach, w dużych ośrodkach, ale tych punktów szczepień musi być odpowiednio dużo.

Mówimy więc z pełną odpowiedzialnością o tym, że należy przygotować ten program jak najlepiej, bo szczepionka może zahamować wirusa. Wierzę w to, że tak będzie i że będziemy wszyscy razem pokazywać, że się szczepimy i że to jest program, który - niezależnie od nazwy - będzie skutecznym remedium na pandemię. Jako ostatni głos w dyskusji zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Krzysztof Tchórzewski. Proszę bardzo. Wysoki Sejmie! Mimo tej gorącej debaty chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim posłom i stronie rządowej za merytoryczną i wnikliwą dyskusję na prawie 3-godzinnym posiedzeniu komisji, gdzie widać było jednak, mimo różnic politycznych, bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże zaangażowanie, jeśli chodzi o prace nad uchwaleniem tej ustawy. Rozpatrywany projekt ustawy jest jednak bardzo istotny, dlatego że w tym, co się dotychczas działo, czyli w zakresie walki z COVID-19, można było nie na poligonie, ale w boju sprawdzić możliwości państwa i możliwości działania tej ustawy, która dotychczas obowiązywała, czyli o Agencji Rezerw Materiałowych.

Jeszcze raz jednak dziękuję za wszystkie uwagi i chcę podkreślić, że poprawki opozycji także były przyjmowane na posiedzeniu komisji.

Dziękuję bardzo panu posłowi. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez odsyłania do komisji. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Na tym wyczerpaliśmy w tym momencie porządek naszego posiedzenia. Ogłaszam przerwę do godz. 18.30.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Bardzo proszę.

posiedzeniu bierze udział 441 posłów. Przypominam, że Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni złożył wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji panującej w elektrowni w Ostrołęce. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o ten punkt. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie w tej sprawie nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji panującej w elektrowni w Ostrołęce. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowania podmiotów leczniczych na zwiększoną liczbę zachorowań na COVID-19 oraz działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął informację do wiadomości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił wniosek, a tym samym przyjął informację do wiadomości. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 819-A. Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i niektórych innych ustaw. Komisja w dniu dzisiejszym rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 819. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Z poprawką tą łączy się poprawka 4. Głosujemy.

Przyjęcie tej poprawki spowoduje zmianę tytułu ustawy. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Przyjęcie tej poprawki spowoduje zmianę tytułu ustawy.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 819, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 812-A. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie dodatkowego sprawozdania Komisji. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Do projektu ustawy o rozliczeniu ceny lokalu lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości w trakcie drugiego czytania zostały złożone cztery poprawki. W dniu dzisiejszym Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły te poprawki i rekomendują Wysokiej Izbie poprawkę 1. odrzucić. Ona się odnosi do art. 4, określającego zasady podejmowania uchwały przez właściwą radę gminy. Odrzucenie tej poprawki jest wskazane dlatego, że określenie sztywnej granicy 35% jako minimum powierzchni użytkowej lokali lub budynków przekazywanych gminie może eliminować takie sposoby pozyskania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, gdzie cena gruntów jest niższa, bo przecież ta wymiana musi być ekwiwalentna.

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 812. W dodatkowym sprawozdaniu komisje przedstawiają poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Sejm poprawki przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 812, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2019 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął sprawozdanie do wiadomości. Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania zawartego w druku nr 292. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie sprawozdania zawartego w druku nr 292, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym przyjął sprawozdanie do wiadomości. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 796-A. Proszę panią poseł Barbarę Bartuś o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Mam przyjemność przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Podczas drugiego czytania zgłoszono dziewięć poprawek, które na dzisiejszym posiedzeniu komisja rozpatrzyła. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 796. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Ich przyjęcie spowoduje zmianę tytułu ustawy, co jest treścią poprawki 1. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 796, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 732. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Wnioski mniejszości zgłoszone zostały do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zwierającego zmiany do ustawy Kodeks postępowania karnego. Z wnioskiem tym łączy się 2. wniosek mniejszości. Nad tymi wnioskami głosować będziemy łącznie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Głosujemy nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 732, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 822. Komisje przedstawiają również wniosek mniejszości, nad którym głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy.

Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania na całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 822, zechce nacisnąć

Sejm uchwalił ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 831. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 831, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości ministra sprawiedliwości Tajwanu. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Głos ma poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska.

Rozpoczynamy wygłaszanie oświadczeń poselskich.

Bardzo proszę, panie pośle. Czy jest pan poseł?

Wysoka Izbo! Nigdy w historii ostatnich 30 lat nie było tak upolitycznionego rządowego finansowego rozdania jak w przypadku Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Fundusz nie miał dzielić, miał ożywić gospodarkę w całej Polsce, miał przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-u, miał wesprzeć rozwój lokalny, miał być ogólnopolskim impulsem dla rozwoju, tymczasem stał się wykluczający dla wielu miast, gmin i powiatów. Stał się lekceważący dla mieszkańców regionu, gdzie nie dotarła ani jedna złotówka, a przecież wszyscy i wszędzie płacimy takie same podatki. Stał się nieobiektywnym batem dla tych burmistrzów, wójtów i starostów, którzy nie chcą partyjnie wiązać się z PiS-em. Setki samorządów nie otrzymały w ostatnim naborze ani złotówki.

Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Będę kontynuować to, co powiedziała pani poseł Wielichowska na temat sytuacji na Dolnym Śląsku. I tak: Bolesławiec - zero, Osiecznica - zero, Warta Bolesławiecka - zero. Paszowice - zero, Wądroże Wielkie - zero, gminy górskie, będące w trudnej sytuacji, Jelenia Góra - zero, Karpacz - zero, Kowary - zero, Szklarska Poręba - zero. Stara Kamienica - zero, Lubawka - zero, Marciszów - zero, Zgorzelec - zero, gmina wiejska Zgorzelec - zero, Sulików - zero, Zawidów - zero, Pieńsk - zero, Leśna - zero, Gryfów Śląski, najbiedniejsze gminy - zero, Lubomierz - zero, Lwówek Śląski - zero, gmina Pielgrzymka - zero, gmina Świerzawa, o najniższych dochodach na mieszkańca - zero, Złotoryja - zero, Zagrodno - zero. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Często są to gminy o najwyższym poziomie bezrobocia, które nie uzyskały wsparcia. Wymienię: gmina Oborniki Śląskie - zero, gmina Prusice - zero, powiat głogowski - zero, gmina Strzelin - zero, gmina Kondratowice - zero, gmina Wiązów - zero, gmina Przeworno - zero, gmina Szczytna - zero, gmina Chojnów - zero, gmina Ścinawa - zero, gmina Milicz - zero, gmina Twardogóra - zero, gmina Międzybórz - zero, gmina Chocianów, jedna z najbiedniejszych na Dolnym Śląsku - zero, gmina Malczyce - zero, gmina Wisznia Mała - zero, gmina Żmigród - zero, gmina Brzeg Dolny - zero, gmina Wińsko, także jedna z najbiedniejszych rolniczych gmin - zero, gmina Wołów - zero, gmina Wrocław i powiat wrocławski - zero, gmina Długołęka - zero, gmina Kąty Wrocławskie - zero. To jest lista, która powinna być listą waszych wyrzutów sumienia. względem mieszkańców, którzy oczekiwali na pomoc. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Tomasz Lenz, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Skandal, jaki ma miejsce w związku z podziałem środków na inwestycje lokalne, dotyczy tego, że PiS chce po prostu dawać te pieniądze wyłącznie tym, którzy jedzą im z ręki, którzy im się kłaniają. a nie tym, którzy pieniądze potrafią dobrze wydać na potrzeby mieszkańców. Pieniądze nie mają barwy politycznej. Mieszkańcy czekają na chodniki, ulice, obiekty sportowe, przedszkola. A PiS chce, żeby w gminie, gdzie wójt popierał PiS, takie przedszkole powstało, a w gminie, gdzie wójt popierał Rafała Trzaskowskiego w ostatnich wyborach, takiego przedszkola nie było. A co to ludzi obchodzi? Co robi PiS? Dzieli Polaków na lepszych i gorszych. Powiaty takie jak bydgoski, chełmiński, grudziądzki, lipnowski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, wąbrzeski, żniński - zero dofinansowania na inwestycje. Gminy w Kujawsko-Pomorskiem - w powiecie aleksandrowskim: gmina Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, Waganiec - zero dofinansowania. Powiaty, które chcę następnie wymienić - proszę chwilę zaczekać, elektronika ma swoje prawa i tym razem nieco mnie zawiodła, ale zaraz będziemy mogli. Mam nadzieję, że to nie jest działanie ministra Schreibera z Kujawsko-Pomorskiego, który nie docenił swojego własnego regionu i nie dał pieniędzy także w swoim województwie. Powiat brodnicki: gmina Bartniczka, gmina Brodnica, gmina Górzno, gmina Jabłonowo Pomorskie, gmina Osiek, gmina Świedziebnia - zero dofinansowania. W powiecie bydgoskim: gmina Dąbrowa Chełmińska, gmina Dobrcz, gmina Osielsko, gmina Solec Kujawski - zero dofinansowania. Powiat chełmiński: gmina Chełmno, gmina miasto Chełmno, gmina Popowo Biskupie, gmina Stolno, gmina Unisław - zero dofinansowania. Powiat golubsko-dobrzyński: gmina Ciechocin, gmina Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń - zero dofinansowania. Gmina Łasin, gmina Radzyń Chełmiński, gmina Rogoźno, gmina Świecie nad Osą - zero dofinansowania. Powiat inowrocławski: gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Inowrocław gmina miejska, Inowrocław gmina wiejska, Janikowo, Rojewo - zero dofinansowania. Powiat lipnowski: gmina Bobrowniki, Kikół, Lipno, Tłuchowo, Wielgie - zero dofinansowania. Powiat mogileński: Dąbrowa, Mogilno, Strzelno - zero dofinansowania. W powiecie nakielskim nic nie otrzymała gmina Kcynia. Powiat radziejowski: Dobre, Piotrków Kujawski, Radziejów - zero dofinansowania.

Powiat świecki: Dragacz, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie - zero dofinansowania. Powiat ziemski toruński: Chełmża gmina wiejska, Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka - zero dofinansowania. Powiat tucholski: gmina Cekcyn - zero dofinansowania. Powiat włocławski: Baruchowo, Chodecz, Fabianki, Kowal miejska, Kowal gmina wiejska, Lubanie, Lubraniec, Włocławek gmina wiejska - zero dofinansowania. Jesteśmy oburzeni tak jak samorządowcy i mieszkańcy naszego regionu, że tak zostaliśmy potraktowani. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Rząd obiecał samorządom pomoc i wsparcie na inwestycje w związku z kryzysem. Pieniądze zostały rozdzielone nie według kryteriów czy algorytmu, tylko według klucza politycznego. W województwie lubelskim, które jest jednym z najbiedniejszych w Polsce i w całej Unii Europejskiej, ta pomoc, szanowni państwo, wygląda m.in. tak: Biała Podlaska - zero, Drelów - zero, Janów Podlaski - zero, Kodeń - zero, Konstantynów - zero, Międzyrzec Podlaski - zero, Rokitno - zero, Rososz - zero, Sosnówka - zero, Terespol - zero, Tuczna - zero, Wisznice - zero, Zalesie - zero, Biała Podlaska - zero, Aleksandrów - zero, Biłgoraj - zero, gmina Biłgoraj - zero, Józefów - zero, Potok Górny - zero, Tarnogród - zero, Terespol - zero, Dorohusk - zero, Dubienka - zero, Kamień - zero, Rejowiec - zero, Rejowiec Fabryczny - zero, Ruda Huta - zero, Siedliszcze - zero, Wojsławice - zero, Żmudź - zero, Dołhobyczów - zero, Horodło - zero, Hrubieszów - zero, Mircze - zero, Uchanie - zero, gmina Batorz - zero, Dzwola - zero, Modliborzyce - zero, Fajsławice - zero, Gorzków - zero, Izbica - zero, Krasiczyn - zero, Krasnystaw - zero, Łopiennik Górny - zero, Sienica Różana - zero, Annopol - zero, Dzierzkowice - zero, miasto Kraśnik - zero, gmina Kraśnik - zero, Abramów - zero, Kamionka - zero, Lubartów - zero, gmina Lubartów - zero, Michów - zero, gmina Ostrówek - zero, Uścimów - zero, Borzechów - zero, Bychawa - zero, Garbów - zero, Głusk - zero, Jabłonna - zero, Konopnice - zero, Krzczonów - zero, Niemce - zero, Strzyżewice - zero, Wólka - zero, Zakrzew - zero. I jeszcze ponad 100 gmin, w tym gmina Lublin i gmina Puławy. To jest po prostu skandal. Dzielicie ludzi na gorszych i lepszych. Dziękuję. Bardzo proszę pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych miał służyć wszystkim samorządom. Takie było jego podstawowe założenie. Natomiast PiS, rozdzielając pieniądze, przyznał je tylko swoim, bo chciał ukarać samorządowców nieposłusznych. Jednak nie ukarał samorządowców, tylko ukarał mieszkańców tych samorządów. 0 zł na Lubelszczyźnie dostały m.in.: Lublin, gmina Cyców, gmina Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, Krzywda, miasto Łuków, gmina Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica, Końskowola, Markuszów, miasto Puławy, gmina Puławy, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń, Nowodwór, Stężyca, Piaski, Rybczewice, Trawniki, Bełżec, Jarczów, Susiec, miasto Tomaszów Lubelski, gminy Tyszowce, Orchówek, Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, miasto Włodawa, gminy Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Skierbieszów, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Zamość. Obiecujemy, że żaden z samorządowców pokrzywdzonych przez PiS nie zostanie z tą krzywdą sam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan premier Mateusz Morawiecki upodobał sobie zera. Chyba kolekcjonuje rząd składających się z zer. Jedno zero wszyscy już znamy, ale skąd umiłowanie pana premiera do zera dla Polek i Polaków zamieszkujących polskie wsie, miasta i miasteczka? Tego nie wiemy. Dlaczego pan, panie premierze, tak nieuczciwie traktuje polskie samorządy terytorialne? W województwie lubuskim: powiat zielonogórski - zero.

Babimost - zero, Bytom Odrzański - zero, Cybinka - zero, Dąbie - zero, Deszczno - zero, Gozdnica - zero, Jasień - zero, Kargowa - zero, Kolsko - zero, Kostrzyn nad Odrą - zero, Kożuchów - zero, Krosno Odrzańskie - zero, Krzeszyce - zero, Małomice - zero, Maszewo - zero, gmina miejska Nowa Sól - zero, gmina o statusie wiejskim Nowa Sól - zero, Nowogród Bobrzański - zero, Ośno Lubuskie - zero, Przytoczna - zero, Santok - zero, Szczaniec - zero, Słubice - także zero, Strzelce Krajeńskie - zero, Szprotawa - zero, Świdnica - zero, Świebodzin - zero, Torzym - zero, Trzebiechów - zero, Trzebiel - zero, Tuplice - zero, Wschowa - zero, Wymiarki - zero, Zabór - zero, Zwierzyń - zero, Zielona Góra - także zero. Panie Premierze! W lubuskich gminach żyją tacy sami Polacy jak w innych miejscach naszego pięknego kraju, ale niestety pan nie był uprzejmy przyjąć merytorycznych kryteriów, na podstawie których dzieliłby pan tenże rządowy fundusz inicjatyw lokalnych. Pan przyjął proste i jedyne chyba kryterium, które jest pan w stanie zrozumieć i pojąć: kryterium przynależności do danej partii politycznej. Oczywiście nagradza pan tylko koleżanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Dla tych lubuskich gmin środki finansowe się znalazły, dla innych gmin, rządzonych przez wiele lat przez sprawnych lokalnych liderów, menadżerów te pieniądze się nie znalazły. Panie Premierze! Czas skończyć. Bardzo proszę, pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 20. rok pełnię służbę w polskim parlamencie, ale po raz pierwszy wychodzę na trybunę w trybie oświadczeń poselskich. Powód naprawdę jest ważny.

W tym wypadku ten podział dotyczy gmin. Jak wygląda sytuacja w województwie łódzkim? Miasto Łódź otrzymuje zero dotacji, gmina Drzewica - zero dotacji, gmina Mniszków - zero dotacji, gmina Opoczno - zero dotacji, gmina Poświętne - zero dotacji, gmina Sławno - zero dotacji, gmina Żarnów - zero dotacji, gmina Dobryszyce - zero dotacji, gmina Gidle - zero dotacji, gmina Kamieńsk - zero dotacji, gmina Radomsko - zero dotacji, gmina Cielądz - zero dotacji, gmina Regnów - zero dotacji, gmina Sadkowice - zero dotacji, gmina Bolimów - zero dotacji, gmina Kowiesy - zero dotacji, gmina Godzianów - zero dotacji, gmina Maków - zero dotacji, gmina Nowy Kawęczyn - zero dotacji, gmina Słupia - zero dotacji, gmina Inowłódz - zero dotacji, gmina Lubochnia - zero dotacji, gmina Rzeczyca - zero dotacji, gmina Grabica - zero dotacji, gmina Łęki Szlacheckie - zero dotacji, gmina Moszczenica - zero dotacji, gmina Kluki - zero dotacji, gmina Drużbice - zero dotacji, gmina Ujazd - zero dotacji, gmina Żelechlinek - zero dotacji. Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Miał być rządowy fundusz inwestycji lokalnych, a jest rządowy fundusz dla działaczy PiS i przez działaczy PiS organizowany za publiczne pieniądze. Zresztą to przy okazji poważnej debaty na temat budżetu pokazuje w jasny sposób, jak PiS próbuje budować państwo PiS za nasze, publiczne pieniądze. Nie tak dawno premier Morawiecki powiedział, że ten fundusz inwestycji to będą pieniądze na najbardziej palące problemy. Więc jak czytamy, ile tych gmin i miast nie dostało, to okazuje się, że premier w ogóle nie ma żadnej wiedzy, co to są palące problemy i na co te publiczne pieniądze powinny pójść. Pan minister Grabarczyk przed momentem wymienił część województwa łódzkiego, to ja pozwolę sobie wymienić drugą część tych wszystkich miast i powiatów, które nie dostały ani złotówki według tego podziału. Rozpocznę od powiatu kutnowskiego: Bedlno, Krośniewice, Kutno, Nowe Ostrowy, Oporów, Żychlina, Łanięta, wszystkie te miasta - zero. Tam PiS też nie rządzi, dlatego jest zero. Powiat łęczycki: Daszyna, Grabów, Piątek i Łęczyca - zero. Powiat pabianicki: Ksawerów, Pabianice - zero.

A swoją drogą nie tak dawno radni dali nawet odznaczenie dla prezydenta Dudy w Wieluniu. Też nie dostali, bo tam PiS nie rządzi. Powiat wieruszowski: Bolesławiec, Galewice i Wieruszów - zero. Powiat zduńskowolski: gmina, miasto Szadek, gminy Zapolice, Zduńska Wola - zero. Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Parzęczew i Stryków - równe zero. I powiat sieradzki: Błaszki, Goszczanów, miasto Warta i Wróblew - zero. Dlatego złożyliśmy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo proszę, pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska.

Pan poseł Marek Sowa, a potem przygotowuje się pan poseł Aleksander Miszalski. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Trzeba to wprost powiedzieć: Mateusz Morawiecki jest twarzą największego politycznego oszustwa w historii 30 lat polskiej samorządności. W Małopolsce przyznał takie dotacje. Małopolska zachodnia: powiat chrzanowski - 0 zł, Chrzanów - zero, Libiąż - zero, Trzebinia - zero, Babice - zero, powiat myślenicki - zero. Gminy: Lubień - zero, Raciechowice - zero, Siepraw - zero, Wiśniowa - zero. Powiat oświęcimski - zero, miasto Oświęcim - zero, gmina Oświęcim - zero, Chełmek - zero, Kęty - zero, Osiek - zero, Polanka Wielka - zero, Przeciszów - zero. Powiat suski: Sucha Beskidzka - zero, Maków Podhalański - zero, Budzów - zero, Stryszawa - zero, Zembrzyce - zero. Powiat wadowicki: Andrychów - zero, Brzeźnica - zero, Tomice - zero, Wieprz - zero. Podhale i Sądecczyzna: powiat gorlicki - zero, miasto Gorlice - zero. Gminy: Biecz - zero, Gorlice - zero, Lipinki - zero, Moszczenica - zero, Sękowa - zero. Powiat limanowski, miasto Limanowa - zero, Jodłownik - zero, Kamienica - zero. Gmina Mszana Dolna - zero, Niedźwiedź - zero. Powiat nowosądecki: Muszyna - zero, Chełmiec - zero, Gródek nad Dunajcem - zero, Grybów - zero, Korzenna - zero, Łabowa - zero, Podegrodzie - zero. Powiat nowotarski: miasto Nowy Targ - zero, powiat nowotarski - zero. Powiat tatrzański: Biały Dunajec - zero, Bukowina Tatrzańska - zero, Kościelisko - zero. Szanowni Państwo! Mateusz Morawiecki w Małopolsce wręczył 92 zerowe czeki (Dzwonek) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziękuję, panie pośle. Przygotowuje się pani poseł Aleksandra Gajewska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rządzie, którego nie ma! Zrobiliście program bez kryteriów, bez merytoryki, bez oceny wniosków, program sami swoi. Chcieliście oszukać samorządowców, ale tak naprawdę oszukaliście mieszkańców - i to często mieszkańców, którzy na was w Małopolsce bardzo często głosowali. Tam, gdzie PiS składał wnioski, PiS rządzi, 89 wniosków przyznanych na 89 złożonych. Tam, gdzie pozostali rządzą, 18 na 112, czyli 15%. No i żeby nie być gołosłownym: miasto Bochnia - zero, Rzezawa - zero, Żegocina - zero, Drwinia - zero, gmina Bochnia- zero, Iwkowa - zero, Czchów - zero, miasto Brzesko - zero, Radgoszcz - zero, Bolesław - zero, Dąbrowa Tarnowska - zero, Radziemice - zero, Koniusza, Pałecznica, Koszyce, wszystko w powiecie proszowickim - zero, Tarków - zero, Gromnik - zero, Wierzchosławice - zero, Lisia Góra - zero, Skrzyszów, Radłów - zero, Biskupice, Gdów, Wieliczka, Niepołomice - zero, Michałowice - zero, Zabierzów - zero, Zielonki - zero, Iwanowice, Sułoszowa - zero, Wawrzeńczyce - zero, Skała - zero, Świątniki Górne, Liszki - zero, Gołcza, Książ Wielki, Miechów - zero, Wolbrom - zero, Bukowno - też zero, Kraków - oczywiście zero. Mieszkańcy Małopolski wam tego nie zapomną. Bardzo proszę, pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Przygotowuje się pani poseł Katarzyna Piekarska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyznam, że nie przypominam sobie czasu, kiedy ostatnio PiS wygrał w Warszawie wybory. I za to PiS nie lubi Warszawy, nie lubi warszawianek, nie lubi warszawiaków, nie lubi prezydenta Trzaskowskiego. Nie lubi, wychodzi na to również, mieszkańców Mazowsza, bo ich również postanowił pominąć w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. I tak: gmina Leoncin dostała zero, gmina Nasielsk - zero, gmina Pomiechówek - zero, gmina Zakroczym - zero, Nowy Dwór Mazowiecki - zero. Powiat ostrołęcki - zero, gmina Baranowo - zero, gmina Goworowo - zero, gmina Kadzidło - zero, gmina Lelis - zero, gmina Rzekuń - zero, Ostrołęka - zero, gmina Andrzejewo - zero, gmina Brok - zero, Małkinia Górna - zero, Szulborze Wielkie - również zero, Wąsewo - zero, Celestynów - zero, Karczew - zero, Kołbiel - zero, Osieck - zero, Sobienie-Jeziory - zero. Powiat piaseczyński - zero, gmina Góra Kalwaria - zero, Konstancin-Jeziorna - zero, Lesznowola - zero, gmina Piaseczno - zero, Prażmów - zero, Płock - zero. Cały powiat płocki - zero, gmina Bielsk - zero, gmina Bodzanów - zero, gmina Łąck - zero, gmina Nowy Duninów - zero, gmina Radzanowo - zero, gmina Słubice - zero, gmina Słupno - zero, gmina Staroźreby - zero, Baboszewo - zero, Dzierzążnia - zero, Joniec - również zero, gmina Naruszewo, gmina Nowe Miasto - zero, gmina Płońsk - zero, Raciąż - zero, Suchocin - zero, gmina Załuski - zero, Płońsk - zero. Powiat pruszkowski - zero, gmina Brwinów - zero, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków - zero. Powiat przasnyski - zero, gmina Chorzele - zero, Czernice Borowe - również zero, Jednorożec - zero, Krasne - zero, Przasnysz - zero, Borkowice - zero, Gielniów - zero, Klwów - zero, Potworów - zero, Przysucha - zero, Rusinów - zaskoczę państwa - zero, Wieniawa - zero. Powiat pułtuski, gmina Obryte - zero, gmina Pokrzywnica - zero, gmina Zatory - zero, gmina Jastrzębia - zero, gmina Kowala - zero, gmina Pionki - zero, gmina Przytyk - zero i Skaryszew - zero. Ale to nie koniec, będą kontynuowały to moje koleżanki. Przygotowuje się pani poseł Katarzyna Lubnauer. Szanowna Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy!

I to jest tak: gmina Białobrzegi, gmina Promna, gmina Radzanów, powiat ciechanowski, Ciechanów, i to mimo siedmiu wniosków, dostały zero. Gmina Glinojeck, gmina Gołymin-Ośrodek, gmina Ojrzeń, gmina Opinogóra Górna, gmina Sońsk. Garwolin, Parysów, Pilawa, Sobolew, Wilga, Łaskarzew. Powiat gostyniński, gmina Pacyna, gmina Sanniki, gmina Szczawin Kościelny. Powiat grodziski, gmina Baranów, gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna. Powiat grójecki, gmina Chynów, gmina Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Warka. Głowaczów, Gniewoszów, gmina Grabów nad Pilicą, gmina Magnuszew, gmina Sieciechów. Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, gmina Stara Kornica. Powiat makowski, gmina Czerwonka, gmina Karniewo, gmina Płoniawy-Bramura, gmina Różan, Rzewnie, Szelków. Dębe Wielkie, gmina Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica. To jest naprawdę skandal. Dalej: gmina Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo, Mława, gmina Czosnów. Te wszystkie gminy, które wymieniłam, to są gminy na Mazowszu, które dostały zero środków. I to jest absolutny skandal, bo jak mówił czy mówiła pewna pani premier: te pieniądze tym obywatelom, którzy tam mieszkają, się po prostu należały, a dostali zero. Dziękuję, pani poseł. Przygotowuje się pan poseł Mirosław Suchoń. Jak, proszę państwa, PiS myśli o pieniądzach publicznych: „Jest to pewna schizofrenia ze strony opozycyjnych samorządowców, którzy regularnie krytykują rząd, plują na niego, a później wyciągają do tego rządu ręce po pieniądze” Oni nie dzielą pieniędzy, które sami zarobili, tylko te, które podatnicy mieszkający w całej Polsce wpłacili do budżetu państwa.

Proszę państwa, pięć największych miast Polski: Warszawa - 1790 tys. mieszkańców, Kraków - 780 tys. mieszkańców, Łódź - 677 tys. mieszkańców, Wrocław - 643 tys. mieszkańców, Poznań - 534 tys. mieszkańców, w sumie prawie 4,5 mln mieszkańców.

Dziękuję bardzo. Przygotowuje się pani poseł Joanna Frydrych. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Fundusz inwestycji lokalnych to miał być taki solidarnościowy wehikuł. Solidarnościowy wehikuł, który w tym trudnym czasie epidemii pozwoli gospodarkom naszych małych, większych ojczyzn złagodzić skutki epidemii i odbudować naszą siłę. Niestety PiS postanowił podzielić Polaków na lepszych i gorszych, na tych, którzy otrzymają wsparcie, i na tych, którzy tego wsparcia nie otrzymają. I do tego użył wyłącznie kryterium politycznego, żadnych merytorycznych kryteriów. Niestety także na Podbeskidziu, Śląsku Cieszyńskim, Żywiecczyźnie i Ziemi Pszczyńskiej w wielu miejscach to było zero. I tak w województwie opolskim, które tego wsparcia potrzebuje w sposób absolutnie kluczowy: Opole, największe miasto województwa, miasto wojewódzkie - 0 zł, powiat brzeski, Brzeg - zero, Olszanka - zero, Skarbimierz - zero, powiat głubczycki, Głubczyce - zero, Kietrz - zero, Branice - zero, powiat kędzierzyńsko-kozielski, Kędzierzyn-Koźle - zero, Cisek - zero, Polska Cerkiew - zero, Reńska Wieś - zero, powiat kluczborski, Kluczbork - zero, powiat krapkowicki, Krapkowice - zero, Gogolin - zero, Zdzieszowice - zero, Walce - zero, Świerczów w powiecie namysłowskim - zero, powiat nyski, Głuchołazy - zero, Korfantów - zero, Nysa - zero, Otmuchów - zero, Kamiennik - zero, Łambinowice - zero, Pakosławice - zero, powiat oleski, Olesno - zero, Gorzów Śląski - zero, Olesno - zero, Praszka - zero, Radłów - zero, powiat opolski ziemski, Chrząstowice - zero, Dąbrowa - zero, Łubniany - zero, Murów - zero, Tarnów Opolski - zero, Turawa - zero, w powiecie prudnickim Lubrza - zero, powiat strzelecki, Strzelce Opolskie - zero, Kolonowskie - zero, Leśnica - zero, Ujazd - zero, Zawadzkie - zero, Izbicko - zero, Jemielnica - zero. Cała Polska musi dziś usłyszeć, że zero to prawdziwy program rządu dla Polek i Polaków. Te gminy, ci mieszkańcy, którzy zostali pokrzywdzeni, muszą dzisiaj usłyszeć, jak bardzo niesprawiedliwy jest podział tych środków i jak bardzo daleko od solidarności, która powinna kierować działaniami rządu, stoi dzisiaj rząd PiS. Dziękuję, panie pośle. Przygotowuje się pan poseł Robert Tyszkiewicz, także Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wydawanie środków publicznych powinno odbywać się w sposób transparentny, z określeniem jasnych kryteriów i jasnych reguł. Przyznawanie tych środków według linii politycznej to jawna dyskryminacja mieszkańców miast i gmin, które zostały tych środków pozbawione. A dlaczego? Bo ich włodarze nie są związani z PiS. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program zero+ dla niezależnych samorządów, a jego beneficjentami w województwie podkarpackim są: Ustrzyki Dolne - zero, Domaradz - zero, Haczów - zero, Nozdrzec - zero, Brzostek - zero, Dębica - zero, Pilzno - zero, Czarna - zero, Żyraków - zero, Jarosław - zero, Pawłosiów - zero. Roźwienica - zero, Wiązownica - zero, Cmolas - zero, Raniżów - zero, Dukla - zero, Iwonicz-Zdrój - zero, Krosno - zero, Korczyna - zero, Wojaszówka - zero, Cisna - zero, Cieszanów - zero, Oleszyce - zero, Grodzisko Dolne - zero, Łańcut - zero, Radomyśl Wielki - zero, Borowa - zero, Czermin - zero, Gawłuszowice - zero, Padew Narodowa - zero, Wadowice Górne - zero, Nisko - zero, Przemyśl - zero, Bircza - zero, Przeworsk - zero, Kańczuga - zero, Sieniawa - zero, Jawornik Polski - zero, Ropczyce - zero, Rzeszów - zero, Błażowa - zero, Dynów - zero, Sokołów Małopolski - zero, Hyżne - zero, Krasne - zero, Świlcza - zero, Zarszyn - zero, Strzyżów - zero, Wiśniowa - zero, Gorzyce - zero i Grębów - zero. Tak PiS dzieli samorządy, dzieli Polki i Polaków. Ale polskie przysłowia są bardzo mądre i ponadczasowe. Przytoczę jedno: dopóty dzban wodę nosi, dopóki ucho się nie urwie. Absolutna władza PiS-u też wkrótce się skończy. Przygotowuje się pani poseł Agnieszka Pomaska. Wysoka Izbo! Szczególnie bolą zawiedzione obietnice. Województwo podlaskie, Polska wschodnia miała być za rządów PiS krainą miodem i mlekiem płynącą, a spłynęła wielkim politycznym kłamstwem, wielkim politycznym oszustwem. Myśmy zadali sobie trud i policzyliśmy, ilu mieszkańców Podlasia zostało oszukanych przez rząd PiS-u i pozbawionych pieniędzy na oczekiwane przez nich inwestycje. Na 1100 tys. mieszkańców tego niewielkiego regionu 670 tys. osób, 670 tys. ludzi zostało pozbawionych pieniędzy z tytułu programu inwestycji lokalnych. Miał być program inwestycji lokalnych, a jest program inwestycji partyjnych, których jedynym wyznacznikiem, jedynym kryterium jest legitymacja PiS-u w kieszeni działaczy samorządowych. Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o miasta, wspólnoty, powiaty, gminy województwa podlaskiego, które zostały pozbawione środków, to lista przedstawia się naprawdę zatrważająco. Zacznijmy od największych miast, miast na prawach powiatu, których w regionie jest trzy: Białystok - zero, Suwałki - zero. Jeżeli chodzi o powiaty, które wnioskowały o środki na inwestycje: powiat augustowski - zero, powiat bielski - zero, powiat hajnowski - zero, powiat moniecki - zero, powiat sejneński - zero, powiat siemiatycki - zero, powiat zambrowski - zero. W powiecie augustowskim: miasto Augustów - zero, miasto Lipsk - zero. W powiecie białostockim: Choroszcz - zero, Michałowo - zero, Suraż - zero, Zabłudów - zero, gmina Dobrzyniewo Duże - zero, gmina Gródek - zero, gmina Juchnowiec Kościelny - zero, gmina Zawady - zero. W powiecie bielskim: Bielsk Podlaski - zero, Brańsk - zero, gmina Bielsk Podlaski - zero, gmina Rudka - zero, gmina Wyszki - zero. W powiecie grajewskim: Rajgród - zero, Szczuczyn - zero. W powiecie hajnowskim: Hajnówka - zero, Kleszczele - zero, gmina Czyżew - zero, gmina Dubicze Cerkiewne - zero, gmina Narew - zero, gmina Narewka - również zero. W powiecie kolneńskim: gmina Mały Płock - zero, gmina Turośl - zero. W powiecie łomżyńskim: gmina Łomża - zero, gmina Miastkowo - zero, gmina Piątnica - zero, gmina Zbójna - zero. W powiecie monieckim: Knyszyn - zero, Mońki - zero, gmina Jasionówka - zero, gmina Krypno - zero zł na inwestycje. W powiecie sejneńskim: Sejny - zero, gmina Puńsk, zamieszkała przez mniejszość litewską, a jakże (Dzwonek) - również zero. W powiecie siemiatyckim: Siemiatycze - zero, gmina Siemiatycze - zero, gmina Mielnik - zero, gmina Milejczyce - zero, gmina Nurzec-Stacja - zero. W powiecie sokólskim: Suchowola - zero, słynna na całą Polskę gmina Korycin, gdzie sery korycińskie się produkuje - również zero, bo nie rządzi tam PiS. W powiecie suwalskim: gmina Filipów - zero, gmina Rutka-Tartak - zero, gmina Szypliszki - zero. W powiecie wysokomazowieckim: gmina Klukowo - zero, gmina Kulesze Kościelne - również zero. W powiecie zambrowskim: miasto Zambrów - zero, gmina Rutki - zero. Taki jest obraz inwestycji lokalnych oferowanych przez PiS dla mieszkańców województwa podlaskiego. Nigdy tego nie zapomnimy i twardo to na Podlasiu rozliczymy. Panie i Panowie Posłowie! Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej już w sierpniu br. ostrzegali, że kryteria przyznawania środków z funduszu inwestycji lokalnych są niejasne. W tej sprawie skierowaliśmy m.in. interpelację. I co odpisał wiceminister Robert Nowicki? Odpisał, że nie przewidziano pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia dyspozycji wypłat środków, bo przygotowanie odpowiedzi stanowiłoby znaczny wysiłek organizacyjny. Jak patrzymy na aktywność przedstawicieli rządu w uprawianiu propagandy za publiczne środki, to ja się pytam albo w zasadzie apeluję: Weźcie się do roboty. Weźcie się do roboty, a nie mówcie, że nie macie czasu na uzasadnienie wniosków. To po pierwsze. Po drugie, chciałam zwrócić uwagę, że to nie są jakieś wirtualne pieniądze i wirtualne inwestycje. To nie jest odebranie czegoś fikcyjnego gdzieś w przestrzeni, tylko to są konkretne inwestycje, to są konkretne środki, w konkretnych gminach, miastach i powiatach. Dla przykładu w gminie Potęgowo pieniędzy nie będzie na budowę żłobka i termomodernizację szkoły podstawowej. To są pieniądze odebrane gminie Potęgowo przez obecny rząd.

Panie ministrze, pan kłamał, okłamywał pan mieszkańców województwa pomorskiego i Potęgowa. W Malborku nie będzie modernizacji ul. Nowowiejskiego. W Nowym Dworze nie będzie ścieżki rowerowej, nie będzie remontu dróg. W Pucku nie będzie przebudowy ul. Nowy Świat, puckiego centrum kultury, budowy nowej mariny czy rozbudowy kanalizacji. W mieście Gdańsk nie będzie pieniędzy na objazd Bramy Nizinnej, bezkolizyjny przejazd na Orunię czy wał przeciwpowodziowy. W Słupsku nie będzie rewitalizacji Starego Rynku, budowy mieszkań komunalnych.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Król, Koalicja Obywatelska. Przygotowuje się pani poseł Mirosława Nykiel. Pani Marszałek! Przypomnę, że z tego miejsca Beata Szydło mówiła, że aby wystarczyło dla wszystkich, wystarczy nie kraść. Sprawdzimy, czy wystarczyło dla wszystkich.

Dodam, że Chorzów, Imielin i powiat bieruńsko-lędziński - miasto, gmina i powiat - to okręg wyborczy Mateusza Morawieckiego. Startował z tego okręgu do Sejmu i zdradził swoich wyborców. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przygotowuje się pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

To oni nie będą mieć lepszych obiektów oświatowych, dróg, połączeń kolejowych, lepszych przedszkoli, obiektów służby zdrowia. Ten partyjny podział to hańba i blamaż PiS-u. Tak naprawdę podzieliliście pieniądze Polek i Polaków według partyjnego poważania. Teraz wymienię te hojnie obdarowane miejscowości. Bielsko-Biała - zero, Czechowice-Dziedzice - zero, Żywiec - zero, Cieszyn - zero, Jaworze - zero, Szczyrk - zero, Goczałkowice-Zdrój - zero, Kobiór - zero, Miedźna - zero, Pawłowice - zero, Dębowiec - zero, Ustroń - zero, Wisła - zero, Zebrzydowice - zero, Lipowa - zero, Łękawica - zero, Milówka - zero, Blachownia - zero, Dąbrowa Zielona - zero, Kamienica Polska - zero, Kłomnice - zero, Koniecpol - zero, Konopiska - zero, Mstów - zero, Mykanów - zero, Przyrów - zero, Starcza - zero, Kłobuck - zero, Krzepice - zero, Lipie - zero, Miedźno - zero, Wręczyca Wielka - zero. Wiecie, jakiego wyniku powinien spodziewać się PiS w najbliższych wyborach w tych miejscowościach? zero. Przygotowuje się pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ostatnimi czasy zaczęło być modne rządowe. Mamy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który ani nie jest funduszem, ani nie jest rządowy. Czyli rząd rozdaje coś, co nawet nie jest jego. Wprawdzie pan premier jest dysponentem tych środków, ale zabiera je z funduszu przeciwdziałania skutkom COVID-19, a ten fundusz jest jeszcze zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który pieniądze zaciąga na ten cel częściowo z budżetu państwa, z emisji obligacji i z funduszy europejskich i innych zagranicznych. Tak że ani rządowy, ani premiera. Rozdaje się nie swoje, a niektórym nie daje się nic. Po pierwsze, żadnych czytelnych kryteriów, i to jest najważniejszy błąd, ani żadnych procedur. To jest niezgodne ze świętą zasadą finansów publicznych, gdzie dyspozycja musi być odpowiednia, przejrzysta i równa dla wszystkich.

Nie dostał powiat wodzisławski, który też nie jest ulubieńcem PiS-u, a w powiecie wodzisławskim podobnie nie kochane Marklowice. Z powiatu rybnickiego Jejkowice, a także Rudnik, który miał m.in. projekty na udostępnienie niepełnosprawnym obiektów, które służą im pomocą. Panie Premierze! Zwróciłam się do pana i z interpelacją, i z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Niech pan raz ma odwagę i odpowie w tym trybie tym wszystkim gminom, powiatom, które dostały zero, dlaczego i uzasadni tak, jak należy to zrobić, zgodnie z zasadami finansów publicznych, z szacunkiem dla pieniędzy nie pańskich, bo to są pieniądze Polaków, które - tak jak już wspomniano - im się należą. Ale należy im się przede wszystkim rozliczenie i wytłumaczenie takiego trybu. To nie jest pana folwark [[Dzwonek]] i nie pana pieniądze. Przygotowuje się pan poseł Jacek Protas. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo! Otóż wydawałoby się, że województwo świętokrzyskie będzie bardziej łaskawie potraktowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak rzeczywistość stała się bardziej brutalna, ponieważ ok. połowy gmin województwa świętokrzyskiego wsparcia z funduszu inwestycji lokalnych po prostu nie otrzymało. Szanowni Państwo!

Powiat kazimierski: Czarnocin, Kazimierza Wielka, Chęciny - zero. Powiat kielecki: Chęciny, Daleszyce, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Sitkówka, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Łagów, Łopuszno - zero. Powiat konecki: Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Słupia - zero. Powiat opatowski: Opatów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice - zero. Powiat ostrowiecki: Bodzechów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów - zero. Powiat pińczowski: Kije, Michałów, Złota - zero.

Powiat staszowski: Osiek, Połaniec, Łubnice - zero. Powiat włoszczowski: Krasocin, Moskorzew, Secemin - zero. Łącznie 55 gmin - zero.

Wielka szkoda, bo rzeczywiście okazuje się, że największe ośrodki, nawet miasta prezydenckie tak jak Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski czy Skarżysko-Kamienna, zostały zupełnie pominięte. Jakże jest to żenujące, że jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, ówczesny wojewoda, tak naprawdę mówi wprost o tym, że to ona przyczyniła się do tego, że te środki trafiły do tej, a nie innej gminy. A więc jest to przynależność, kryterium jest tylko polityczne, partyjne czy też terytorialne. Tak być nie powinno. Dlatego też liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwości się opamięta i weźmie pod uwagę to, że skrzywdziło mieszkańców ponad połowy gmin województwa świętokrzyskiego, i te pieniądze kiedyś przyjdą. Póki co w połowie mamy zero.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan premier Mateusz Morawiecki szumnie zapowiadał, że dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych skończy się podział Polski na Polskę A i Polskę B, ale zapomniał dodać, że zacznie się podział Polski na Polskę PiS i całą resztę, na lepszy i gorszy sort. Zobaczmy, jak to wygląda, porównując województwa. Region podkarpacki - 452 mln zł z tego funduszu, warmińsko-mazurski - 138 mln. Podobna powierzchnia, podobna populacja, podobny poziom rozwoju. Jak to wygląda na osobę? Czyżbyśmy w naszym regionie byli tym gorszym sortem? Przez to 0 zł z funduszu dostały miasta prezydenckie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, powiaty: lidzbarski, giżycki, iławski, mrągowski, olsztyński, szczycieński - 0 zł, gminy: Frombork, Płoskinia, Braniewo, Wilczęta, Płośnica, Pasłęk, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Rychliki - 0 zł, Prostki, Stare Juchy, Ełk, Gołdap, Banie Mazurskie, Giżycko, Ryn, Kruklanki, Miłki i Wydminy - 0 zł, Iława, Kisielice, Susz, Reszel, Orneta, Lubomino, Mikołajki - 0 zł, Sorkwity, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec - 0 zł, Olecko, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda - 0 zł, Ostróda, Miłomłyn, Morąg, Łukta, Biała Piska, Orzysz - 0 zł, Szczytno, Wielbark, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Budry - 0 zł.

Tak wygląda polityka równomiernego rozwoju, tak wygląda polityka wyrównywania szans między regionami, powiatami i gminami w wykonaniu PiS. Puste słowa i kłamstwa premiera, który już wiele razy przez sąd został skazany za kłamstwa. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przygotowuje się pan poseł Adam Szłapka. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Fundusz inwestycji lokalnych jest finansowany de facto przez wszystkich Polaków. To nie jest fundusz wyborców, funkcjonariuszy PiS, a tak został niestety potraktowany, także w Wielkopolsce. Połowa samorządów w Wielkopolsce nie otrzymała ani złotówki na inwestycje. Powiat gnieźnieński: Gniezno, Kiszkowo, Mieleszyn, Niechanowo, Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo - zero, Borek Wielkopolski, Pogorzela - zero, Granowo, Kamieniec, Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo - zero, Jaraczewo, Kotlin, Jarocin, Żerków - zero. Powiat kaliski: Blizanów, Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin, Stawiszyn - zero, Bralin, Chodów, Kościelec, Osiek Mały, Przetycz - zero. Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Rychwał, Ślesin - zero. Powiat międzychodzki - zero: Międzychód, Sieraków - zero. Powiat obornicki - zero: Ryczywół, Oborniki - zero, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice - zero. Powiat ostrzeszowski - zero: Grabów nad Prosną, Ostrzeszów - zero, Piła - zero, Białośliwie, Kaczory, Ujście, Wyrzysk, Wysoka - zero, Obrzycko, Duszniki - zero, Ostroróg, Szamotuły, Wronki - zero, Zaniemyśl, Środa Wielkopolska - zero. Powiat śremski: Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem - zero, Budzew, Kawęczyn, Przykona, Tuliszków - zero. Powiat wągrowiecki - zero: Wągrowiec, Wapno, Gołańcz, Skoki - zero. Powiat wolsztyński - zero: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn - zero. Powiat wrzesiński - zero: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla - zero, Zakrzewo Krajenka, Okonek - zero. I oczywiście, proszę państwa, stolica Wielkopolski: Poznań - również zero. Trzeba zapamiętać to nie tylko premierowi i rządowi, trzeba zapamiętać to również wszystkim posłom PiS i całej Zjednoczonej Prawicy, bo nie ujęli się za tymi miejscowościami z czysto politycznego powodu: dlatego że tam nie wygrywają. Pan Artur Łącki przygotowuje się. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jedną z cech opisujących państwa, które mają problem z demokracją, z praworządnością, instytucjami, silnymi instytucjami, jest zatarcie granicy między rządzącą partią a państwem. Dla waszych aparatczyków, dla waszych kacyków państwo to partia, a partia to państwo. Wam władza nie jest potrzebna do tego, żeby pomagać obywatelom, żeby rozwiązywać problemy obywateli, tylko po to, żeby załatwiać własne interesy i tę władzę umacniać, żeby niszczyć instytucje i wyciągać zasoby państwa tylko po to, żeby realizować partyjne interesy. I dokładnie o tym świadczy to wszystko, co zdarzyło się z funduszem inwestycji lokalnych. Wykorzystujecie pieniądze, które są pieniędzmi podatników, obywateli tylko po to, żeby wspierać swoich i karać tych, którzy odważyli się nie zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. To jest skandal, to jest niszczenie państwa i za to wszyscy odpowiecie. A oto gminy w Wielkopolsce, które zostały przez was ukarane za to, że nie są gminami PiS-owskimi: Poznań - zero, Puszczykowo - zero, Czerwonak - zero, Komorniki - zero, Rokietnica - zero, Tarnowo Podgórne - zero, Buk - zero, Kórnik - zero, Mosina - zero, Murowana Goślina - zero, Stęszew - zero, Czempiń - zero, Krzywiń - zero i tak można wymieniać i wymieniać kolejne gminy. Niszczycie Polskę i każecie obywateli za to, że uczestniczą w normalnych, demokratycznych wyborach. Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Łącki. Przygotowuje się pani poseł Wanda Nowicka, Lewica.

Dzielić zaczął nas już wtedy, kiedy krzyczał, że my stoimy tam, gdzie ZOMO, a oni gdzie indziej. Ale skąd to wiedział, skoro sam spał do południa? Dzieli na tych, którzy odpowiadają za swoje przestępstwa, i na tych, którzy nie muszą, którym można wybaczyć, bo zgrzeszyli, bo któż nie ma pokus. Dzielą na tych, którzy dostają gazem po oczach, pałą w łeb i mandat do zapłaty, i na tych, którzy bezkarnie poniewierają kobiety w strajkach, łamią im ręce i biją pałkami. Dzieli przedsiębiorców na tych, którzy dostają jakąś tam pomoc z dziurawych durszlaków COVID-owych, na tych, którzy mieli nieszczęście mieć inny REGON, więc nie dostaną nic. A teraz zaczęli jeszcze dzielić samorządy na te, które dostaną pomoc z rządowego funduszu tylko dlatego, że głosowały, jak chciał prezes, i na te, które nie dostaną, bo źle głosowały.

Wyjaśnimy, kto i według jakich kryteriów podzielił [[Dzwonek]] te pieniądze z funduszu inwestycji lokalnych, trwa nasza poselska kontrola w KPRM-ie, jutro złożymy w Najwyższej Izbie Kontroli wniosek o przeprowadzenie kompleksowej kontroli. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Dziś przypada 98. rocznica zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza. 16 grudnia 1922 r. pierwszy prezydent Rzeczypospolitej został zastrzelony przez prawicowego fanatyka kilka dni po objęciu urzędu. Był to efekt kampanii, jaką przeciwko Narutowiczowi wszczęła nacjonalistyczna prawica. Zamach na prezydenta Narutowicza poprzedzony był szowinistyczną nagonką. Media i politycy związani z endecją, z Narodową Demokracją zarzucali mu, że był ateistą, używali antysemickiej retoryki, otwarcie wzywali do tego, żeby się go pozbyć. Dzisiaj widzimy wszyscy, że polityka oparta na ksenofobii i nienawiści, która doprowadziła do jego śmierci, powróciła. Obecnie otacza nas podobna atmosfera, słyszymy tę samą retorykę i słowa o wrogach Polski, o obcej agenturze, a zindoktrynowani przez nieodpowiedzialnych polityków młodzi ludzie noszą bluzy z napisem: Śmierć wrogom ojczyzny i nawołują do wieszania na drzewach przeciwników politycznych. Gdy język nienawiści jest coraz bardziej oswajany, prędzej czy później może to prowadzić do przemocy i rozlewu krwi. 2 lata temu ofiarą tej współczesnej kampanii nienawiści padł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Tak kończy się przekraczanie granic debaty publicznej i bezlitosne szczucie na przeciwników politycznych, odmawianie im patriotyzmu, polskości, a nawet człowieczeństwa. Trzeba wreszcie wyciągnąć wnioski ze śmierci pierwszego prezydenta wolnej Polski, tak samo jak ze śmierci prezydenta Gdańska, zanim będzie za późno. Dość już ofiar nienawiści. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Chciałem powiedzieć kilka słów odnośnie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dla przykładu podam miasto Sosnowiec, które także dostało w tym roku w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 30 mln zł.

Środki były jak najbardziej sprawiedliwe podzielone przez rząd pana Mateusza Morawieckiego, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Obchodzimy 50. rocznicę grudniowych protestów na Wybrzeżu krwawo stłumionych przez kierowaną przez komunistyczne władze Milicję Obywatelską i wojsko. Sejm podjął dzisiaj stosowną uchwałę dotyczącą tamtejszych wydarzeń. Wszystko zaczęło się 14 grudnia od pracowników stoczni im. Tak naprawdę jednak 50 lat temu nadchodziła końcówka władzy Gomułki. Stoczniowcy ruszyli pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, gdzie wywiązały się walki uliczne i zatrzymano 330 osób. Na ulice wyjechały czołgi, spłonął budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a władza zaczęła strzelać do protestujących. Członkowie komitetu strajkowego zostali brutalnie pobici. Napięta sytuacja spowodowała, że podjęto decyzję o zamknięciu stoczni. Mimo to wicepremier Kociołek, zwany później katem Trójmiasta, w telewizyjnym przemówieniu wezwał robotników, by przyszli do pracy. Ci, którzy wykonali polecenie premiera, zostali ostrzelani z karabinów maszynowych, m.in. Zbyszek Godlewski, pierwowzór tytułowego bohatera „Ballady o Janku Wiśniewskim” Krwawa pacyfikacja przyniosła 20 ofiar śmiertelnych, wieleset osób zostało rannych, 1000 osób aresztowano. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.